Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wszystkie zebrania odbędą się w sali nr 217 w budynku Senatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 252. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. W przypadku odrzucenia wniosku o odrzucenie rozstrzygniemy sprawę skierowania tego projektu ustawy do komisji. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Rząd w zeszłym roku podniósł VAT na wodę mineralną, ale uparcie twierdzi, że podatek od cukru nie jest kolejnym pretekstem do łupienia Polaków, tylko ma ograniczyć spożycie cukru, żeby Polacy byli zdrowsi. A więc ja mam pytanie: Panie premierze, jeżeli uważa pan, że ma pan prawo dyktować Polakom, jak mają żyć, żeby byli zdrowsi, to kiedy mamy się spodziewać programu: jogging+, w ramach którego zapanuje powszechne, codzienne, obowiązkowe bieganie Polaków, oczywiście z prezesem Kaczyńskim na czele peletonu, mam nadzieję, co na pewno poprawi zdrowie Polaków?

Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska, z pytaniem. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy ma piękny tytuł: o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. To 20 stron. Wszystko jest w uzasadnieniu. Tylko tu. Ale co będzie obowiązywać jako prawo? Te 20 stron. Nie tytuł, nie piękne słowa ministra zdrowia, tylko te 20 stron. Od czego? Od małpek i od napojów. Napojów zrobionych z czego? Napojów zrobionych z polskich jabłek, z polskich malin, z polskich truskawek. Dziękuję, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To standardy europejskie, o czym wczoraj mówiłam. Kraje europejskie wprowadzają te opłaty, dlatego że jest wielkie zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi. Taka choroba jak cukrzyca po prostu pogrąża.

Szanowni państwo, razem zadbajmy o zdrowie Polaków. Dziękuję, pani poseł. Proszę państwa, ja jednak bardzo proszę. Każdy z państwa ma prawo zadać pytanie, ale bardzo proszę, żeby sala jednak. Panie pośle, proszę nie dyskutować, dobrze? Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Ten podatek i przede wszystkim podatek od małpek, które w tej chwili są przyczyną tego, że młodzież coraz bardziej się rozpija, jest podatkiem po prostu słusznym.

Nie wiemy, jak to się stało, będziemy to wyjaśniać. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Janusz Cieszyński. Wysoka Izbo! Ja bym przestrzegał przed obawami przed skierowaniem tego projektu do prac w komisji, ponieważ, szanowni państwo, opłatą nie będzie objęte to, co państwa najbardziej interesuje, czyli sok z buraka. Dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 210, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystąpimy obecnie do rozstrzygnięcia sprawy skierowania projektu ustawy do komisji. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby projekt ustawy został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie tego projektu ustawy dodatkowo do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poddam pod głosowanie. Sprzeciwu nie słyszę.

Państwo doskonale słyszeliście, co przeczytałam. Dziękuję. Bardzo proszę.

No, pędzicie z tym tak, jakbyście myśleli, że od tego się pali kalorie. Pan Łukasz Schreiber wczoraj powiedział: Podatek cukrowy to niestosowna nazwa. To najwyżej jest pewnego rodzaju opłata, ale nie chodzi o podatki, żeby komuś zabrać pieniądze. Staramy się obniżać podatki na tyle, na ile to możliwe. Gratuluję. To jest tak: Podatek to nie jest podatek, tylko opłata. Nauczcie się wreszcie. Czas się nauczyć, tak? Czas się nauczyć. Poza tym to dla naszego dobra. Starają się też obniżać podatki, ale im nie wychodzi. Są strasznie nieskuteczni. Skuteczność macie zerową w obniżaniu podatków. Proszę państwa, to jest podatek cukrowy. Ja uwielbiam słodycze. Ja tę sprawę będę traktował osobiście. Dziękuję, panie pośle. Proszę.

O święta naiwności! To naprawdę co będzie obowiązywać? Jeśli rząd PiS chce zrealizować to wszystko, o czym mówi pan minister, co jest tu zawarte, chce walczyć z otyłością, to dlaczego nie zrobi tego, co podaje w uzasadnieniu? Chodzi o to, żeby one były drogie i żeby Polacy za nie więcej płacili, ale pili nadal dużo. to dlaczego opodatkowuje się napoje z polskich jabłek i truskawek, a nie opodatkowuje się cukru? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! No tak się składa, na wasze wszystkich nieszczęście, że dzień wolności gospodarczej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przypada akurat najszybciej, znacznie szybciej, o miesiąc szybciej niż pod rządami Platformy. PCK. Tak się składa, bo biorąc pod uwagę tę logikę, należałoby także wycofać się z opodatkowania. Tylko problem polega na tym, i to mówię do wszystkich miłośników wolności, że później ci wszyscy ludzie trafiają do publicznej służby zdrowi i mają być leczeni oczywiście za pieniądze wszystkich. No to jest rzeczywiście logika. Faktycznie. A te pieniądze pójdą na sport dla dzieci, do szkół, na infrastrukturę sportową. Rzeczywiście zamiast pić napoje słodzone, zachęcam do tego joggingu.

Proszę bardzo, pan poseł Marek Rutka, Lewica. Panie Premierze! W pewnej mierze ten przedstawiony projekt wygląda jak prezent dla ponadnarodowych wielkich korporacji producentów napojów kosztem rodzimych i często rodzinnych producentów z kilkudziesięcioletnią tradycją. Ustawa zawiera szereg wadliwych rozwiązań dotyczących systemu poboru opłat, w tym przepisy dające możliwość unikania opłaty przez duże sieci handlowe, zamawiające bezpośrednio u producentów napoje tzw. marek własnych. Wobec tego oczywiście zgłaszamy wniosek o to, aby to trafiło do komisji. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do komisji. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o dodatkowe skierowanie projektu ustawy zawartego w druku nr 210 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Proponuję, na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, aby Sejm wyznaczył komisji termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go w dniu dzisiejszym. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji, aby Sejm wyznaczył komisji termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający jego rozpatrzenie w dniu dzisiejszym, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 252)

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 252, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Ogłaszam 2 minuty przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe.

W takim razie bardzo proszę pana posła o zadanie pytania. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W lipcu 2019 r. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł. ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązanie ma charakter systemowy, a nie jednorazowy. Pragnę zapytać, ile osób w 2019 r. skorzystało z dodatkowego świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi za zadanie pytania. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Paweł

Wysoka Izbo! Najpierw wygłoszę komentarz nie na temat, ale myślę, że kiedy już ustawa o zapewnianiu dostępności zacznie działać z pełnym skutkiem, to ta sala będzie mieć duże kłopoty. Odpowiadając na pytanie dotyczące świadczenia 500+, chcę powiedzieć, że wszystkie organy rentowe, czyli ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej, przyjęły 672 700 wniosków o to świadczenie uzupełniające, z czego 469 275 w ZUS-ie i 201 tys. w KRUS-ie. Reszta to są liczby zupełnie nieznaczące w skali całego przedsięwzięcia. Przy tym ciekawe, że wnioski złożone przez kobiety stanowiły 63%, a przez mężczyzn 37%.

Ważne jest, że - zaraz dojdziemy do kwestii, które mogą nasuwać pytania, a nie wszyscy będą mogli je zadać - 31% tych wniosków to były wnioski, które nie wymagały dodatkowego stawania na komisji lekarskiej, ponieważ zawierały także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pozostałe wnioski, czyli 69%, tego orzeczenia nie zawierały, co oznacza, że te osoby musiały stawać na komisji, po to żeby tę niezdolność do samodzielnej egzystencji stwierdzić.

Pozostałe to są już liczby dwucyfrowe w ilościach, więc nie będę o tym opowiadał.

Jeżeli będzie to dla państwa ciekawe, to mogę też podać, jak to wyglądało w innych organach rentowych.

Jeśli chodzi o rok bieżący, w projekcie planu finansowego na 2020 r. kwota zaplanowana na wypłatę świadczenia to jest 4 miliony 540.

W zasadzie to są główne rzeczy, które (Dzwonek) chcę powiedzieć.

Świadczenia nie pobieram, ale głównie ze względów etycznych.

Ta kwota 4543 mln jest prawie 10 razy wyższa od pierwotnie zakładanej kwoty Funduszu Solidarnościowego, więc nie ma mowy o pogarszaniu sytuacji osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Sławomir Skwarek. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dodatkowe moje pytanie jest bardzo proste. Chciałbym poprosić, ponieważ bardzo często do naszych biur poselskich zgłaszają się osoby niepełnosprawne, o przypomnienie podstawowych kryteriów, jakie muszą być spełnione, żeby uzyskać świadczenie. To świadczenie, jak już to pewnie wybrzmiało z mojej poprzedniej wypowiedzi, jest adresowane do osób, które mają orzeczenie o tzw. całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przyznam, że jest to sformułowanie bardzo niefortunne, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, kiedy zajmiemy się reformą systemu orzecznictwa, takie sformułowania, które ani nie są zgodne z duchem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ani nie szanują godności osoby niepełnosprawnej, znikną. Natomiast w tej chwili to tak funkcjonuje. To jest orzeczenie, które wydają komisje ZUS-owskie lub porównywalne, czyli KRUS-owskie itd. Takich instytucji jest kilka. A więc jeżeli osoba posiada wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to ono nie jest wystarczające i trzeba je uzupełnić o takie właśnie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dziękuję bardzo panu ministrowi za udzielenie odpowiedzi. Kolejne pytanie będą zadawali państwo posłowie: Bartłomiej Sienkiewicz, Sławomir Nitras, Marek Sowa, Katarzyna Maria Piekarska i Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, w sprawie niepowoływania od 2 lat Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej - do prezesa Rady Ministrów. Na pytanie odpowie sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan Paweł Szrot. Bardzo proszę o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W maju 2018 r. wygasła kadencja jednej z najważniejszych instytucji dialogu polsko-żydowskiego i, co tu dużo mówić, jednego z filarów takiej miękkiej siły państwa polskiego, czyli Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W jej ostatnim składzie byli m.in. dyrektor instytutu Yad Vashem, dyrektor Muzeum Holocaustu, przewodniczący Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, ocaleni, wybitni przedstawiciele nauki i kultury. Nowa rada nie została przez pana premiera powołana od prawie 2 lat. Byłej przewodniczącej oraz członkom rady przedstawiciele rządu nie udzielili żadnych informacji co do jej dalszych losów. Niedawne wydarzenia wokół 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, które organizowała Fundacja Yad Vashem w Jerozolimie, ukazały absolutną bezradność polskiej dyplomacji.

Symbolem tej bezradności była nieobecność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w trakcie tych obchodów w Jerozolimie. Zabrakło tej miękkiej siły. W związku z powyższym zwracam się do pana premiera o wyjaśnienie powodów zaniechania powołania rady. Czy to zaniechanie było wynikiem zaniedbania, bałaganu urzędniczego, czy wręcz przeciwnie, stoi za tym jakiś zamysł polityczny? A jeśli tak, to jaki? Tertium non datur - albo bałagan, albo polityka, trzeciej drogi nie ma. Oczekuję wyjaśnienia, dlaczego pan premier uśmiercił jedną z najważniejszych instytucji w dziedzinie oddziaływania Polski odniesieniu do kluczowego problemu jak stosunki polsko-żydowskie i czy tym samym pan premier poczuwa się do współodpowiedzialności za kryzys wynikły wokół obchodów wyzwolenia (Dzwonek) obozu oświęcimskiego. Dziękuję bardzo. Proszę pana ministra Pawła Szrota o udzielenie odpowiedzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Chciałbym z całym naciskiem stwierdzić, że Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów i od prezesa Rady Ministrów zależy, w jakim tempie, w jakim składzie i w jakim momencie zostanie powołana. Panie Pośle! Powołanie takiej rady wymaga wielu szczegółowych, dyskretnych działań ze strony polskiego rządu, tym bardziej że rada ta, jak pan dobrze wie, składa się zarówno z komponentu krajowego, polskiego, jak i komponentu zagranicznego. Ja tutaj tego nie przesądzam - rada, owszem, mogła odegrać pewną rolę w wydarzeniach związanych z konferencją w Yad Vashem, ale absolutnie nie zgodzę się z diagnozą, którą pan poseł przedstawił z tej trybuny, że jakoby te wydarzenia miały świadczyć o rzekomej bezradności polskiego rządu. Przeciwnie, wydarzenia te i ich ostateczny wydźwięk świadczyły o sile polskiego rządu i o przemyślanych, zaplanowanych działaniach, które osiągnęły skutek. A skutkiem tego jest następujący fakt: polska narracja historyczna, korzystna dla polskiego narodu, dla Rzeczypospolitej, dla władz Polskiego Państwa Podziemnego, dla żołnierzy polskiego podziemia, przebiła się zarówno w narracji.

Również w opiniach i ocenach większości przedstawicieli środowisk żydowskich zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. I to jest sukces polskiej dyplomacji.

Nieobecność pana prezydenta była efektem przemyślanych działań.

I powtarzam: chodzi tutaj o wiele szczegółowych uzgodnień, działań, częściowo zakulisowych, chodzi tutaj o kuchnię dyplomatyczną. I tu chciałbym powiedzieć, że istnieją pewne okoliczności, które pozwalają mieć nadzieję, że ta rada w nieodległym czasie będzie powołana. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Sławomir Nitras. Bardzo proszę. Proszę więc powiedzieć, jakie są plany wasze, jaka ma być ta korekta, jakie cele macie zamiar osiągnąć i jakimi metodami.

Wy w ogóle nie rozumiecie chyba słów „miękka polityka”, wy rozumiecie słowa „młotek, przecinak, kombinerki”, a nie coś, co jest elementarnie wysublimowane. Przecież tu nie chodzi tylko o radę. To się wpisuje w pewien ciąg relacji polsko-żydowskich. Przecież pan mówi, że prace trwają i że może powołać, kiedy chce. Tak samo z dyrektorem muzeum Polin - też może powołać, kiedy chce, tylko go nie ma. Wygrał konkurs i go nie ma. Przecież to są jawnie antyżydowskie działania. To samo dotyczy IPN-u. Przecież pan prof. Kurtyka w roku 2009 podpisał umowę o współpracy IPN-u. z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Boicie się czegoś? Zamykacie się na świat? Żeby zamknąć, zabetonować? To jest pytanie o to, jakie efekty chcecie osiągnąć. Pan minister odniesie się. Proszę bardzo. Panie Pośle! Usłyszałem przed chwilą, że w mojej wypowiedzi przejawia się „straszna antyżydowska fobia”

Jest przeciwnie - wiele tutaj mówiłem o efektach, które rząd polski uzyskał, prowadząc swoją politykę w przyjętych przez siebie formie i trybie. Te efekty są takie, że wielka część środowisk żydowskich zarówno w Izraelu, w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych i w innych częściach świata popiera narrację historyczną, polegającą na prawdzie oczywiście, którą rząd polski wielokrotnie prezentował na różnych forach. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Kolejne pytanie dotyczy likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. Skierowane jest ono do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a pytanie to będzie zadawał pan poseł Marek Rutka z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Ministrze! Decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po 64 latach funkcjonowania z dniem 1 kwietnia br. Urząd Morski w Słupsku ulegnie likwidacji. 1 kwietnia dla ok. 300 pracowników urzędu morskiego nie będzie jednak do śmiechu.

Powyższa decyzja zapadła wbrew stanowisku władz samorządowych, m.in. prezydenta Słupska czy burmistrza Ustki, wbrew pracownikom urzędu morskiego, pomimo protestów zakładowej organizacji związkowej „Solidarność” Opinia związkowców została całkowicie zlekceważona, podobnie jak opinia ogólnopolskiego związku oficerów i marynarzy. W końcu jest ona wbrew wcześniejszemu stanowisku samego rządu i stanowisku pana premiera Morawieckiego, który jeszcze kilka lat temu zapewniał: To jest potrzebne, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać z małych miejscowości i wiosek, w szczególności za granicę. Chcemy, żeby tutaj zostali i pracowali dla Polski. Chciałbym przytoczyć fragment pisma, które Paweł Szrot, obecny zresztą dzisiaj na sali, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierował do pani Anny Moskwy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Uwagę zwraca brak szczegółowego uzasadnienia projektowanego zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie, iż zmiana przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego realizowania zadań administracji morskiej, wydaje się niewystarczające w odniesieniu do planowanej poważnej reorganizacji struktury terenowej administracji państwowej. Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytania: Czy w wyniku likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku którakolwiek z obecnie zatrudnionych osób straci pracę? Drugie: Czy likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku wpłynie negatywnie na rozwój gospodarczy regionu i czy ministerstwo dokonało stosownych analiz sytuacji? Co stanowiło społeczno-gospodarczą podstawę decyzji o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku? Wreszcie: Czym podyktowane jest niedawne zatrudnienie w Urzędzie Morskim w Gdyni na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw inspekcji morskiej pana Macieja Jeleniewskiego, osoby, która w listopadzie ub.r. została odwołana ze stanowiska wicedyrektora do spraw inspekcji morskiej w Słupsku? A była to osoba, która zajmowała się inwestycjami, które w raporcie NIK bardzo ostro skrytykował. A ten raport, przypomnę, był jedną z podstaw zlikwidowania Urzędu Morskiego w Słupsku. I ostatnie: Czy decyzja ministerstwa została skonsultowana ze związkami zawodowymi, przedstawicielami organizacji społecznych i samorządem terytorialnym? Proszę jednocześnie o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli pani Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie pośle, rzeczywiście od 1 kwietnia Urząd Morski w Słupsku będzie funkcjonował w innym wymiarze, w innej strukturze organizacyjnej. Tak jak wielokrotnie odpisywaliśmy, znajduje się to też w uzasadnieniu tej decyzji, motywacją były powody efektywnościowe i ekonomika wydatków środków publicznych, przede wszystkim w tej części administracyjnej dotyczącej dużych przedsięwzięć, dużych przetargów i dużych inwestycji. W naszej ocenie realizacja tych dużych i niezwykle ważnych zadań, które stoją nie tylko przed tym urzędem morskim, ale w ogóle przed administracją morską, będzie możliwa, lepsza w dwóch strukturach połączonych stricte ze strukturą administracyjną w podziale na województwo pomorskie i zachodniopomorskie. Jednocześnie też bezpodstawne jest straszenie pracowników, bo w dużej mierze te obawy i niepokoje, które się pojawiły lokalnie, wynikały tak naprawdę z działań politycznych i pobudek politycznych, jeżeli chodzi o wywołanie tych niepokojów. One nie były pierwotne, tylko wtórne. Są absolutnie nieuzasadnione. Nikt z pracowników, i to wielokrotnie podkreślaliśmy i dzisiaj podkreślamy, nie straci pracy. Zmiana tej struktury organizacyjnej absolutnie nie oznacza, że rezygnujemy z inwestycji na tym terenie, tylko wręcz przeciwnie, chcemy je realizować lepiej, szybciej, efektywniej w wymiarze tych dużych struktur organizacyjnych. On się nam sprawdził, wpłynął pozytywnie. Udało nam się dokonać też podwyżek wynagrodzeń, szczególnie w tych kluczowych pionach, a więc ta optymalizacja też tutaj jest z tym związana. Absolutnie nie wiązałabym drugiej części wypowiedzi pana posła z jakimś motywem osobistym, z przenoszeniem pracownika czy dyrektora.

Pan dyrektor spełnia wszystkie wymagania. Decyzja została podjęta na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń, kompetencji i wykształcenia.

W takim razie. Pani minister powiedziała coś takiego: urząd morski będzie funkcjonował w innej formie. Czy to oznacza, że będzie funkcjonował?

Najpierw został on zdymisjonowany, a teraz awansował, co więcej, na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku jest informacja o tym, że nadal jest wicedyrektorem do spraw inspekcji morskiej w Słupsku. Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni jest informacja, z jego zdjęciem, że jest zastępcą dyrektora do spraw inspekcji morskiej. Czy pracuje on w dwóch miejscach jednocześnie? Nie wydaje mi się, żeby Izba się tym zajmowała.

Nikt nie straci pracy. Moje pytanie brzmiało: Czy pan Maciej Jeleniewski pracuje w dwóch miejscach jednocześnie?

Odpowiedzi udzieli pan Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Czekamy na ministra.

Pani Minister! Taka sytuacja jest dla nas zagrożeniem, bowiem może przyczynić się do wystąpienia ewentualnej suszy, której skutki będą oddziaływać na nas najsilniej od kilkudziesięciu lat. Pierwszą myślą, która w takim wypadku mogłaby być jednym z pomocniczych narzędzi, jest poziom retencjonowanej wody w Polsce. Wskaźnik ten wynosi 6,5% i niewątpliwie wymaga podwyższenia. Niezbędne wydaje się również przygotowanie programów indywidualnych, jak i zbiorowych, które mogłyby przeciwdziałać ewentualnej suszy. W związku z powyższym pragnę zapytać panią minister i prosić o udzielenie odpowiedzi, jakie działania planuje podjąć ministerstwo, by zmniejszyć lub też zminimalizować ryzyko wystąpienia w Polsce suszy spowodowanej niską ilością opadów atmosferycznych. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Pośle!

Pan poseł wspomniał, że powódź też się pojawia, to jest oczywiście prawda. Natomiast to, co jest współczesnym problemem, to gwałtowność tych zjawisk, zarówno w wymiarze suszy, jak i w wymiarze powodzi.

Oczywiście jest prawdą, że mamy w Polsce mało wody.

Na poziomie ministerstwa rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmuje się mikroretencją, czyli szeroko pojętymi systemami nawadniania poprzez małe zbiorniki i studnie głębinowe.

To jest na poziomie mikroretencji. Działania na poziomie małej, średniej i dużej retencji są prowadzone przez Wody Polskie i nasze ministerstwo. Może przedstawię je w takim wymiarze, co jest robione i co będzie robione w dalekosiężnych prognozowaniach. Te dwa programy chcemy zintegrować w tym roku w jeden duży program. One są prowadzone równolegle przez nas i przez Wody Polskie. To, co w tym programie jest i będzie robione, to wielotorowe działania. Prowadzimy też projekty remontów śluz i jazów, żeby zwiększyć ilość wody, i to jest coś, co jest i będzie robione w tych wszystkich programach. Jednocześnie jest tam cały pakiet zalesienia, tworzenia zadrzewień, przebudowy drzewostanów, także odtwarzanie stawów hodowlanych, wdrożenie miejskich planów adaptacji i to wszystko, co jest związane z retencją w miastach - to przede wszystkim Ministerstwo Klimatu. Małe zbiorniki i duże zbiorniki.

Oczywiście działania mikroretencji są bardzo ważne, natomiast bez dużej retencji, budowy dużych wielofunkcyjnych zbiorników nie będziemy w stanie tego osiągnąć. My też w gospodarce wodnej zastosowaliśmy, stosujemy podejście zintegrowane, czyli nie patrzymy na inwestycje w gospodarce wodnej przez pryzmat czy to wyłącznie powodzi, czy to suszy, czy to funkcji transportowej, tylko pod kątem integracji tych wszystkich celów, tak żeby jedna inwestycja, np. Wilkówka, Jamno czy inne słynne przeprowadzone inwestycje w Polsce, tak naprawdę nie zaburzyła bilansu wodnego, tylko służyła optymalizacji tych zasobów i jednocześnie chroniła nas przed powodzią i suszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe pan poseł za chwilę zada, tak? W swoim dodatkowym pytaniu chciałbym prosić o informację, czy ministerstwo będzie starało się realizować przedstawione rozwiązania z wykorzystaniem środków zewnętrznych, np. pochodzących z Unii Europejskiej, czy takie środki są, lub też czy w pierwszej kolejności będzie się wskazywać Unii na zwiększone potrzeby w tym zakresie i konieczność zwiększenia nakładów finansowych. Dziękuję.

Jeżeli chodzi o nową perspektywę, to oczywiście ona jeszcze nie jest w na tyle dojrzałym kształcie, żeby powiedzieć konkretnie, co będzie możliwe.

Oczywiście stykamy sią na poziomie Unii Europejskiej z dużą dyskusją dotyczącą tego, że to jest ingerencja w hydromorfologię rzek, również przy projektach przeciwpowodziowych, co oczywiście wydaje się niezrozumiałe, natomiast mamy ambicję, żeby jak najwięcej środków na ten obszar, na szeroko pojętą gospodarkę wodną, bez rozróżniania na jaką funkcję, w tej nowej perspektywie się znalazło.

Dosyć śmiała teza, panie pośle. Ono było takie trochę. Nie znam. Nie?

Natomiast były takie inwestycje, stąd mówiłam o podejściu zintegrowanym przy inwestycjach w gospodarkę wodą, żeby rzeczywiście nie patrzeć na źródło finansowania - skoro Unia np. finansuje inwestycje przeciwpowodziowe, to realizujemy inwestycje przeciwpowodziowe i nie patrzymy na pozostałe aspekty. Dziękuję bardzo, pani minister. Ponieważ dotarł do nas już pan minister Adam Gawęda, panowie posłowie Krzysztof Gadowski, Tomasz Piotr Nowak, Wojciech Saługa i Marek Sowa mogą zadać swoje pytanie. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jeszcze nie tak dawno na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości widniało hasło, że bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte będzie na węglu pochodzącym z Polski. W 2015 r. na rynku w Rudzie Śląskiej prezes, przyszły minister energii i przyszły wiceminister energii z Rudy Śląskiej krzyczeli: dość węgla z Rosji, skończymy z tym! Jak to wyglądało w przeciągu ostatnich lat?

Większość tego węgla pochodzi z Rosji, prawie 70 mln t. W 2018 r. było to prawie 14 mln t. To prawie 50% tego, co produkuje Polska Grupa Górnicza, największa polska grupa górnicza zatrudniająca 42 tys. osób. Okazuje się, że to nie wszystko.

Jak podają związkowcy, ponoć jedna z grup energetycznych, która kapitałowo jest zaangażowana w Polską Grupę Górniczą, sprowadza węgiel, sprowadziła go prawie 5 mln t, tyle ile leży pod kopalniami. Jak donoszą ostatnio media, spółki z udziałem Skarbu Państwa nie tylko zajmują się importem, one zajmują się też dystrybucją. Przez 4 lata (Dzwonek) coraz więcej węgla importujemy do Polski. Dziwi, że rząd nie potrafi sobie poradzić nawet ze spółkami Skarbu Państwa, które sprowadzają ten węgiel. Panie Ministrze! Dzisiaj kierujemy do pana pytania. Jakie spółki Skarbu Państwa sprowadziły do Polski przez ostatnie 4 lata węgiel? Ile tego węgla sprowadziły? Gdzie ten węgiel trafił? Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy z ust przedstawicieli rządu, że w ogóle spółki Skarbu Państwa nie sprowadzają węgla, ale kilka dni temu minister aktywów państwowych wyraźnie powiedział, że spółki Skarbu Państwa nie będą już importować węgla. Jaka jest prawda, panie ministrze? Żądamy tej informacji. Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie!

Wszyscy, którzy zajmują się procesami i zarządzaniem w sektorze górniczym, w innych sektorach również, ale w tym szczególnie, wiedzą, że procesy inwestycyjne, procesy udostępnienia nowych pól eksploatacyjnych, ścian wysokowydajnych to są procesy inwestycyjne, które przynoszą efekty w perspektywie 2, 3, a czasami nawet i 4 lat.

Rok do roku nastąpiło zmniejszenie. Głównym kierunkiem, z którego importowany jest węgiel, pozostaje Federacja Rosyjska, z której w 2019 r. zaimportowano łącznie 10,8 mln t, co odpowiada spadkowi importu rok do roku o 2,5 mln t z kierunku rosyjskiego, z Federacji Rosyjskiej. Spółki Skarbu Państwa lub spółki, w których Skarb Państwa posiada udziały, sprowadzały w 2019 r. węgiel również do Polski ze względu na ograniczenia wynikające z obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, a także dotyczące przepisów o statystyce publicznej. Informacje o imporcie węgla mogą być udostępniane wyłącznie w zagregowanej formie. To też dość mocno chcę podkreślić. Łączna ilość węgla energetycznego zaimportowanego do Polski przez spółki Skarbu Państwa lub spółki, w których Skarb Państwa posiada udziały, wyniosła nieco powyżej 4 mln t. Przeszło 9 mln t węgla energetycznego zaimportowano do Polski poprzez prywatne podmioty i są to decyzje zarządcze tychże właśnie podmiotów prywatnych. Według informacji statystycznych opracowanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej do energetyki zawodowej i przemysłowej trafia ok. 17% importu, czyli ok. 2,8 mln t. Węgiel brunatny nie jest importowany do energetyki. W ubiegłym roku do energetyki zawodowej i przemysłowej z polskich kopalń trafiło 97% węgla kamiennego i brunatnego. To jest bardzo ważna informacja, bo to wskazuje, że rzeczywiście główny wolumen węgla kierowany do energetyki zawodowej pochodzi właśnie z naszych kopalń, ze spółek Skarbu Państwa. Należy zaznaczyć, iż w poprzednich latach nastąpił spadek wydobycia rodzimego węgla. To właśnie było powodem tego, że znacząca część tego surowca musiała być zakontraktowana i zaimportowana z zewnątrz. Warto też wskazać na pewne trendy, które pokazują, że w Polsce jest nadal duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny, głównie w gospodarstwach domowych jest on wykorzystywany. Wiemy doskonale, że nowe kotły piątej klasy spełniające te parametry są stosowane w wielu gospodarstwach domowych. W 2017 r., po ustabilizowaniu sytuacji w branży, można było rozpocząć procesy inwestycyjne, które również są skierowane w stronę tego, żeby poprawiać jakość węgla, kierować ten surowiec w sposób usystematyzowany również do tych odbiorców, którzy wykorzystują kotły wysokiej sprawności (Dzwonek) i o dobrych parametrach, które nie powodują zanieczyszczenia niską emisją. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Wojciech Saługa. Dziękuję, panie marszałku. Panie Ministrze! Premier waszego rządu. i ówczesny minister właśnie z Rudy Śląskiej wielokrotnie na Śląsku mówili, że górnictwo wstało z kolan, że już wszystkie problemy - jak tylko wy doszliście do władzy - zostaną rozwiązane, a odpowiedzialne za zły stan górnictwa były rządy Ewy Kopacz i poprzednie. Ale tym wystąpieniem potwierdza pan to, że górnictwo jest dalej na kolanach, a tamte słowa to były puste słowa. Dlaczego, panie ministrze, mimo zapotrzebowania na węgiel spada jego wydobycie? Dlaczego mimo tysiąca ton na zwałach wciąż sprowadzamy węgiel z zagranicy? Dlaczego np. kopalnie Grupy Tauron nie są w stanie dostarczyć węgla do własnych elektrowni? Jak pan wytłumaczy to, że właśnie spółka Tauron Wydobycie stoi na skraju bankructwa, mimo że jest dostawcą węgla do państwowych elektrowni? Importujemy smog ze wschodu, a my dopłacamy do likwidacji kopalń. Tak wstajemy z kolan? Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytanie.

Wysoka Izbo! W moim wystąpieniu dotykałem faktów.

Otóż w roku 2015, kiedy rządziły w Polsce Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, wszystkie spółki, nie jedna, nie dwie, były na skraju upadłości. Groziła im likwidacja i procesy upadłościowe. My, rząd Prawa i Sprawiedliwości, brałem wtedy udział w audycie otwierającym, to był początek roku 2016, doprowadziliśmy do tego, że uniknęliśmy procesu upadłościowego. Wszystkie spółki przeszły ten bardzo trudny okres obronną ręką - przepraszam za ten kolokwializm, ale tak właśnie się działo - i doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj one są stabilne finansowo.

Ani jeden z tego typu instrumentów ochronnych finansowych nie został wprowadzony. To była nasza odwaga, że zaudytowaliśmy wszystkie spółki, pokazaliśmy faktyczny stan, fatalny stan polskiego górnictwa, i przeprowadziliśmy proces naprawczy. Rzeczywiście ten proces sprawił, że żadna spółka nie została zlikwidowana i utrzymujemy miejsca pracy. To nie jest łatwe, bo w procesach funkcjonowania górnictwa trzeba szukać najlepszych rozwiązań, również tych, które nie oddziałują w znaczący sposób na powierzchnię, aby mieszkańcom, którzy mieszkają na terenach górniczych, można było również zapewnić normalne, godziwe mieszkanie, rozwój i realizację biznesowych kierunków. Tauron Wydobycie przygotował proces naprawczy i realizuje plan naprawczy. Rzeczywiście jest to spółka bardzo trudna, bo wcześniej bardzo mocno niedokapitalizowana. To nie jest łatwy ani szybki proces. Każdy, kto jest związany z branżą górniczą, wie, że procesy budowy szybu, budowy wyrobisk głównych, przekopów, udostępniających wyrobisk, to procesy wieloletnie, w tej perspektywie co najmniej 6-, 7-letnie. Potencjał wydobywczy coraz to lepiej jest dostosowany do potrzeb energetyki zawodowej i naszego rynku. To są główne nasze zadania, a to najważniejsze to utrzymanie miejsc pracy i stabilność wszystkich spółek i kopalń. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zadadzą państwo posłowie Michał Szczerba i Monika Rosa. Odpowie na nie pani Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Sprawa, którą chcemy dzisiaj poruszyć, jest absolutnie pilna i ważna. Chodzi o dramatyczną sytuację oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Mianowicie, Wysoka Izbo, nie przybywa ośrodków oferujących kompetentną pomoc terapeutyczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Przybywa za to prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Powoduje to, Wysoka Izbo, że do lekarzy psychiatrów kierowane są w trybie pilnym osoby niewymagające tego typu pomocy. Skutkuje to również tym, że osoby z nasilonymi objawami i ryzykiem samobójczym lub zachowaniami agresywnymi oczekują miesiącami na wizytę i leczenie. Otrzymaliśmy ostatnie dane, z których wynika, że w Polsce było 98 samobójstw wśród dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic. To sytuacja zatrważająca. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę samobójstw. Szanowni Państwo! Te dramatyczne warunki leczenia, katastrofalną sytuację psychiatrii dziecięcej przedstawił ostatnio reportaż Onetu - „Miłość w czasach zarazy” Zauważył także tę sytuację Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w zeszłym roku przekazała pierwsze pieniądze na wsparcie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - ok. 3 mln zł. Udało się kupić m.in. 800 łóżek. Ale są to, pani minister, działania niewystarczające.

Na jakim etapie są prace nad reformą psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży? To jest absolutnie ważny temat, którym powinniśmy się zająć. Dziękuję. Proszę teraz panią minister o udzielenie odpowiedzi. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Ja już bodajże miesiąc temu informowałam państwa o działaniach, jakie podejmuje minister zdrowia w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzeczywiście obecny stan trwał od wielu lat, bo od kilkunastu lat nie podejmowano żadnych działań mających na celu dostosowanie obecnego modelu opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży do obowiązujących standardów światowych czy też europejskich. Dlatego też my już od 2018 r. podjęliśmy konkretne działania, aby zmienić ten system, aby go uczynić bardziej przyjaznym, a przede wszystkim aby dzieci i młodzież, u których pojawiają się pierwsze symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego, mieli udzieloną pomoc jak najszybciej, w warunkach przyjaznych, czyli najlepiej w środowisku, w którym żyją, łącznie ze środowiskiem szkolnym, aby ta pomoc była dostarczona w odpowiednim momencie i odpowiedniej jakości. Jeżeli chodzi o aktualny stan, to mamy w kraju 34 oddziały psychiatryczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które udzielają świadczeń w trybie całodobowym. Ale oprócz tego typu instytucji wsparcia udzielają również w zakresie zdrowia psychicznego dzienne oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, których mamy zakontraktowanych 38. Świadczenia psychologiczne udzielane są w 127 placówkach, a świadczenia psychiatryczne, ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży w 166. Należy podkreślić, że z roku na rok wzrastają nakłady na ochronę zdrowia. W stosunku do 2018 r. jest wzrost nakładów na ten rodzaj świadczeń o prawie 30%, czyli przeznaczamy coraz większą kwotę na te świadczenia. Oczywiście mamy świadomość, że dosypywanie do systemu pieniędzy bez zmiany systemu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dlatego też informowałam państwa, że przygotowaliśmy konkretne zmiany oparte na standardach światowych, które pozwolą doprowadzić do tego, że dziecko w przypadku zaburzenia zdrowia psychicznego będzie miało udzieloną pomoc w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. System ten budowany jest na świadczeniach środowiskowych i ambulatoryjnych, które do tej pory nie były kontraktowane. Drugi poziom to jest poziom oddziałów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i zespoły leczenia środowiskowego. Takie usytuowanie tych podmiotów, które udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, spowoduje, że do szpitali psychiatrycznych, na oddziały zamknięte będą trafiały dzieci, u których rzeczywiście występuje stan zagrożenia życia bądź też diagnostyka nie może być wykonana w innych warunkach jak tylko w warunkach świadczenia całodobowego. Natomiast większość tych problemów będzie rozwiązywana na pierwszym i drugim poziomie. Więc, panie pośle, chcę pana poinformować, o tym zresztą już wspominałam w poprzedniej mojej wypowiedzi, że rozpoczynamy proces kontraktowania poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Rozpoczął się półtora tygodnia temu zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, że w lutym będą rozpisane pierwsze konkursy. W tej chwili w 15 województwach ogłoszone zostały konkursy na zakontraktowanie poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Łącznie określono 317 rejonów, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia chce zakontraktować takie poradnie. Środki na te poradnie zostały zabezpieczone. To są dodatkowe środki, które przeznaczamy, oprócz tych, które były w planie na zakontraktowanie świadczeń właśnie z tego pierwszego poziomu.

Chcemy, aby ten zespół współpracował ściśle z rodziną, bo tam bardzo często rozpoczynają się problemy. I dlatego minister zdrowia podjął konkretne działania, zabezpieczył środki. Proces kontraktowania się rozpoczął i mamy nadzieję, że pierwsze tego typu poradnie wystartują już od 1 kwietnia i że do końca roku ta mapa poradni na terenie naszego kraju będzie sukcesywnie model, który zbudowaliśmy, który wdrażamy, który będzie finansowany, bo jest zabezpieczenie, jest oparty na standardach światowych, ale również (Dzwonek) na doświadczeniach pozyskanych w wyniku pilotażu realizowanego w kilku ośrodkach w kraju.

Dziękuję bardzo, pani minister. Dodatkowe pytanie zada pani poseł Monika Rosa. Panie Marszałku! Pani Minister! Pierwsze interpelacje dotyczące psychiatrii dziecięcej zostały wysłane do państwa ponad rok temu.

Ilu specjalistów psychiatrii dziecięcej obecnie pracuje w Polsce z dziećmi?

70% z nich ma myśli samobójcze, 70% ma depresję i problemy psychiczne. Nie spotykają się oni ze wsparciem ze strony psychologów szkolnych, o którym pani mówiła. Dziękuję bardzo. Proszę, pani minister. Wysoka Izbo! Jak państwu już mówiłam, te zmiany, które wprowadzamy w tej chwili - bo one wchodzą już w życie, to są konkretne działania - musiały być dogłębnie przemyślane. Zbieraliśmy informacje co do różnych modeli, które stosowane są w różnych krajach, i dzięki temu udało nam się stworzyć model, który jest zgodny ze standardami światowymi i najbardziej przyjazny dzieciom. W ubiegłym roku, bo pani pytała też o kadry, uregulowaliśmy kwestię kształcenia psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Określiliśmy też zasady zdobywania tych uprawnień. Jeżeli chodzi o specjalistów psychiatrii, obecnie w kraju mamy 440 specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, ale chcę podkreślić, że ten nowy model budowany jest w oparciu o psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Chcemy, aby dziecko miało pierwszy kontakt z psychologiem i psychoterapeutą, aby nie było stygmatyzowane, że leczy się w oddziale psychiatrycznym, że leczy się w poradni psychiatrycznej. Jeżeli ten zespół, o którym mówimy, zdiagnozuje potrzebę kontaktu z lekarzem, to dziecko natychmiast zostanie przekazane do lekarza.

Państwo wspominacie o problemie samobójstw. Wiele różnych czynników powoduje, że te zaburzenia są coraz częstsze. Oczywiście te poradnie mają stanowić bardzo istotną rolę i wyłapywać pierwsze symptomy depresji, tych zaburzeń, o których pani poseł mówiła. Również, co warto zaznaczyć, w „Narodowym programie zdrowia” mamy priorytety określone w ramach, w których realizuje się zadania z zakresu zdrowia psychicznego. W tym roku modelujemy „Narodowy pogram zdrowia”, gdzie szczególnie kładziemy nacisk na profilaktykę samobójstw i wspieranie dzieci w trudnych sytuacjach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli chodzi o wycenę świadczeń, została zwiększona wycena świadczeń. W tej chwili są dodatkowe środki.

Oczywiście potrzebujemy dobrej współpracy z samorządami.

Dziękuję bardzo, pani minister. Kolejne pytanie zadadzą panowie posłowie Grzegorz Lorek i Marek Polak. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Koronawirus jest kolejnym niezwykle niebezpiecznym wirusem, który powoduje coraz więcej zachorowań, szczególnie że okres inkubacji wirusa wynosi ponad 20 dni. Pani minister, mam w tej sprawie kilka pytań. Jakie działania podejmują w tej sprawie ministerstwo zdrowia oraz sanepid? Czy dzięki nim zapewnione jest bezpieczeństwo obywateli RP? Czy jest możliwa identyfikacja DNA wirusa w polskich laboratoriach, aby skrócić proces diagnostyczny w przypadku podejrzenia zachorowania? Czy wszystkie placówki zdrowia otrzymały konkretne instrukcje, jak postępować z chorym z podejrzeniem o zakażenie tym wirusem? Czy np. mailowo NFZ czy też sanepid powiadomiły gabinety lekarskie, szczególnie lekarza rodzinnego, jak należy postępować w tym przypadku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Kilka dni temu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia wybuch epidemii koronawirusa określił mianem poważnego zagrożenia dla świata. Nie brak też opinii, że jego pojawienie się w Polsce to tylko kwestia czasu. Dlatego chciałbym zapytać, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani na ewentualne pojawienie się koronawirusa w naszym kraju. Jakie środki zapobiegawcze są obecnie podejmowane, aby temu zapobiec? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy panią minister o udzielenie odpowiedzi. Wysoka Izbo! Rzeczywiście problem występowania koronawirusa jest problemem, który jest przedmiotem analiz różnych instytucji. Chciałabym w imieniu rządu polskiego zapewnić państwa, że jesteśmy przygotowani. Na bieżąco współpracujemy z wszelkimi z agendami Światowej Organizacji Zdrowia, jak również z wszelkimi instytucjami europejskimi, które również zajmują się tym tematem. My wykonujemy to w związku z tym, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że jest to zagrożenie transgraniczne. To zobowiązuje również polski rząd do uruchomienia procedur, nie tylko tych procedur, które są określone i działają na terenie naszego kraju w przypadku zagrożenia epidemiologicznego, ale również procedur międzynarodowych. Instytucją, która została przez rząd wyznaczona do nadzoru, koordynowania prac związanych z ewentualnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jest główny inspektor sanitarny, który nadzoruje całość działań związanych z profilaktyką, ochroną polskiej ludności.

Jeżeli chodzi o aktualne dane dotyczące działań, jakie podejmujemy w naszym kraju, związanych z epidemią wywołaną koronawirusem, to aktualnie nadzorem epidemiologicznym w naszym kraju objęte są 1643 osoby, 14 osób jest objętych kwarantanną, a 48, w tym 35 osób, które wróciły Wuhan, jest obecnie hospitalizowanych. Obecnie wiemy, że w prowincji Hubei przebywa jeden Polak, który nie chce wracać do naszego kraju, natomiast służby Ministerstwa Spraw Zagranicznych mają z nim kontakt. Ambasada polska jest w kontakcie z tymi osobami. Jeżeli te osoby zechciałyby wracać do kraju, to zawsze taka pomoc będzie im udzielana.

Obecnie te testy są wykonywane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny. Te testy dostarczają nam pełnej informacji na temat ewentualnej obecności tego wirusa u osób, które mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi.

Wszystkie szpitale zostały powiadomione poprzez głównego inspektora sanitarnego o trybie postępowania. Zostały wdrożone odpowiednie procedury. Również analizujemy nasze zasoby pod względem liczby łóżek intensywnej terapii, możliwości wspomagania oddychania, aparatów ECMO. Należy pamiętać też o tym, że jest centralna baza rezerw materiałowych, w której też mamy spore zapasy na wypadek zagrożenia naszego kraju. Tak że te wszystkie kwestie są na bieżąco monitorowane. Chcę przypomnieć, że główny inspektor sanitarny wydał też odpowiednie dyspozycje, które obowiązują w miejscach przylotu pasażerów do naszego kraju. Czyli na lotniskach obowiązują procedury, zgodnie z którymi te osoby, które mogły mieć kontakt z koronawirusem, są identyfikowane, są monitorowane. Ponadto monitorujemy też zasoby leków antywirusowych, które mamy do dyspozycji. W związku z tym rząd polski ma pod kontrolą całokształt zagrożeń związanych z ewentualnym rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Mamy dokładne dane, która stacja pogotowia ratunkowego, który zespół dysponuje środkami ochrony, jakimi rodzajami środków ochrony osobistej dysponuje, po to aby w przypadku pojawienia się zagrożenia można było dysponować zespołami przygotowanymi do tego celu.

Wszystkie służby działają według określonych procedur obowiązujących w takich przypadkach.

Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Marek Polak. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Pani Minister! Niektóre międzynarodowe porty lotnicze wdrożyły procedury ochronne polegające na używaniu specjalnych skanerów mierzących temperaturę ciała każdego pasażera. Na takie procedury nie zdecydował się żaden port lotniczy w Europie, w tym także w Polsce.

Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo, pani minister. Kolejne pytanie zadają panowie posłowie Grzegorz Matusiak i Marek Wesoły, w sprawie perspektyw finansowych na odbudowę linii kolejowej Jastrzębie Zdrój - Katowice w związku z programem „Kolej+” - pytanie do ministra infrastruktury. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

To też jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców wracających m.in. do Jastrzębia z bagażami, ponieważ przewoźnik, który dokonuje transportu, nie zawsze ma możliwość zabrania bagaży. W związku z tym jest bardzo duża potrzeba, żeby kolej została uruchomiona też ze względu na to, że bardzo dużo młodych ludzi, studentów korzysta z uczelni w Katowicach i byłaby to bardzo dobra forma transportu, przede wszystkim szybka i bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi za zadanie pytania. Odpowiedzi udzieli pan Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Szanowni Państwo! Przykład Jastrzębia-Zdroju, miasta niemalże 100-tysięcznego - bo 90 tys. to prawie 100 tys., można powiedzieć - jest modelowym przykładem związanym z wykluczeniem komunikacyjnym w zakresie transportu kolejowego. Identyfikacja takiego problemu stanęła u podstaw rozpoczęcia działań zaradczych przeciwdziałających tej sytuacji, które się materializują w ramach programu „Kolej+”, który składa się z trzech komponentów, elementów: inwestycyjnego, przewozowego i przeciwdziałającego likwidacji.

Te dwa akty prawa, uchwała i ustawa, pozwolą na to, aby realizować program „Kolej+”, którego głównym założeniem jest powstrzymanie degradacji i rewitalizacja infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to program kierowany do miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, bez dostępu do transportu kolejowego, czyli Jastrzębie-Zdrój oczywiście w tym pakiecie się mieści.

Ale program, o czym jeszcze kilka słów później, będzie programem otwartym, wymagającym aktywności samorządu, więc to jest lista przykładowa, a nie zamknięty katalog. Więc to będzie program, którego realizatorem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe jako narodowy zarządca infrastruktury, a jest on kierowany do samorządu terytorialnego, który we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi będzie te działania prowadzić. Jednostki samorządowe powinny łączyć się w większe grupy, żeby wspólnie móc zafunkcjonować. W pierwszej kolejności będą dofinansowane zadania mające na celu uzupełnienie istniejącej sieci kolejowej o nowe odcinki linii kolejowych, rewitalizację istniejących linii kolejowych oraz przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych w regionach, a w drugiej kolejności - zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji w tym zakresie. Katalog otwarty, wskazany w ramach założeń, przyjęty jako taki, który stanowi pewną intencję rządową.

Istotną informacją jest to, że samorząd będzie musiał ponieść wkład w wysokości 15% kosztów inwestycji.

Z tego, co wiem, konsultacje pomiędzy samorządem a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi wstępnie już chyba trwają i są prowadzone, więc to jest też dowód na to, że prawdopodobnie tutaj spotkamy się z wnioskiem.

Upłynęło już całkiem sporo czasu, żeby dokonać przemyśleń i żeby te samorządy, które są rzeczywiście zainteresowane - jak tylko otworzy się nabór - mogły się do niego zgłaszać. Znam samorządy, które już naprawdę są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o koncepcje. Pan poseł wspomniał o kwestiach związanych z połączeniami autobusowymi - namawiam samorządy do tego, aby wziąć w tym udział i skorzystać z dofinansowania (Dzwonek) w ramach funduszu autobusowego. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Marek Wesoły. Panie Ministrze! Niejako odpowiedział pan już na moje pytanie, które chciałem zadać, rozszerzyć.

Czy będą mogły uczestniczyć w tym programie? Czy ten okres 8 lat to właśnie jest taki okres, kiedy jeszcze program będzie aktywny, otwarty? Czy samorządy, o których pan wspomniał, które jeszcze nie zdążyły z tymi wnioskami lub gdzieś tam to przegapiły i przespały, będą mogły jeszcze próbować aplikować do tego programu? Niektóre te inwestycje są dużymi inwestycjami, często przekraczającymi możliwości gmin. Musieliśmy jakiś katalog opracować, żeby potoczyła się dyskusja na temat ram finansowych.

Katalog jest otwarty. Jeśli samorządy będą zgłaszały inne propozycje - to oczywiście do naboru. Nabór odbędzie się niedługo, więc namysł powinien już się kończyć. Ważnym elementem jest to, żeby rzeczywiście samorządy różnych szczebli ze sobą współpracowały. Konfiguracja współpracy jest absolutnie dowolna. Zakładam, że i gmina, i powiat, i województwo samorządowe powinny być zainteresowane dobrym transportem zbiorowym, traktując to jako inwestycję w rozwój swojego regionu, powiatu czy małej ojczyzny. Tu współpraca musi być. Musi być deklaracja marszałka jako organizatora transportu regionalnego, że on po wykonaniu takiej inwestycji uruchomi rozkład jazdy, czyli uruchomi przejazd.

Witam państwa. Pan poseł Waldemar Andzel oraz pani poseł Ewa Malik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcieliby zadać pytanie w sprawie pozyskania funduszy na odrestaurowanie zamku w Będzinie.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie to nie tylko kopalnie i huty, ale też zamki i pałace. Na Górze Zamkowej w Będzinie nad Czarną Przemszą można podziwiać zamek z XIII w. Miejsce jest mi szczególnie bliskie, ponieważ stamtąd pochodzę. Według legendy Kazimierz Wielki, przebywając w tym miejscu, powiedział: Tu będziem wypoczywali. Stąd wzięła się nazwa miasta Będzin. I tak mała osada przerodziła się w tętniące życiem miasto.

W latach 30. XIX w. zamek przeszedł gruntowną renowację, której autorem był włoski architekt Franciszek Maria Lanci. To właśnie efekt jego pracy oraz odbudowy z lat 50. ubiegłego stulecia możemy dziś podziwiać. Zamek położony jest w samym centrum miasta, na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy, otacza go fosa oraz wysoki podwójny mur obwodowy. Z zamku rozciąga się rozległy widok na całą okolicę. Organizowane są tu zjazdy rycerskie i różne wydarzenia historyczne. We wnętrzu zamku od 1956 r. funkcjonuje Muzeum Zagłębia. Zamek jest wizytówką miasta Będzina, ale nie tylko, jest dowodem waleczności i niezależności Polaków. Dzięki średniowiecznej budowli nigdy nie zapomnimy o naszych korzeniach. Jest on również naszą dumą. Dodatkowo w Polsce zabytki podlegają ochronie prawnej. Stąd kieruję pytanie do pana ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy: Czy jest możliwe unijne dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie na zamku nad Czarną Przemszą w Będzinie? Zamek wymaga renowacji, ponieważ dalsze zniszczenia będą w znaczącym stopniu pogarszały możliwości (Dzwonek) odrestaurowania obiektu. Czy dodatkowo możemy liczyć na upiększenie miejsca wokół zamku, ewentualnie stworzenie tam nowych atrakcji? Dziękuję bardzo. Zanim oddam mikrofon panu ministrowi, to, panie pośle, mam dla pana dobrą informację. Możemy to przyspieszyć, będzie głosowanie, bo są wnioski o to, żeby dać z budżetu państwa na ten zamek. W związku z tym po prostu razem spróbujemy to zrobić i będziemy obydwaj szczęśliwi. W imieniu ministra funduszy i polityki regionalnej odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pan minister Grzegorz Puda.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie należy zaznaczyć, że Śląsk - województwo śląskie - został wskazany w krajowych dokumentach strategicznych, przede wszystkim trzeba tu powiedzieć o „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, jako obszar strategicznej interwencji polityki regionalnej. Region ten zmaga się, jak państwo doskonale wiecie, z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, stąd wymaga szczególnego zainteresowania polityki państwa prowadzonej ze szczebla krajowego i, nie da się ukryć, regionalnego. Jednym z kluczowych celów jest dążenie do zmiany profilu województwa śląskiego, mówię również o terenie Zagłębia.

Tak się składa, że województwo śląskie składa się z kilku subregionów, więc mówię w tej chwili o wszystkich ważnych z punktu widzenia kultury subregionach. Oczywiście ta zmiana profilu regionów, o której mówi „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, musi być kompleksowa. Co ważne, musi być zakorzeniona w tym, co stanowi, co jest takie - my to mówimy potocznie - śląskie, a także o potencjale dziedzictwa kulturowego. Jednym z tych najważniejszych elementów dziedzictwa są zamki i ich pozostałości, w tym wspomniany przez pana posła zamek w Będzinie. Jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej jestem wielkim zwolennikiem wsparcia zabytków, dziedzictwa kulturowego w województwie śląskim, w tym jego cennych zamków. Jednym z zadań naszego ministerstwa na rzecz wzmacniania pozycji konkurencyjnej regionów jest objęcie w ramach prowadzonej polityki rozwoju regionalnego działań adresowanych do najważniejszych obiektów zabytkowych, aby uchronić je przed dewastacją i bezpowrotnym zniszczeniem.

Dobrze by było, aby te podmioty, w których pieczy znajdują się takie zabytki jak zamek w Będzinie, dysponowały długoterminowym planem rozwoju zabytku, aby mógł on pełnić rolę czynnej i znaczącej w regionie instytucji kultury. W ten sposób ratujemy nie tylko zabytek, ale jesteśmy w stanie także wspierać jego nowe funkcje, wspierać turystykę i szeroko rozumianą kulturę przez duże K. Osobiście uważam, że istotne jest łączenie takich zabytków w tematyczne szlaki historyczno-kulturowe, dzięki czemu te szlaki będą mogły wzmacniać atrakcyjność całego regionu. Ważne jest również łączenie takich miejsc w szlaki edukacyjne, które będą następnym pokoleniom, głównie następnym pokoleniom, pokazywały, jak istotna jest rola historii w tym, co robimy dzisiaj. Będzin uzyskała unijne dofinansowanie w kwocie 14 mln zł z regionalnego programu województwa śląskiego na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”

Samo województwo śląskie, z czego osobiście jestem dumny, pozyskało prawie 380 mln zł unijnego wsparcia dla dziedzictwa kultury i instytucji kultury. Wśród inwestycji tego regionu można podać przykład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach bądź remont budynku kościoła Świętej Trójcy w Bytomiu. Odpowiadając na drugą część pytania dotyczącą otoczenia obiektów zabytkowych, należy podkreślić, że możliwość takiego wsparcia jest bardzo ważna i uwzględniona w trwających pracach nad zakresem wsparcia przyszłych programów operacyjnych. W obecnej edycji funduszy europejskich projekty związane z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zabytków mogły być realizowane przez odrębne programy. Podobny zakres wsparcia chcielibyśmy utrzymać w kolejnej perspektywie, w kolejnym programowaniu na lata 2021–2027.

Jeżeli pan poseł będzie miał więcej pytań dotyczących tego typu obiektów czy w Zagłębiu, czy na Śląsku, czy w całym województwie śląskim, jesteśmy oczywiście do dyspozycji państwa, pana posła, państwa posłów. Chętnie będziemy udzielać informacji. Czekamy na to, jak w nowej perspektywie będziemy mogli korzystać ze środków unijnych. Naszym zdaniem kultura to nie tylko wydatek, ale przede wszystkim kultura to duża inwestycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Bardzo chciałem panu ministrowi podziękować za odpowiedź i rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że dba o zabytki, w tym także właśnie o ten niezwykle ważny i bliski mojemu sercu zamek średniowieczny w Będzinie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wracamy do pytania nr 5. Panie poseł Lidia Burzyńska i Joanna Borowiak oraz Barbara Bartuś z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałyby zadać pytanie w sprawie funkcjonowania systemu e-recepta - do ministra zdrowia. W imieniu ministerstwa będzie odpowiadał sekretarz stanu pan minister Szczurek. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani Minister! Wysoka Izbo!

Dzisiaj można użyć stwierdzenia, że jest to już przeszłość, ponieważ dzięki możliwości zastosowania e-recepty pacjent w celu kontynuacji leczenia po prostu wykonuje telefon i otrzymuje czterocyfrowy kod, jak również udaje się do apteki i tylko znajomość PESEL-u pacjenta umożliwia mu wykupienie recepty. E-recepta zostanie dostarczona bezpośrednio pocztą elektroniczną. Moje pytanie jest, pani minister, następujące: Jak wygląda wdrażanie i praktyczne funkcjonowanie e-recepty? To po pierwsze. Dziękuję. Jeszcze raz panią serdecznie przepraszam, ale pomyliły mi się kartki, bo miał być pan Sławomir Gadomski, minister, ale. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Troszeczkę przeszkadzacie państwo z Platformy. Panie pośle, mam uprzejmą prośbę o to, żeby pan nie przeszkadzał pani minister. Proszę bardzo.

W pierwszej kolejności podłączane były apteki, a później podmioty lecznicze. Praktycznie w 2018 r. zakończył się proces podłączania wszystkich aptek do platformy P1, czyli wszystkie apteki już były gotowe do przyjmowania i realizowania recept.

Natomiast pozostałe recepty są już realizowane w formie elektronicznej.

Tak że system działa. Oczywiście, w przypadkach awarii systemu, tak jak powiedziałam, istnieje możliwość wystawienia papierowej recepty i zrealizowania jej na dotychczasowych zasadach.

Chcę podkreślić, że nie jest wymagane posiadanie telefonu komórkowego. Pacjenci mogą otrzymywać e-receptę w wybranej przez siebie formie, m.in. mogą otrzymać jako SMS na telefon komórkowy, e-mail na wskazany adres skrzynki mailowej, ale mogą też otrzymać wydruk informacyjny od lekarza, w przypadku gdy nie dysponują takimi możliwościami. W tym wydruku jest podany numer PESEL, kod, może też być informacja na temat stosowania tego leku. Tak że osoby, które nie posiadają tych urządzeń, absolutnie nie są pozbawione możliwości realizacji e-recepty, wręcz odwrotnie. Chciałabym podkreślić, że realizujemy cykliczne szkolenia dla seniorów, które mają umożliwić korzystanie m.in. z tych kanałów elektronicznych w takim sposób aby nie trzeba było drukować nawet tych druków informacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani minister. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister, muszę rozpocząć od podziękowań, wielkich podziękowań, bo jest to duży przełom, to jest duże ułatwienie dla pacjentów, którzy biorą stale leki - szczególnie właśnie dla takich pacjentów. Nie muszą już zapisywać się do lekarza, stać w kolejce, nie zajmują tej kolejki. Naprawdę to jest rozwiązanie przełomowe. Myślę, że dzięki temu te kolejki znacząco zostaną zmniejszone, bo będzie już łatwo kolejną receptę na lek, który się bierze czasem latami, uzyskać. Ale mam też pytanie.

Myślę, że to też by było bardzo ważne i bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pani minister, może to panią zaskoczy, ale przyłączam się do podziękowań, gdyż też jestem pacjentem i korzystam. Proszę bardzo. Ja oczywiście te podziękowania od państwa, przede wszystkim od pana marszałka, przekażę panu ministrowi prof. Łukaszowi Szumowskiemu, gdyż on wyznacza główne trendy i kierunki działania resortu w zakresie ochrony zdrowia. Szanowna pani poseł, jeżeli chodzi o te ułatwienia, oczywiście to są duże ułatwienia nie tylko dla seniorów, niemniej chciałabym podkreślić jedno: w przypadku teleporady, o której pani poseł mówiła, rzeczywiście jest to możliwe. Większość pacjentów korzysta jednak osobiście z porady lekarza. System ochrony zdrowia, tak jak powiedziałam na początku, wymaga ustawicznej pracy, jeżeli chodzi o ucyfrowienie. My w tej chwili w bazie danych mamy sporo danych dotyczących realizowanych procedur na rzecz konkretnych pacjentów, natomiast jeszcze często te systemy są niespójne, wiele podmiotów leczniczych na własną rękę informatyzowało swoje obszary i w związku z tym należy podejmować działania, które mają na celu uspójnienie tych wszystkich systemów.

To pozwoli nam zebrać, zgromadzić wszelkie dane na temat stanu zdrowia pacjenta, jak również przyjmowanych leków. Do tej pory zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci, korzystając z porady np. neurologa, reumatologa, diabetologa czy innego specjalisty, otrzymują różnego rodzaju recepty i realizują je w różnych aptekach. Nie ma kontroli nad polipragmazją, a bardzo często właśnie takie zjawisko występuje.

Oczywiście jest to też taki system kontroli, jeżeli chodzi o leki wypisywane i ordynowane dla konkretnego pacjenta. Co do rozszerzenia listy leków 75+, czyli bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia, na pewno jednym z elementów, które blokowały możliwość wystawiania tych recept przez innych specjalistów, był właśnie ten niedostatek elektroniczny. Po wprowadzeniu pełnego systemu na pewno będziemy rozważać taką możliwość po to, żeby pacjenci nie musieli po receptę przychodzić ponownie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Całość opieki nad pacjentem powinien sprawować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale na pewno będziemy rozważać możliwość rozszerzenia. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, to pytanie kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie działań rządu w związku z lawinowo rosnącymi cenami i kosztami utrzymania polskich rodzin, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Marzenę Okła-Drewnowicz. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Ja wiem, że już zaczęło boleć. Bo mimo że są obiektywne przesłanki tego, że drożyzna może być, to jednak rząd jest od tego, żeby wprowadzać takie systemy i takie mechanizmy, żeby ta drożyzna nie dotykała tak bardzo polskich rodzin, szczególnie tych najsłabszych. Na początek może kilka przykładów. Coraz droższe mięso. Oczywiście mam na myśli wieprzowinę.

Otóż wtedy kiedy docierał on do centralnej Polski, wasz minister chciał budować zapory na granicach. Stąd wiemy, dlaczego dzisiaj schabowy jest kilka razy droższy niż jeszcze kilka lat temu. Mało tego. Do czego doprowadziliście? Dlaczego to mięso, szczególnie wieprzowina, jest tak drogie? Jeszcze w 2015 r. stad trzoda chlewnej było 250 tys., ale już w 2019 r. została połowa. Kolejne przykłady. Ceny odpadów. Będę powoływała się na ogólne dane instytucji rządowej, Głównego Urzędu Statystycznego albo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proszę bardzo: ceny odpadów. To państwa nominat, ówczesny prezes UOKiK pan Marek Niechciał powiedział, że podwyżki cen odpadów rozpoczęły się w 2017 r., a potem z roku na rok ceny zaczęły rosnąć. Niestety cierpią polskie rodziny. Jeśli chodzi o żywność, ten słynny paragon, na który dzisiaj, wiem, jesteście przygotowani, to w 2015 r., kiedy wasz prezydent Andrzej Duda poszedł zrobić zakupy, za kilka produktów zapłacił 37,02 zł.

Szanowni Państwo! Podatek cukrowy, warzywa, cukier. Mówicie: susza. Dzisiaj jest zupełnie inny trend światowy, który nazywa się renaturyzacja. Tak robi cała Europa. Dzisiaj szykuje się w Polsce wielka susza, wielka, dlatego że nie potraficie sobie też poradzić ze środowiskiem naturalnym.

Energia elektryczna. Ale nic dziwnego, jak stawiacie głównie na węgiel, i to ten z Rosji. natomiast niszczycie odnawialne źródła energii. Wasz minister Tchórzewski ogłosił zezłomowanie wszystkich istniejących wiatraków. Za to zapłacą polskie rodziny. Co z nich zostaje? Dane GUS-u pokazują, że z 500+ zostaje 270 zł. a emerytom po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, po opłaceniu rachunków, wydatków tak naprawdę na codzienne życie pozostaje 8 zł dziennie. To jest przerażające.

Wam łatwo jest oddawać pieniądze, które my skumulowaliśmy.

Dziękuję serdecznie. Będzie czas na zdawanie pytań.

Udzielam głosu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za to pytanie, bo myślę, że pytanie, które było skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokaże szereg działań, które podejmowaliśmy w ostatnich 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. pokazujących, na ile sytuacja polskich rodzin się poprawiła i dalej się poprawia.

Myślę, że polskie rodziny, które korzystają z tych wszystkich programów, które rząd realizuje, najlepiej o tym mogą zaświadczyć.

W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 4918 zł. Oznacza to przyrost w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego o prawie 5%. Jeżelibyśmy popatrzyli na dynamikę w ostatnich latach. Przeciętne wynagrodzenie wzrastało w tym okresie na poziomie 11%. To jest ta różnica między naszymi rządami a państwa rządami. W ostatnich 30 latach w ciągu jednej kadencji to był najwyższy wzrost wynagrodzeń. Jeśli chodzi o kwestię związaną z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, to warto tutaj też podać przykłady, o których mówimy.

Pan poseł zawsze lubił takie porównania, to panu podam zaraz przykłady, jak to wygląda.

Będziemy to porównywać do płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia.

Po prostu siła nabywcza i wynagrodzenia to są rzeczy, które są zbieżne, ale to trzeba wiedzieć i się trzeba czegoś nauczyć.

Proszę państwa. Panie ministrze, mam prośbę. Niech pan.

To są olbrzymie środki, które wpłynęły do budżetów polskich rodzin. Jakoś nie przypominam sobie, żeby za waszych czasów było coś podobnego.

Chodzi o program, który wspiera osoby niepełnosprawne, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

To jest ogromny wzrost nakładów na politykę rodzinną Te środki trafiają do polskich rodzin.

Chciałem przywitać uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Dobrej wraz z wychowawcami. Witamy was serdecznie. Proszę państwa, mam mały dylemacik, który zmusza mnie do podjęcia decyzji.

Wysoka Izbo! Dzisiejszy temat informacji bieżącej zaproponowany przez Platformę Obywatelską wpisuje się w takie polskie powiedzenie: tonący brzytwy się chwyta. Wystąpienie pana ministra bardzo wyraźnie pokazało państwu, jak bardzo poprawiła się sytuacja dochodowa polskich rodzin.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Marzenę Okła-Drewnowicz z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Tak jak pani chciała, pani poseł. Twardo walczymy. No dobrze. Niestety to za mało, żeby się odnieść, ale chcę powiedzieć tylko tyle, chcę powiedzieć tylko.

2 mln osób nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Czy prawdą jest, że jeszcze w 2015 r. liczba emerytów, którzy mieli najniższe emerytury, wynosiła niespełna 80 tys., a za waszych rządów w ubiegłym roku to już jest 300 tys. Ostatnie pytanie. Pan powołuje się na to, że wprowadzacie, że realizujecie systemowe rozwiązania, takie jak: maluch, program „Senior+”, a jeszcze bym dopowiedziała, że roczne urlopy rodzicielskie, czy też jeszcze mogę dopowiedzieć: dofinansowanie do niań. Pytanie, kto to zrobił. Więc pytanie: Co zrobiliście w przypadku wprowadzania systemowych rozwiązań? Znam tę odpowiedź niestety, bo nic. I to jest cała wasza praca, jeśli chodzi o systemowe rozwiązania. Pani poseł, widziałem w pani oczach przez chwilę konsternację. Pani jeszcze będzie miała na koniec 5 minut. No super.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż chcę powiedzieć, że dla pracowników sfery budżetowej, emerytów, rencistów. Tak de facto to ludzie, którzy nie są w stanie żyć do pierwszego, ponieważ koszty życia poszły mocno w górę. Otóż pan minister przed momentem mówił na mównicy, a można powiedzieć, że nawet udowadniał, że jest taniej. 8 stycznia zakupiłem te same produkty spożywcze co prezydent Andrzej Duda.

Myślicie, że ludzie nie chodzą do sklepów, nie kupują, nie wiedzą, że jest drożyzna? Chcecie wmówić, że jest taniej? Nie wmówicie. Ale wiecie, co jest najgorsze? Mieszkańcy Brzezin się zgłaszają, że. Zgłaszają się do premiera, żeby cokolwiek z tym zrobił. Wy nic z tym nie zrobiliście. Jedyne, co robicie, to na posiedzeniu tego Sejmu wprowadzacie kolejny podatek i opłatę (Dzwonek), żeby ściągnąć 3 mld zł. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Ministrze! Tak naprawdę to należałoby zrobić to, co pan minister zrobił, a więc podziękować państwu za tę informację bieżącą, za to, że można przedstawić fakty.

Dlaczego nieszczere? Państwo dzisiaj zadajecie pytanie, co zrobił rząd, a was ludzie, przeciętny obywatel obchodzi tyle, co po wyborach w rozmowach u Sowy było powiedziane: dzisiaj to benzyna może już być nawet po 7 zł.

I tutaj, z ław, tak jak dzisiaj krzyczeliście: A niech się młodzi emeryci wezmą do pracy. Wszystkie projekty ustaw, które miały polepszać los emerytów, były odrzucane. A pan tutaj dzisiaj mówi o tym, że wzrosły koszty pogrzebu. To właśnie Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska z PSL obniżyli nawet zasiłek pogrzebowy. I dzisiaj mówicie o cenach produktów.

Pani poseł Izabela Leszczyna. Bardzo dziękuję. Otóż jest śmiech wśród posłów PiS-u, gdy mówimy o tym, że w Polsce wzrasta skrajne ubóstwo, gdy mówimy o tym, że seniorom nie wystarcza na jedzenie, że kupują najtańsze niezdrowe produkty. Śmiech z tej strony sali pokazuje prawdziwą twarz PiS-u i prawdziwą twarz tej partii. Im wystarczy na wszystko. PiS-owi wystarczy na wszystko, bo oni pod stołem brali nagrody, które im się przecież należały. Drugi problem tej debaty jest taki, i to jest skandaliczne, że minister pracy nie rozumie, o czym dzisiaj rozmawiamy. My mówimy o inflacji. Mówimy o drożyźnie+. Wy w ogóle nie wiecie, o czym mówicie. Minister powinien wiedzieć, że te wszystkie dobrodziejstwa, które pan stąd wymienił, to były działania proinflacyjne. Potwierdził pan po prostu naszą tezę. One uderzają w dochody ciężko pracujących Polaków, bo bogactwo bierze się z pracy. Zrozumcie to wreszcie. A wy ludzi zniechęcacie. Od 4 lat zniechęcacie ludzi do pracy. Minister powinien też wiedzieć, że Narodowy Bank Polski odpowiada ze stabilność cen, za wartość polskiego pieniądza, czyli prezes Glapiński. Ale chyba jest tak, że prezes Glapiński jak pani Przyłębska z Trybunału Konstytucyjnego słucha dyrektyw partyjnych i zapomniał o tym, że ma narzędzia i ma obowiązek dbać o to, żeby ceny nie rosły najszybciej w całej Europie.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze, dziękuję. Prosimy panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Kto jak kto, ale minister powinien wiedzieć, że nie chodzi o wartość nominalną wynagrodzenia czy emerytury, tylko o siłę nabywczą portfela. To jest jedna kwestia. Druga - pan minister również powinien wiedzieć, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z zasiłków. A jedna z pań tu powiedziała: Halo, tu Ziemia. To ja powiem panu, jak wyglądają fakty. Drożyzna dziś to już nie tylko i wyłącznie żywność, nie tylko i wyłącznie rachunki za prąd i inne media, wywóz nieczystości itd. Drożyzna dzisiaj dotyka najbardziej wrażliwej, trudnej sfery naszego życia, czyli zdrowia.

Szanowni państwo, lek Prograf, który przyjmują pacjenci po przeszczepie nerek, wątroby. Przyszedł do mnie pacjent, wyborca, który kwartał temu kupił taki lek - zapotrzebowanie kwartalne, ale ta sama liczba opakowań, kapsułek, ten sam rodzaj, producent, ta sama apteka - za 31,84 zł. Wiecie, ile zapłacił na koniec stycznia po kwartale za (Dzwonek) dokładnie tę samą dawkę, tę samą ilość i ten sam lek? Wiecie, jaki to jest wzrost? 270%. dotykająca najbardziej wrażliwej sfery naszego życia. Panie Ministrze! No chyba sami państwo nie wierzycie w to, co mówicie z tej mównicy. Przed chwilą usłyszeliśmy od pani poseł z Platformy, że Platforma Obywatelska, oddając władzę w kraju, skumulowała pieniądze. No to państwo myślicie, że po 4 latach Polacy zapomnieli, jaka była prawda? To ja w takim razie państwu przypomnę. To wasz minister finansów w 2015 r. mówił: Pieniędzy nie ma i nie będzie. Po prostu tych pieniędzy nie zostawiliście, zostawiliście państwo w tragicznej sytuacji finansowej. A dzisiaj mówicie, macie odwagę powiedzieć: My zostawiliśmy skumulowane pieniądze. No naprawdę szczyt hipokryzji. Właśnie wracam z posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej, na którym omawialiśmy informację. o sytuacji osób starszych w Polsce, i tam przedstawiciele seniorów pozytywnie oceniali odczuwalną, realną poprawę sytuacji materialnej.

Realny wzrost płac za naszych rządów o ponad 19%. Płaca minimalna wzrosła o 850 zł. Panie Ministrze!

Zapraszam pana posła Tomasza Piotra Nowaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przyczajony tygrys, ukryty smok - to jest inflacja. Ona drzemie. Ona dopada nas, kiedy stajemy przy półce sklepowej. Ostatnio w sklepie spotkałem staruszkę, emerytkę, która miała 100 zł w ręce i chciała kupić produkty, które jeszcze 2 miesiące temu kupiła za te 100 zł. Moja emerytura nie starcza na te podwyżki, które są w tej chwili. Przyczajony tygrys, ukryty smok - to inflacja. Ale także ceny energii, które sztucznie staracie się zdusić. One już w tej chwili wybuchają we wszystkich firmach produkcyjnych, które dostarczają do sklepu towary. 40-procentowy wzrost cen energii dla firm. To musi się przełożyć - i przekłada się - na portfel emeryta, portfel tej drobnej kobiety, która z płaczem odeszła od lady, nie mogąc zrealizować podstawowego portfela zakupowego. Przyczajony tygrys, ukryty smok - to jest inflacja, która zeżre także nasze oszczędności, która spowoduje, że nasze przyszłe emerytury stracą na wartości. Jeśli będzie utrwalanie w tej chwili takiego systemu jak np. w energetyce (Dzwonek), zamiatanie wszystkiego pod dywan i udawanie, że ten system, który jest, jest systemem, który powoduje, że jest najtańsza energia, to znajdziemy się w wielkim niebezpieczeństwie. Pani poseł Urszula Rusecka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Pani poseł pytała, jaka jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości. To ja jej odpowiem. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości polskim rodzinom po prostu żyje się lepiej. No to tak zniechęcamy, że za państwa rządów inflacja wynosiła ponad 13%, a za naszych rządów - 5,1. Ja panu odpowiem, mój panie drogi, że za naszych czasów dochody za 4 lata, państwa dochody, wzrosły o 146 mld. A za państwa rządów, 8-letnich, dochody wzrosły tylko o 53 mld. A jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, to proszę sobie przeczytać raport NIK-u z 2015 r., kiedy szefem NIK-u był wasz poseł.

Ile wynosił dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2015 r., a ile wynosi teraz? Proszę państwa, nie uda się wam ta hucpa i ten temat, który teraz próbujecie forsować w kampanii.

Wtedy możemy rozmawiać o tym, że to jest naprawdę dobry budżet. Schab - plus 40%, ziemniaki - plus 70%, kapusta kiszona - plus 100%. To informacja dla pana prezesa.

Można by pomyśleć, że rząd prowadzi świadomą politykę prozdrowotną. Nie od dziś przecież wiadomo, że tradycyjne polskie dania niekoniecznie są zdrowe. Energia+, gaz+, śmieci+, woda+. Woda to chyba jednak minus, bo jest jej w Polsce mało, krytycznie mało, a o działaniach rządu, by to zmienić, nie słyszałem w ogóle. Dramatycznie rosną koszty utrzymania w domach pomocy społecznej. Tego nie wiecie. Tylko zabieracie pieniądze samorządom. Samorządy są pozostawione na pastwę losu. W wyniku tych wszystkich plusów spada rentowność małych i średnich przedsiębiorców. Co opowiadali? Obnażyli kłamstwa pana ministra, który mówi o podatku cukrowym. Opamiętajcie się. Przyznajcie się, że nie potraficie rządzić. do swoich piaskownic, panie Ziobro i panie Morawiecki, do skansenów, panie prezesie i panie Terlecki. Tam jest wasze miejsce. Ostatnią minutkę.

Tak? Może by panu dało do myślenia to, że są inni posłowie i dzięki temu, że pan mówił minutę dłużej, właśnie posłanka Platformy wypadła z ostatniego miejsca. Pani posłanka Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! ASF panuje już w całej Polsce. Mamy bardzo sprawny program drożyzna+, mamy bardzo sprawny program 41 nowych opłat i podatków. Mamy program energia+, bo Polacy płacą coraz więcej za energię. I w tym momencie rodzi się jedno podstawowe pytanie: Co z pracownikami sfery budżetowej?

Nawet nauczyciele, których podwyżkami się tak chwalicie, nie dostali tak wysokiej podwyżki. A co z pracownikami kultury? Co z pracownikami sądów? Co z pracownikami wszystkich praktycznie instytucji państwa? Bardzo łatwo podnosi się podatki. Bardzo łatwo się dekretuje, szczególnie w przypadku pracowników firm prywatnych, wyższą najniższą krajową. Ale kiedy zadbacie o tych, za których odpowiadacie, czyli tych, którzy są opłacani z budżetu? Najwyższy czas, żebyście zakończyli program drożyzna+.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Barbara Dziuk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Janusz Cichoń z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Rozmawiamy o inflacji, panie ministrze, a to w gruncie rzeczy podatek, i to podatek szczególnie dotkliwy dla osób najbiedniejszych. Skąd się ta inflacja bierze i jaki jest we niej udział rządu? Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że gigantyczny, bo to rząd PiS-u tę inflację napędza. Korzystanie z wód w przemyśle, rolnictwie i energetyce. Ścieki, odprowadzanie tych ścieków w rolnictwie, w przemyśle, opłata denna, deszczówka, opłata przejściowa od energii elektrycznej, opłata od nieruchomości komercyjnych, podatek od instytucji finansowych, opłata emisyjna od paliw, opłata paliwowa, śmieci - to nie wszystkie podatki, które wprowadziliście bądź podnieśliście. W tle za chwilę pojawi się opłata mocowa, podatek od sprzedaży detalicznej. Zapłacą za to Polacy, wzrośnie inflacja. Wygląda na to, że mamy do czynienia po stronie PiS-u z taką nieustającą promocją. Polacy do promocji podchodzą nieco inaczej. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Anna Ewa Cicholska z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Wysoka Izbo! Możecie nie wiem jak krzyczeć, nie zakłamiecie państwo rzeczywistości. Los polskich rodzin, szczególnie tych wielodzietnych, emerytów, rencistów, seniorów - za rządów Prawa i Sprawiedliwości ich sytuacja znacznie się poprawiła. Żyją o wiele lepiej, nareszcie mogą żyć godnie. Szanowni Państwo!

To wy zamroziliście za swoich rządów podwyżki dla sfery budżetowej. Panie Ministrze!

Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Codziennie obserwujemy, jak rząd PiS, jak dobra zmiana zagląda do naszych portfeli. Wasze zapewnienia sprzed 5 lat o dobrobycie, jaki nas czeka, nie mają pokrycia w faktach. Zaczynając od codziennych zakupów podstawowych produktów żywnościowych, obserwujemy wzrost cen, np. jajek - dwukrotnie, cukru czy chleba - przynajmniej o 1/4. Wraz z wzbogaceniem się społeczeństwa ich wydatki na żywność powinny maleć, tymczasem koszty zakupu żywności wzrosły. Średni koszt zakupu podstawowych produktów żywnościowych w ciągu 5 lat wzrósł o 27%. Jak więc bogacimy się jako społeczeństwo, skoro mimo wyższych pensji możemy kupić tyle samo co 5 lat temu? Mamy tu przykład tego, jak nieodpowiedzialna polityka, którą stosujecie, wpływa na wzrost inflacji i zabiera Polkom i Polakom ciężko zaoszczędzone i zarobione pieniądze. Ale oczywiście to tylko jeden sposób zaglądania do portfeli Polaków. Samorządy w całej Polsce mają problem ze swoimi budżetami, a powodem tej sytuacji są wprowadzone przez was dereformy. Ograniczyliście ich dochody z PIT-u, np. w Olsztynie, z którego pochodzę, zwrot podatku PIT zmniejszył przychody miasta o 37 mln zł - to jest 14%. Nałożyliście jednocześnie większe wydatki, jak wynagrodzenia nauczyli, czego nie rekompensujecie w subwencji oświatowej. Kolejne to podniesienie płacy minimalnej i pozostawienie samorządów bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. To zamach na samorządy, aby postawić je w niekorzystnym świetle. Panie ministrze, dlaczego jak jest tak dobrze, to wszystko drożeje? Proszę pana posła Pawła Hreniaka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Myślę, że państwo z opozycji źle dobrali temat dzisiejszej dyskusji, bo naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o wsparcie dla polskich rodzin. Do 2016 r. nie było żadnego całościowego programu wsparcia polskich rodzin, co skutkowało m.in. tym, że w roku 2015 wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego były na wyższym poziomie niż obecnie. W związku z tym pytanie do państwa z opozycji: Jak myślicie, kiedy Polakom, polskim rodzinom żyło się lepiej - dziś czy za rządów Platformy Obywatelskiej i ich koalicjantów? Wskazują na to m.in. wskaźniki, o których powiedziałem. Panie ministrze, pytanie do pana ministra: Ile polskich dzieci w 2015 r., a ile dziś jest objętych wsparciem z budżetu państwa? Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Jarosława Urbaniaka, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Posłanki i Panowie Posłowie z PIS-u! Zaklinacie rzeczywistość. To wszystko nieprawda. To nawet kontrolowany przez was GUS w swoich danych pokazuje, że polskim rodzinom żyje się coraz gorzej, bo nie umiecie zarządzać Polską, bo nie znacie się na ekonomii. Przecież, panie ministrze, pan w pierwszych słowach przyznał się do porażki. Pan powiedział, że rząd PiS od 5 lat podejmuje liczne działania. Tak, bardzo liczne, tylko że nieskuteczne. W tym tkwi problem, że jesteście kiepscy w tym zarządzaniu. Przecież większość waszych wypowiedzi mówi o 500+. Zaproponowaliśmy temat dzisiejszej debaty: drożyzna, a nie średnia inflacja. A drożyzna to ceny towarów podstawowych: chleba, masła, sera, mięsa.

My mówimy o tym, z jaką trwogą emeryt otwiera kopertę z zakładu energetycznego, żeby zobaczyć, jak mocno zdrożał prąd. My mówimy o tym. a wy nic z tym nie robicie. Pan minister Cichoń wymienił zaledwie kilka podatków (Dzwonek), które wprowadziliście lub podnieśliście. To jest przyczyna tej drożyzny. Dziękuję serdecznie. Przepraszam panią poseł Krzywonos, ale niestety nie mogę pani udzielić głosu, gdyż potencjalny czas zabrał pan poseł Artur Łącki.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dziękuję opozycji za troskę o polskie rodziny, za troskę o ludzi, o mieszkańców naszego kraju.

W związku z tym mam pytania do pana ministra, ponieważ mówił pan o programach wspierających polskie rodziny. W związku z tym mam pytania do pana ministra. Jak wygląda wzrost świadczeń w przeliczeniu na jedno dziecko? O ile więcej środków z budżetu państwa jest przekazywanych dla rodzin w porównaniu ze środkami w roku 2015?

Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z danymi się nie dyskutuje, dane się przyjmuje.

Jaki, panie ministrze, jest wniosek? Polki i Polacy wydają więcej na swoje utrzymanie.

Zazwyczaj te gospodarstwa składają się ze starszych kobiet. Druga sprawa. Polacy coraz więcej wydają na prywatne usługi medyczne i na leki.

Wysoka Izbo!

Kiedy rosły koszty utrzymania i drożyzna za rządów PO-PSL, jedynym argumentem ze strony rządzących było strzelanie z broni gładkolufowej do protestujących górników, którzy bronili swoich miejsc pracy i prawa do godnego wynagrodzenia. To są fakty. Mam prośbę, aby pan minister w swoim czasie zreedukował trochę opozycję i wskazał na prosty mechanizm, a mianowicie siłę nabywczą pieniądza, jeżeli chodzi o relacje wynagrodzenia minimalnego i możliwości zakupu ewentualnie wybranych towarów, jak również wynagrodzenia średniego i wybranych artykułów spożywczych. Na koniec zaś cytat dla szanownej opozycji: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spada u nas najszybciej spośród europejskich krajów. Choć 7 lat temu byliśmy w ogonie Europy, teraz sytuacja finansowa Polaków jest lepsza niż Hiszpanów, Włochów czy Węgrów. Kto to napisał? Dziękuję serdecznie. Proszę pani, przeprosiłem już za to, w związku z tym nie mam ochoty po raz drugi przepraszać. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Inflacja jest PiS-owi na rękę, bo inflacja uratuje ten rzekomo zrównoważony budżet i tylko ona może ten budżet uratować. Pan to sam potwierdził, dlatego że pan się nawet nie zająknął o jakichkolwiek mechanizmach czy jakiejkolwiek koncepcji rządu, aby panować nad inflacją. Nie ma żadnych instrumentów? No nie ma, waszym zdaniem nie ma. Czy parę emerytów czy parę nauczycieli z budżetówki stać na przeprowadzanie remontu mieszkania?

A więc jest pięknie? Udział żywności w wydatkach gospodarstw domowych sięgnął 25%, znowu wrócił na ten poziom. Trzeba to zauważyć. Więc pytam, co zrobicie, aby np. stabilizować albo zatrzymać ten trend na rynku usług. Dziękuję serdecznie. No dobrze. Zapraszamy. Nie ma pana posła? Pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak, tak, drożyzna+.

A z tą drożyzną to dopiero początek. To, czym się chwalicie, czyli cała ta polityka prorodzinna, wszystkie wasze plusy, zostało już w dużej części pochłonięte przez szalejącą drożyznę. Spowolnienie gospodarcze, powtarzam, jest faktem, a skutki tego spowolnienia odczuwają Polki i Polacy. Nie słuchaliście opozycji, nie zapobiegliście inflacji, a wręcz przeciwnie. Ubiegłoroczne działania rządu związane z cenami prądu, podniesieniem płacy minimalnej, nowymi stawkami VAT już i tak trudną sytuację spotęgowały.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Henryka Krzywonos-Strycharska jest dopisana. Pani poseł, proszę bardzo. Pan poseł Paweł Rychlik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Marek Sowa, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister nie powiedział o kilku sposobach, którymi można sobie z drożyzną poradzić. Oto przykłady.

Jest również inny sposób radzenia sobie z drożyzną. Tak jak poradzili sobie działacze PiS-u z Dolnego Śląska. Można też sobie poradzić z drożyzną, tak jak sobie poradził pewien poseł, który ma niektórych w nosie. Przypomnę, że będąc w 2016 r. wiceprezesem PGNiG zarobił ponad 2 mln zł. Poseł Kowalski. Ale nas nie interesuje jak sobie radzą PiS-owcy. Nas interesuje, jak z drożyzną mają sobie poradzić ludzie pracujący np. w jednym ze szpitali w zachodniej Małopolsce. Został zaaneksowany. Dyrektor musi płacić 25% więcej za energię, kilkadziesiąt procent więcej za śmieci. Nie stać go na podwyżki.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Agnieszka Górska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie kadencje wprowadził szereg ustaw, wychodząc naprzeciw problemom polskich rodzin, dzięki czemu znacząco poprawiła się sytuacja rodzin, zarówno sytuacja materialna, jak i sytuacja, jeśli chodzi o opiekę, bazę szkolną czy przedszkolną.

Szanowni państwo, to dopiero była drożyzna plus. Przypomnę, że nie było wsparcia 500+, tej drugiej strony, która finansowo niwelowałaby drożyznę zafundowaną przez Platformę Obywatelską i PSL. Dopiero wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości znacząco odbudowało pozycję polskiej rodziny. Rząd wskazał, to oczywiste, że dzieci, rodzina to przyszłość każdego narodu, sprawy rodziny traktując jako działania priorytetowe. Dziś rodziny, samorządy i inne instytucje mogą korzystać z nowych form wsparcia dzięki polityce prorodzinnej Prawa i Sprawiedliwości.

Nie chcę tego robić. Szanowny Panie Marszałku!

Mówię: wprowadzenie, bo to nie jest przypadek - to były systematyczne, zaplanowane, przemyślane działania. Albo... 41 nowych podatków, nowe, skomplikowane obciążenia biurokratyczne i nieopanowane rozdawnictwo, które odbywa się kosztem aktywnych, przedsiębiorczych, pracujących Polaków.

Tam, gdzie mieszkają seniorzy, silne uderzenie, i nie dlatego, że spółdzielnie chciały, tylko dlatego, że taka jest polityka rządu premiera Morawieckiego. Żywność - kilkadziesiąt procent. Wreszcie skok na oszczędności emerytalne i grabież 15% środków zgromadzonych na emerytury. I, rzecz haniebna, wywłaszczenie dzieci i małżonków z oszczędności emerytalnych po zmarłych rodzicach i małżonkach. To jest doprawdy haniebna sytuacja. I to jest dramatyczna prawda o rządach premiera Morawieckiego i jego rządu. A państwo udają propagandowo, że nic się nie dzieje. Kogo chcecie oszukać? Panie ministrze, przecież mieszkamy w tym samym regionie, a pan tak mówi, jakby nie zauważał tej drożyzny, która się u nas również pojawiła. I to jest efekt rządów premiera Morawieckiego i jego ministrów. I pytanie: Czy o to chodziło, żeby Polacy musieli zastanawiać się w sklepie, za co kupić i jak przetrwać znowu do pierwszego? Pan poseł Jakub Rutnicki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wystarczy pójść na targowisko, pójść do sklepu. Wiecie, co ludzie mówią? Tak drogo jak za PiS-u jeszcze nigdy nie było.

To jest wasza wina i wy to konkretnie robicie. Jak wygląda sytuacja? Jeszcze kilka miesięcy temu z tej mównicy premier Morawiecki mówił, że ceny prądu nie wzrosną, szanowni państwo - nie wzrosną. A jakie są fakty? Wzrosły o kilkanaście procent. Cena masła o 40%, wzrost cen żywności rok do roku. Rekord wzrostu cen żywności, o ponad 7% rok do roku. A wiecie, dlaczego?

powiedziała, że się należały. Tak, należały się, bo na końcu ich nie oddaliście. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja w przeciwieństwie do niektórych polityków PiS nie chowam się za ochroniarzami i wychodzę do ludzi. Wychodzę do ludzi na targach, wychodzę do ludzi na ryneczkach i rozmawiam z nimi. No i co? ...mieszkańców Polski, ale też województwa podlaskiego? To jest po prostu powszechnie panująca drożyzna, drożyzna w sklepach.

Te dwa produkty to wzrost o 50%.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Jak dziś rano trzeba było z PiS-em głosować za kolejnym podatkiem, kolejną drożyzną, Lewica była w komplecie i była aktywna, a w tej chwili w czasie debaty jedyny poseł z Lewicy, który zabrał głos, to Dariusz Joński. Szanowni państwo, ja wiem, doskonale wiem, jak państwo będziecie to uzasadniać, jak będzie to prezentował rząd. Będzie mówił tak jak minister Skurkiewicz. Szanowni państwo, rząd mówi: Ludzie zarabiają więcej, dobrze im się powodzi, stać ich. Ale to jest tak samo prawdziwe jak to, co powiedział minister Skurkiewicz w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych, i było to bezczelne: Ludzie dali więcej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo im się lepiej powodzi. Szanowni państwo, to bzdura. Kolejna bzdura. Zawieźcie go w tej kampanii, niech zrobi takie same zakupy. Zestawcie te dwa paragony.

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w trybie sprostowania.

Widzę, że pan Joński jak zwykle błyskotliwy i inteligentny. Cieszę się. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Chciałam. Jeżeli jesteście tacy miłosierni, to już dziś zdejmijcie kryterium dochodowe - do 500 zł - dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W ogóle wydaje mi się, że nawet nie wiecie, co to znaczy być niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

To jest prawda. To jest prawda, dlatego że wiele osób dzwoni do mojego biura i mówi, że dokłada bardzo dużo pieniędzy. Niepełnosprawni masła nie jedzą. Niepełnosprawni jedzą margarynę. Powiem tak: niepełnosprawni w Polsce dzisiaj żebrzą o 1%, zbierają plastikowe nakrętki. Nie mają na turnusy rehabilitacyjne, na pampersy, siedzą w czterech ścianach, bo nie mają asystentów. Skandaliczne zachowanie podczas 40 dni protestu. To są te zamknięte toalety, okna.

Przecież miało być lepiej. Zapraszam pana posła Konrada Berkowicza z Konfederacji. Wysoka Izbo! Na początek zacytuję pana prezydenta Andrzeja Dudę, który niedawno powiedział: Musicie mieć państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. To są niestety normalne mechanizmy gospodarcze. Nic nie zdołamy na to poradzić. Że takie są mechanizmy gospodarcze, że Polaków nigdy nie będzie stać na więcej.

W normalnym państwie siła nabywcza rośnie w momencie, kiedy rozwija się technologia. Tak. ...organizuje się gospodarka, zmniejsza się biurokracja, która przeszkadza przedsiębiorcom w budowaniu gospodarki tego kraju.

Podnosicie ceny produktów, podnosicie podatki i musicie to robić, bo stosujecie nieodpowiedzialne rozdawnictwo. Przestańcie ograbiać Polaków z pieniędzy po to, żeby później za te pieniądze robić z siebie dobroczyńców. Za swoje pieniądze. Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Dziuk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska jest normalnym krajem, ma demokratycznie wybrany rząd.

Mam pytanie do pana ministra. Czy wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz wsparcie w ramach programów przełożyło się na sytuację gospodarstw domowych? Totalna opozycja kwestionuje fakty, a z faktami się nie dyskutuje. Opozycja miała hasło: By żyło się lepiej. Kolegom. A my wprowadzamy zasady i finansowanie, żeby się żyło lepiej Polakom. Panie Ministrze! Gospodarka nasza naprawdę jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o rozwój, w Europie, w świecie. I dzięki temu naprawdę pensje wzrastają, a przede wszystkim jest większy szacunek do każdego Polaka. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Henrykę Krzywonos-Strycharską. Dopuszczam pana posła Ajchlera i zamykam listę, bo za 15 minut musimy zakończyć pytania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Szanowna Izbo! Panie Ministrze! Państwa sztandarowe 500+ nie podlega waloryzacji. Przypominam to od początku. Dlatego też spróbowałam to wszystko porównać i zobaczyć, co można kupić za 500+.

Teraz, proszę państwa, po tym wszystkim chciałam tylko oświadczyć, że posłem się bywa, człowiekiem trzeba być zawsze, więc ja znam swoje miejsce, chodzę na rynki, spotykam się z ludźmi i wiem, co ich boli. Chciałam państwa zaprosić na Kaszuby, by zobaczyć, ile dzieci jest głodnych. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Rafała Adamczyka z klubu parlamentarnego Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Koleżanki Posłanki z Lewicy i Posłowie z Lewicy! Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Wysoka Izbo! Wysoki Sejmie!

i powinniście się bić głęboko w piersi. Ale musicie również wiedzieć, że może to was dotyczyć. A życzę wam przede wszystkim zdrowia. Wysoka Izbo!

Pani poseł, 5 minut. Jeszcze raz, panie marszałku, dziękuję. Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Dobrze byłoby, żeby o kwestiach najbardziej dotkliwych dla Polaków dyskutować naprawdę rzetelnie. Nie da się do końca dyskutować rzetelnie, ponieważ posłowie Prawa i Sprawiedliwości żyją w swojej bańce. Naprawdę państwo nie wiecie, jak żyją polskie rodziny, jak żyją rodziny z dziećmi, szczególnie młode rodziny - i zaraz podam przykład - jak żyją emeryci i renciści. Zgadzam się z państwem w tej części, kiedy mówicie, że pensje rosną i emerytury rosną. Problem polega na tym, że z nich na życie tak naprawdę niewiele zostaje. O tym, że Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie jest już więcej, wszyscy wiemy, bo o tym już mówiłam. O tym, że emerytów najuboższych jest prawie 4 razy więcej w stosunku do roku 2015, też już mówiłam. O tym, że na te podwyżki prądu wpływa wasza nieodpowiedzialna polityka. bo postawiliście głównie na węgiel, niszcząc tak naprawdę odnawialne źródła energii, nie wspierając ich, też mówiłam.

To państwo zniszczyliście np. program „Mieszkanie dla młodych”, bo wy go zlikwidowaliście. Dzięki temu programowi ponad 100 tys. tak naprawdę beneficjentów może mieć już dzisiaj swój własny dach nad głową. Staram się nie patrzeć już w tę stronę. Postaram się jakoś skupić, ale. No więc dziękuję.

Dobrze, ale to może nie bierzmy złych przykładów, tylko bierzmy dobre. Niech pani popatrzy na mnie. Państwo nie tylko ten program zlikwidowaliście, bo to jeszcze tak naprawdę chyba dałoby się jakoś wytrzymać, ale dołożyliście, szczególnie tym młodym ludziom, podatek bankowy. I to dzisiaj ci młodzi ludzie muszą brać kredyty obarczone większymi kosztami prowizji, opłat manipulacyjnych i jeszcze muszą brać ubezpieczenia. Tak to wygląda. Dlatego chcę państwu uświadomić to, że owszem, wynagrodzenia tych młodych ludzi rosną, ale również np. kredyt, który muszą wziąć na dach, który będzie dla ich rodziny, jest po prostu droższy.

Zobaczcie państwo, opłata za prąd - nagle mamy tam tak naprawdę kolejne koszty, np. opłatę mocową.

To wszystko są podatki, daniny, które tak naprawdę zbieracie od polskich rodzin. To powoduje, że dzisiaj koszty utrzymania polskich rodzin są dużo, dużo wyższe.

To dzięki nam one powstały. Przynajmniej dla części dzieci znajduje się miejsce w żłobku. Przedszkole - to my wprowadziliśmy przedszkole za złotówkę. To jest realna pomoc systemowa dla wszystkich polskich rodzin.

Zapraszam pana ministra.

Wysoka Izbo! Dziękuję za wszystkie pytania. Od razu odniosę się do wypowiedzi pani poseł, która występowała przede mną, dotyczącej programu „Maluch+” Pani poseł, przeznaczaliście na program „Maluch” 150 mln zł, my przeznaczamy 450 mln zł.

Ale jeśli popatrzymy na wzrost dochodów, to oczywiście dochody są wyższe i te wskaźniki w Polsce spadają.

Te wynagrodzenia rekompensują to, co jest dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji. Jeszcze raz powtórzę kwestie związane z emeryturami dotyczącymi najsłabszych grup.

Dotyczyć to będzie tych wszystkich, którzy mają emerytury na poziomie 1900 zł.

To jest duży przeskok, ale jakby w poprzednich latach konsekwentnie też to było podnoszone, dzisiaj byśmy mówili o zupełnie innym wskaźniku.

W 2015 r. na wsparcie dla dzieci przeznaczyliście państwo 2 mln, objęło to 2 mln dzieci.

To jest bardzo duże wsparcie i ono też rekompensuje w jakiś sposób kwestie, o których rozmawialiśmy.

Ważne też, myślę, by podać informacje dotyczące tych programów, które są związane z pomocą społeczną, bo oczywiście najsłabsze grupy też obejmujemy pomocą społeczną.

Był podnoszony temat płacy minimalnej i sytuacji na rynku pracy. Trzeba się zdecydować, czy chcemy podnosić płace minimalne, czy nie.

Mamy największą liczbę zatrudnionych w tej chwili w gospodarce, ponad 16 400 tys. To też pokazuje, że droga, którą obraliśmy, jest skuteczna, bo mamy niskie bezrobocie, dobry wzrost PKB, a jednocześnie realizujemy bardzo dużo programów społecznych, rodzinnych, które wspomagają rodziny, wspomagają rodziny emeryckie, wspomagają rodziny, które z tego programu mogą skorzystać.

Tu już jedna z pań posłanek odpowiedziała. 6-procentowy wzrost w tym roku, jeśli chodzi o sferę budżetową. Ale to trzeba przypomnieć.

Dziękuję za tę debatę i za te pytania. Myślę, że przedstawiłem państwu cały szereg działań, które podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, dotyczących wsparcia polskich rodzin, i to wsparcie jest bardzo duże.

To jest ogromny wzrost nakładów na politykę rodzinną. Pani poseł Okła-Drewnowicz w trybie sprostowania. minuta. Dziękuję. Panie Ministrze! Wiem, że jeden i drugi program jest na „m”, ale ja nie powiedziałam, że państwo zlikwidowaliście albo chcieliście zlikwidować program „Maluch” Ja powiedziałam o tym, że państwo zlikwidowaliście program „Mieszkanie dla młodych” dotyczący dofinansowywania mieszkań. Panie ministrze, dziękuję. Dziękuję posłom. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 171 i 198) Bardzo proszę pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie pośle, zapraszam.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rynek kolejowych przewozów otwarto dla konkurencji w roku 2007, natomiast rynek międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich - w roku 2010. Wspomniana dyrektywa otwiera na konkurencję również krajowe rynki przewozów pasażerskich, przyznając uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich.

Główne rozwiązania wprowadzone w przedmiotowym projekcie. Po pierwsze, wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Zgodnie z dyrektywą wprowadza się definicję tegoż przedsiębiorstwa dla określenia modelu relacji między zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem, w sytuacji gdy podmioty te są powiązane kapitałowo, handlowo i organizacyjnie, w sposób określony w przepisach rozporządzenia. Po drugie, wzmocnienie gwarancji niezależności zarządcy, m.in. poprzez wymóg zachowania odrębnej osobowości prawnej zarządcy infrastruktury od przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo - także od innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, oraz poprzez ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom. Nie będzie możliwe zlecanie wykonywania zadań zarządcy przewoźnikowi kolejowemu lub podmiotowi, który jest kontrolowany przez tego przewoźnika albo sprawuje nad nim kontrolę. Chodzi o szereg zakazów dotyczących łączenia w przypadku zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego określonej funkcji lub zajmowania stanowisk kierowniczych. Po trzecie, zapewnienie przejrzystości finansowej zarządcy, m.in. poprzez zakaz wypłaty przez zarządcę dywidend podmiotowi wchodzącemu w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, sprawującemu jednocześnie kontrolę nad tym zarządcą i przewoźnikiem kolejowym, a także zakaz wzajemnego udzielania pożyczek przez zarządcę i przewoźnika kolejowego. Po czwarte, wzmocnienie kompetencji nadzorczych prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. poprzez uprawnienie do żądania od zarządcy informacji o braku zdolności przepustowej czy też sprawowanie nadzoru nad negocjacjami, których przedmiotem są opłaty za dostęp do infrastruktury, oraz nad zawieraniem i wykonaniem umów o współpracy.

Po szóste, poprawa efektywności i transparentności procesu alokacji zarządzania infrastrukturą. Chodzi o możliwość wprowadzenia negocjacji w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, zmiany w zakresie monitorowania punktualności, rekompensat należnych z tytułu opóźnienia pociągu, obowiązku współpracy, informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny w przypadku infrastruktury kolejowej. Pozostałe zmiany w zakresie udostępnienia obiektu infrastruktury usługowej to uwzględnienie zasad dostępu do torów kolejowych znajdujących się w obiekcie infrastruktury usługowej, w tym również w portach, obowiązek ogłoszenia przeznaczenia do wynajęcia lub dzierżawy obiektu, który nie był użytkowany przez kolejne 2 lata, i wskazanie organu, którego zadaniem będzie ocena bezpośrednio zawartych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego. Wyznaczenie prezesa UTK do pełnienia funkcji niezależnego organu, którego zadaniem będzie bezpośrednia ocena zawartych umów w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, na podstawie tych przepisów zapewnia możliwość dodatkowej weryfikacji prawidłowości decyzji podjętej przez organizatora w zakresie bezpośredniego udzielania zamówień. Wysoka Izbo!

Mając powyższe na względzie, proszę Wysoki Sejm o przyjęcie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przyjętym przez Komisję Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Główne rozwiązania zawarte w projekcie to wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa zintegrowanego, wzmocnienie gwarancji niezależności zarządcy infrastruktury kolejowej, zapewnienie przejrzystości finansowej zarządcy. Zapewnia się transparentność finansową zarządcy infrastruktury, w szczególności przepływów i rozliczeń między nim a przewoźnikami lub innymi podmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Wzmacnia się kompetencje nadzorcze prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, poprawia się efektywność i transparentność procesu alokacji i zarządzania infrastrukturą. Pozostałe zmiany są w zakresie udostępnienia obiektu infrastruktury usługowej. Na zarządcę infrastruktury nakłada się obowiązek ogłoszenia przeznaczenia do wynajęcia lub dzierżawy obiektu, który nie był użytkowany przez kolejne 2 lata.

Wysoka Izbo!

Dziękuję serdecznie za poprawkę. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To nie jest zła ustawa, ponieważ każda ustawa, która cementuje nasz związek z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej, poprawia bezpieczeństwo naszego państwa, ale także obywateli. Ta ustawa wiąże nas ściślej z sieciami europejskiej kolei. To dobrze.

Dlaczego? Dlatego że ustawa wprowadza, przepisując wprost z dyrektywy, nową definicję przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości. Przewozy pasażerskie to takie, które będą wykonywane bez przystanków pośrednich pomiędzy dwoma miejscami położonymi od siebie w odległości większej niż 200 km, na liniach kolejowych specjalnie przystosowanych do prędkości nie mniejszej niż 250 km/h, wykonywane średnio z taką prędkością. I teraz na czym polega problem? Problem polega na tym, że Baranów, gdzie ma być ulokowany Centralny Port Komunikacyjny, leży 30 km od Warszawy. Ta linia Y wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sieci TEN-T z 2013 r. Ten podwójny Y jest wrysowany w załączniku tego rozporządzenia, które jest zobowiązaniem dla Polski do wykonania tej linii do 2030 r. To także nie mieści się w proponowanej w ustawie definicji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli przyjmiemy te rozwiązania, to nie będzie można w Polsce zrealizować przewozów kolejami dużych prędkości. Być może na tym zależy rządowi. Nie wiem, czy panu ministrowi. Ale nie zadał pan sobie trudu, aby wyjaśnić rozbieżność tej definicji z definicją, która jest zawarta w dwóch innych dyrektywach europejskich, m.in. w rozporządzeniu, które już przywoływałem, z grudnia 2013 r. o transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Jest też trzecia opcja: specjalnie zmodernizowane linie kolei dużych prędkości posiadające szczególne cechy ze względu na uwarunkowania związane z topografią, rzeźbą terenu, ze względów urbanistycznych. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli pozostawimy tę definicję, którą przyjmujecie bez refleksji, to w Polsce kolei dużych prędkości nie będzie. To znaczy, że nie zrealizujemy zobowiązania wynikającego z rozporządzenia z 2013 r. w sprawie sieci TEN-T. Dlatego Koalicja Obywatelska proponuje dwie poprawki. Jedna, dalej idąca, to skreślenie tej definicji i rozpoczęcie dialogu z Komisją Europejską, żeby wyeliminować te sprzeczności z (Dzwonek) różnych dyrektyw. To rząd powinien zrobić. Druga, nieidąca tak daleko, to modyfikacja tej definicji poprzez wprowadzenie następującego tekstu: „przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości to przewozy wykonywane bez przystanków pośrednich między dwoma miejscami położonymi od siebie w odległości większej niż 200 km lub odległości mniejszej niż 200 km, jeżeli dotyczy to połączeń między istotnymi węzłami transportowymi”

Dziękuję serdecznie panu posłowi. Proszę bardzo. Paulina Matysiak, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Procedowane zmiany zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw mają charakter wyłącznie porządkowy i niestety niewiele wnoszą, jeśli chodzi o to, by poprawić stan polskiej kolei. Podstawą prawdziwej reformy kolei w Polsce powinno być przekształcenie narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych SA w agencję rządową na wzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od blisko 20 lat na skutek ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowo” PKP PLK działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego.

Odpowiedzmy sobie na proste pytania: Czy w interesie spółki akcyjnej jest prowadzenie dużych inwestycji, jeśli w związku z tym rośnie jej majątek, a tym samym w kolejnych latach rosną koszty amortyzacji? Czemu środki unijne na kolej nie są wydatkowane tak, jak mogłyby być? Skąd ogromne opóźnienia w inwestycjach kolejowych, za które krytykowano już poprzedni rząd?

Dążenie do zbilansowania działalności zarządcy infrastruktury kolejowej prowadzącego tę działalność w formie spółki akcyjnej powoduje szereg patologii. Pierwszą z nich jest zaniechanie wielu inwestycji, które byłyby możliwe w innym stanie prawnym. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad staje się spółką handlową, nie powstaje kolejna obwodnica, droga czy autostrada lub, co gorsza, likwidujemy jakąś drogę krajową, bo spółka, nazwijmy ją na potrzeby tej dyskusji, Polskie Drogi Krajowe SA, optymalizuje swój majątek, aby obniżyć koszty amortyzacji oraz poprawić swój bilans. To jest niestety rzeczywistość polskiej kolei od 30 lat, tzw. ostre cięcie. Polska sieć kolejowa w 1989 r. to ponad 25 tys. km linii kolejowych, polska sieć kolejowa w 2019 r. to zaledwie 18 tys. km linii kolejowych. I nie chodzi tu wyłącznie o Jastrzębie-Zdrój, o Łomżę czy Mielec, na które lubi się powoływać premier Mateusz Morawiecki, ale o tysiące przystanków i stacyjek w małych lub większych miastach i miasteczkach, które zostały odcięte od świata, by optymalizować majątek PKP. Czy wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad likwidowałaby drogi i autostrady? Myślę, że minister Andrzej Adamczyk nie ostałby się nawet jednego dnia na swoim stanowisku. A jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom pod rządami ministra Adamczyka likwidowane są kolejne linie kolejowe w naszym kraju. Następna patologia wynikająca z obecnej formy prawnej narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej to stawki dostępu do torów. Aby zbilansować swoją działalność, PKP PLK stosuje jedne z najwyższych stawek w Europie. Wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej obciążają przewoźników zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Kolej staje się mniej konkurencyjna, koszty przewozu towarów koleją oraz ceny biletów są coraz wyższe. Efekt jest taki, że polską koleją podróżuje ponad 3-krotnie mniej pasażerów niż w 1989 r. oraz nadal o kilkadziesiąt milionów mniej niż przed reformą z roku 2000. Tak nie wygląda nowoczesne państwo, proszę państwa, panie ministrze. To można zmienić, ale musimy zacząć w końcu traktować kolej tak, jak traktujemy drogi. Kolej powinna mieć równe szanse. A stanie się tak tylko wtedy, gdy nie będzie obciążona dodatkowym garbem finansowym. Ten projekt o tym nie mówi. Zajmujecie się państwo drobiazgami, zamiast naprawić ten podstawowy problem. Naprawę kolei trzeba zacząć od dobrej organizacji, by wreszcie na wzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powstała agencja rządowa, która będzie odpowiadać za dworce i infrastrukturę kolejową. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy zagłosuje za przyjętymi i proponowanymi przez państwa rozwiązaniami, ponieważ doprecyzowują one kwestie prawne, ale będziemy w tej kadencji składać nasz projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (Dzwonek), bo temat ten traktujemy poważnie. Kolej po wielu latach zaniedbań zasługuje na prawdziwe wsparcie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jacek Tomczak, klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15. Wysoka Izbo! Projektowana ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie o transporcie kolejowym mających na celu wykonanie dyrektyw i wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Projektowane zmiany dotyczą możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom, sposobu ustalania rekompensat za opóźnienie pociągu, zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury, zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej, elementów planu biznesowego, zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi. Projektowane rozwiązania mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, co spowoduje wzrost konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej wynikający z równoprawnego traktowania w zakresie zapewnienia prawa dostępu dla wszystkich zainteresowanych podmiotów niezależnie od kraju członkowskiego, z którego pochodzą. Wprowadzone rozwiązania eliminują dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie. Ponadto w ustawie dodano rozdział 2aa „Gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy”, który ogranicza możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez innych uczestników rynku kolejowego, w szczególności przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami. W tym celu wprowadza się rozwiązania m.in. ograniczające występowanie konfliktu interesów, ograniczające możliwość zlecania zadań zarządcy innym podmiotom, zapewniające transparentność przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. Projekt ustawy rozszerza uprawnienia nadzorcze prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące m.in. negocjacji między aplikantami a zarządcami infrastruktury w przypadku ich prowadzenia, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania określonych informacji dotyczących rozdziału rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem i monitorowania wykonywania umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego.

Procedowany projekt jest istotnym elementem niezwykle ważnego procesu otwierania rynku usług kolejowych w Europie, procesu obarczonego oczywiście pewnymi ryzykami, ale też niosącego szereg szans rozwojowych. Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, oczywiście z poprawkami przedstawionymi przez komisję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, czas na zadawanie pytań. Czy ktoś z państwa jeszcze ma ochotę? Zamykam listę. Bardzo proszę, pani posłanka Daria Gosek-Popiołek z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że nie ma bezpieczeństwa na kolei bez zapewnienia pracownikom dobrych, komfortowych warunków pracy, godnych płac i bez dbałości o to, by zatrudniające ich podmioty przestrzegały prawa pracy. Ma to znaczenie zwłaszcza w momencie, w którym na polskich torach pojawiają się inne, zagraniczne podmioty. Bez maszynisty pociąg nie pojedzie. To nie jest konkurencyjna stawka, która by zachęcała do podjęcia tej pracy, bardzo trudnej, bardzo wymagającej. Zdarzają się niestety zbyt często przekroczenia dozwolonego czasu pracy maszynistów. Brakuje ludzi. Maszyniści muszą wyrabiać nadgodziny. Brakuje wyszkolonej kadry, a sam proces szkolenia, jak mówią o tym maszyniści, nie jest efektywnie zaprojektowany. Maszyniści mówią także o absurdach, np. mają minutę na zdanie czy przyjęcie lokomotywy. Przypomnę, że związki zawodowe zwracały się (Dzwonek) już do ministerstwa w tych sprawach. A więc moje pytanie: Czy i w jaki sposób chcą państwo dbać o prawa pracownicze i dobre warunki pracy na kolei u naszych narodowych przewoźników? Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Paulina Matysiak, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wygaszanie linii kolejowych, tak jak mówiłam przed chwilą, trwa od 30 lat.

Ostatni przykład, fizyczna likwidacja linii kolejowej nr 371 latem 2018 r., jest najbardziej skandaliczny. Likwidacja linii nastąpiła pomimo zapewnień ministra Adamczyka oraz ministra Bittela z 2016 r. i 2017 r., że nie będzie już dalszej likwidacji linii kolejowych, i pomimo protestów organizacji społecznych i mieszkańców. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Wiesław Szczepański, klub parlamentarny Lewica. Kilka dni temu poznaliśmy projekt „Strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) W województwie wielkopolskim planowana jest w ramach tego programu budowa 196 nowych linii kolejowych. Nowy przebieg szybkiej kolei jest skrajnie niekorzystny dla Ostrowa Wielkopolskiego. Tak naprawdę wyklucza Ostrów ze strategicznych połączeń z Wrocławiem i Poznaniem. Tak naprawdę jest to rozbiór ostrowskiego węzła kolejowego. W związku z tym mam pytanie: Co jest powodem takiego rozwiązania? Dziękuję serdecznie. Pani poseł Małgorzata Pępek z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Zapraszam serdecznie panią poseł. Wysoka Izbo! Dobrze, że ta ustawa jest wiążąca z sieciami europejskich kolei. Niemniej jednak chciałabym zapytać. Czy tu nie popełniono błędu?

Dziękuję serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Maska opada.

Dlaczego rząd oszukuje Polaków? Dlaczego rząd przedstawia nierealny projekt, który przewiduje budowę szprych, które będą kolejami dużych prędkości, kiedy przyjmuje jednocześnie w dniu dzisiejszym projekt ustawy, który eliminuje szanse na realizację tego projektu w praktyce? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marek Dyduch, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Dziękuję. Pan poseł Przemysław Koperski, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Dlaczego w tej siatce nie ma połączenia z Bielsko-Białą, nie ma połączenia z południową częścią województwa śląskiego? To już kolejny raz, kiedy mieszkańcy subregionu południowego województwa śląskiego, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Bielska-Białej są dyskryminowani. Od kilkunastu lat czekamy na rewitalizację linii kolejowej nr 190 między Cieszynem a Bielsko-Białą. Do tej pory nie możemy się doczekać tej rewitalizacji, a teraz kolejny cios: państwo uderzacie w splot słoneczny mieszkańców regionu południowego województwa śląskiego, uniemożliwiając nam dotarcie do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mam nadzieję, że ją otrzymam, ja i mieszkańcy mojego regionu. Dziękuję bardzo uderzonemu w splot słoneczny panu posłowi. Zapraszam panią poseł Henrykę Krzywonos-Strycharską z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam krótkie pytanie. Chciałabym spytać, czy koleje dużych prędkości pojadą do Gdańska z prędkością większą niż 250 km/h. Pan poseł Jan Mosiński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem podziękować za ten bardzo dobry projekt, który będzie realizowany, bo on de facto przybliża wiele miejscowości do tego szybkiego toru komunikowania się nie tylko z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale również z Europą. Mam tylko pytanie: Czy w ramach tego projektu, tych 10 szprych, te stacje, te miejscowości, które będą miejscowościami przelotowymi, ale też przystankami, dworcami, będą utrzymane?

Dziękuję serdecznie. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Andrzeja Bittela.

Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni Państwo! Wysłuchałem dyskusji i pytań. Szczerze mówiąc, jestem. Wiem, jestem koło pana.

Ale wracając do rzeczy, bardzo dziękuję za to ciekawe podejście do ustawy, która wdraża IV pakiet kolejowy, część rynkową, unijną dyrektywę Rady i Parlamentu Europejskiego, która dotyczy rynku, regulacji rynkowych, gwarancji niezależności infrastruktury, zarządcy infrastruktury, badania ekonomiczności relacji, połączeń, przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, wszystkich rzeczy, które się łączą z rynkiem. Ta dyrektywa nie dotyczy kwestii technicznych.

Kropka.

Zresztą parametr 200 km - o tym pewnie pan poseł też wie - został wprowadzony w Parlamencie Europejskim pomiędzy lipcem a październikiem 2016 r. na wniosek posła Sassolego, włoskiego eurodeputowanego z frakcji socjalistycznej, i został przyjęty. Ale do praktyki projektowania linii kolejowej, a następnie układania rozkładu jazdy to nie będzie miało zastosowania. Będzie miało zastosowanie do badania, czy trasa alternatywna i ten ruch komercyjny. Czy regulator zatwierdzi taką relację - do tego będzie miało to zastosowanie, a

Ale będą.

Tyle w zakresie tego, co jest w materiałach związanych z igrekiem.

Możemy taką debatę poprowadzić: Czy lepiej mieć przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną w formule generalnej dyrekcji, czy spółkę akcyjną, która funkcjonuje na rynku akcyjnym, jest bilansowana przez państwo, jest spółką misyjną, ma specjalne znaczenie. jest w specjalny sposób uregulowana w prawie? Możemy dyskutować. Kwestie pracownicze też nie mają.

Pani poseł nie widzi. 360 zdemontowanych linii kolejowych. Pani poseł, mam prośbę, żebyśmy się jeszcze raz umówili w sposób jasny. Jeżeli miałaby pani samochód, który ze względu na to, że nie leje się do niego oleju, płynu chłodniczego i innych niezbędnych substancji, nie pompuje koła, przestaje funkcjonować, to.

Natomiast nie należało dopuścić do podejmowania decyzji o likwidacji linii kolejowej. Jeżeli to odróżnimy, to argument o tym, że rząd demontuje, likwiduje linie kolejowe. Tak, fizycznie trzeba rozebrać wyeksploatowany, nikomu do niczego niepotrzebny, niemożliwy do ponownego użycia tor kolejowy, trzeba go rozebrać. Ale utrzymać to, o czym rozmawialiśmy przy innej ustawie, przy ustawie Kolej+, tzn. korytarz nieruchomości, żeby go nie zabudować, żeby go nie przerwać, żeby później dzięki temu można było odtworzyć linię kolejową. Nie przy użyciu tych materiałów czy torów sprzed 50 lat, bo one raczej do tego w dzisiejszych czasach nie posłużą.

Dlaczego nie uruchamiamy?

Nie bardzo wiem, o jakich 196 liniach kolejowych mówił pan poseł Szczepański w kontekście CPK i Ostrowa Wielkopolskiego. Jest koncepcja.

Cieszymy się z tego wzrostu, to jest najlepszy wynik od 20 lat. Oczywiście wiele pracy przed nami, wspólnej, jak zakładam, w tym zakresie.

To pewnie też jest przyczyna, dla której choćby mamy teraz to socjalistyczne podejście do własności państwowej.

Dziękuję serdecznie. W trybie sprostowania, pan poseł Grabarczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja lubię z panem dyskutować. Pan pokochał kolej, i to widać. Ale przyzna pan, że w budżecie na ten rok mamy na inwestycje kolejowe 12 mld, a prawie 10 mld pochodzi z Unii Europejskiej. A przykład Francji, Belgii, Hiszpanii nie jest adekwatny, bo oni już te koleje wybudowali, a nie było wówczas tej definicji, która ogranicza zakres pojęcia przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości. Jeżeli my wpiszemy tę definicję do ustawy i poprosimy o środki na budowę igreka albo którejś z tych szprych, co do których toczymy spór przy innej okazji, to oni powiedzą „nie”, ponieważ wy nie będziecie mogli zrealizować tego celu, nie pojedziecie tam szybciej niż 250 km/h albo nie zachowacie innego parametru, odległości 200 km. Na tym polega spór, który teraz wiedziemy.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówił pan natomiast o tym, żeby być bardziej zaangażowanym. Państwo powinniście być zaangażowani, ponieważ państwo jesteście w rządzie. Ja jestem zaangażowany i mam nadzieję, że mieszkańcy Polski powiedzą wam „dziękuję”, i już za kilka lat, a może kilkanaście miesięcy my będziemy mogli połączyć miasto Bielsko-Biała również z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, sprawozdawca komisji.

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Panie ministrze, ma pan jeszcze 2 minuty. Skorzysta pan z tego, tak? A wracając do rzeczy, powtórzę jeszcze raz. Jeśliby Francja wdrożyła tę dyrektywę, jeśli miałoby to mieć wpływ na ruch i trasowanie pociągów, toby musiała zmienić rozkład jazdy, który w tej chwili obowiązuje.

Kropka. Linia nr 196 jest linią regionalną, więc na pewno przynależy do regionalnego programu operacyjnego właściwego marszałka.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk nr 133) Proszę panią poseł Krystynę Skowrońską o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

To trochę prywaty. Panie ministrze, niech pan pamięta o prywacie pani poseł. To skandal. A przechodząc do projektu, chcę powiedzieć, że w imieniu wnioskodawców mam dużą przyjemność przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zrobiliśmy duży ukłon w ich stronę i wtedy koalicja rządząca zgodziła się na takie rozwiązanie. Chcę powiedzieć, że zmieniając tę ustawę w 2006 r., jeśli chodzi o jej pierwsze przedłożenie, zrobiliśmy wtedy duży krok w stronę takiej sprawiedliwości, że jeżeli w najbliższej rodzinie wspólnie coś się buduje, gromadzi się określony, często może skromny majątek, od którego trzeba po raz drugi płacić podatek, bo przecież jeżeli budujemy dom albo jeżeli.

Chcieliśmy ten błąd naprawić i tu dziękuję pani poseł Krzywonos-Strycharskiej za taką inicjatywę w tamtej kadencji. Przedstawiałam to na posiedzeniu plenarnym Sejmu 16 maja 2019 r. Państwo, o dziwo, przy najbliższej rodzinie zawahali się i powiedzieli, że musicie to bardzo skrupulatnie przeliczyć.

Myśmy to zmienili.

Wtedy państwo mówiliście, pan poseł Janczyk, pamiętam, powiedział, że musi to zostać skonsultowane z rządem.

Bądźcie państwo sprawiedliwi.

Apeluję do wszystkich państwa. Proszę, nie czarujcie nas, nie próbujecie powiedzieć, że w tej sprawie musi się wypowiedzieć rząd. W bardzo wielu sprawach nie wypowiada się rząd.

Henia, my wszyscy ci dziękujemy.

Zróbmy to. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tadeusz Cymański, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rzadko to się dzieje, kiedy mamy takie właśnie ustawy jak ta. Na pewno z domu rodzinnego, na pewno z naszego doświadczenia życiowego, ale również - i chciałbym to podkreślić, wykorzystać tę okazję - z dziedzictwa naszego narodu, kultury, również konfesji.

Oto on: „Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem - i wreszcie te słowa - i by móc ograbiać sieroty” Jednak dbałość o dostrzeżenie najsłabszych w społeczeństwie, a to bez wątpienia sieroty biologiczne, ale również społeczne, to osoby, to dzieci i młodzi ludzie, którzy są w rodzinach zastępczych, którzy są w domach dziecka rodzinnych i innych. Rzeczywiście. Jest tutaj też posłanka z mojego okręgu, pani Henryka Krzywonos, postać historyczna, wiadomo, z jakich powodów. Chcę za to bardzo serdecznie podziękować.

Nie wiem, nie ma mojej znakomitej koleżanki Krystyny Skowrońskiej, ona mogłaby powiedzieć, że jeszcze przed tymi fundamentalnymi zmianami, przed zwolnieniem z podatku spadkowego, ten podatek stanowił kwotę kilkuset milionów. To nie jest potężna sprawa, ale ma ona ogromne znaczenie symboliczne. Może skieruję się bardziej w stronę Lewicy, już nie tej Lewicy - mam nadzieję - kawiorowej, ale tej bardziej socjalnej, społecznej, bo ideologicznie bardzo się różnimy, ale w sprawach społecznych, mam nadzieję, nie. Nie dostrzegliśmy tych sierot i najsłabszych, ale też nie dostrzegliśmy tych najbogatszych.

W ogóle przyjrzenie się jak w lustrze podatkom dochodowym i majątkowym jest dobrą okazją przy tym wspaniałym geście, spóźnionym, dodajmy, w kierunku tych najsłabszych.

40 sekund to już naprawdę czas na pożegnania.

Ten spór będzie się toczył. To nie jest tak.

Jeszcze raz dziękuję rządowi (Dzwonek), mojej formacji i wszystkim, którzy w tej sprawie sobie podadzą ręce. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Uzasadnienie w sprawie zmian ustawowych dotyczących opodatkowania od spadków i darowizn wychowanków zastępczej opieki rodzinnej, druk nr 133. Dziecko w rodzinnym domu dziecka czy w rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne do końca życia. Dlatego też wysoce niesprawiedliwe społecznie jest to, że w przypadku przepisania przez rodzica zastępczego swojego dobytku w formie testamentu lub przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej usamodzielnionemu czy pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna były podopieczny musi odprowadzić podatek od spadków lub darowizn jako osoba obca należąca do trzeciej grupy podatkowej, a więc w pełnej wysokości. Jednocześnie zaznaczam, że dziecko adoptowane czy pasierb nie podlegają temu obowiązkowi podatkowemu. Rodzice czy też opiekunowie zastępczy w rodzinnym domu dziecka powinni więc mieć możliwość darowizn lub testamentowania swoich podopiecznych bez narażania ich na obciążenia podatkowe, na które ich zapewne po prostu nie stać np. w przypadku otrzymania nieruchomości w postaci mieszkania. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wnoszę o przyjęcie przez Sejm zmian ustawowych, które dają prawną możliwość, przy zgodzie obu stron, zaliczenia konkretnego byłego wychowanka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do pierwszej grupy podatkowej w systemie podatkowym, uznając to za sprawiedliwe społecznie dla dzieci wychowywanych w systemie opieki zastępczej.

Przyjęliśmy sześcioro naturalnego rodzeństwa - dzieci, które nie miały szans na adopcję, zostały z nami. Zmieniliśmy im nazwisko, pokazaliśmy, jak funkcjonuje normalna rodzina, nie żałując niczego, mimo że jako rodzina byliśmy posądzani o różne niecne rzeczy, że zarabiamy, że robimy na tym interes. Dzisiaj ten interes nazywa się 500+. Wtedy staraliśmy się naszym dzieciom pokazać, co znaczy inny świat, co znaczy wyjazd za granicę, co znaczy nauczyć się języka, co znaczy poznać... co znaczy dom, co znaczy miłość.

Czasem myślę, że robiłam to jak Korczak. Pracując z rzecznikiem praw dziecka, po prostu zastanawiałam się, czy to było jakimś zwiastunem - to, że te dzieci wzięłam. Przecież jako sygnatariusz porozumień sierpniowych nawet przez chwilę nie myślałam o tym, żeby założyć rodzinę, a jednak tak się stało.

Dlatego też bardzo proszę, bardzo - pomyślcie państwo sercem i pomóżcie nam wszystkim, i mnie, i moim dzieciom, i nie tylko mnie. Powiem o panu, który mnie błaga, bo umiera w Wejherowie, w naszych stronach, i cały czas mówi: Mam wychowanka. Mój wychowanek kończy 18 lat, chciałbym odejść, ale chciałbym mu zostawić mieszkanie. Dlatego proszę w imieniu swoim i moich dzieci, różnych dzieci, i w imieniu tego pana. I bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Wysoka Izbo! Dziękuję za to poruszające wystąpienie pani Henryki Krzywonos, które pokazało, o jak ważnej sprawie decydujemy i jaką niesprawiedliwość uda nam się, wiele na to wskazuje, skutecznie naprawić. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zajmujemy się projektem, który tę niesprawiedliwość może ograniczyć i realnie pomóc tysiącom ludzi, którzy naprawdę szczerze na to wsparcie zasługują. Nie mamy wątpliwości, że polskie państwo powinno ze wszech miar wspierać rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Osoby, które podejmują się trudu wychowywania dzieci w ramach pieczy zastępczej, zasługują na wszelkie wsparcie. W ramach obowiązującego prawa spadkowego te bliskie sobie osoby są traktowane jak ludzie sobie obcy.

Przepisy w tej ustawie są tak sformułowane, że dotyczą dziedziczenia przez dzieci, przez rodziców, a nie w drugą stronę. Jeżeli uznajemy bliską relację osób pozostających w tej relacji rodzica i dziecka będącego w pieczy zastępczej, to warto zadbać o to, żeby to działało także w drugą stronę, żeby realnie traktować te osoby jako osoby bliskie, żeby rodzice zastępczy mogli w tym momencie dziedziczyć po swoich dzieciach, czyli aby absolutnie zrównać tę sytuację z sytuacją, która ma miejsce w przypadku rodzin biologicznych. Chciałbym jeszcze odwołać się do bliskich mi słów, nie ukrywam, posła Tadeusza Cymańskiego. Skoro naprawiamy tę jedną niesprawiedliwość, która jest zawarta w tym, jak wygląda dzisiaj polskie prawo spadkowe, to warto zapamiętać, przypomnieć sobie też o tej drugiej, że polskie prawo spadkowe nie rozróżnia w tym momencie spadków w wysokości 1 tys., 10 tys. czy nawet 50 tys. zł i miliardowych fortun, które są dziedziczone w sposób zupełnie nieopodatkowany. We wszystkich krajach europejskich obowiązują progresywne podatki spadkowe.

To na marginesie tych bardzo potrzebnych zmian, o których dzisiaj rozmawiamy, ale o tym też warto pamiętać. Pamiętajmy, żeby naprawić tę drugą. Raz jeszcze pełna wdzięczność dla inicjatorów tych jakże potrzebnych zmian. Zadbajmy o to, żeby dzieciaki będące w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka nie były dłużej dyskryminowane. Pan poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Szanowni Państwo!

Nawiążę do sformułowań zawartych w uzasadnieniu. W sposób taki bardzo przejrzysty, czytelny, poprawny, określają one cel rozwiązania ustawowego, a więc zwolnienie od podatku tzw. nabycia własności lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia lub darowizny, nabycia przez osoby przebywające w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Oczywiście ten zapis jest konieczny, że darczyńcą lub spadkodawcą była osoba, która tworzyła tę rodzinę zastępczą lub prowadziła rodzinny dom dziecka.

One przychodzą może późno, ale lepiej późno niż wcale. Dobrze, żebyśmy mieli tego typu sytuacji więcej. Bardzo proszę, pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poseł Cymański cytował tu Biblię, a przecież nie trzeba tak daleko sięgać w kwestii podatków, wystarczy siódme przykazanie: nie kradnij. O tym właśnie chciałbym powiedzieć, bo oczywiście tę ustawę trzeba poprzeć i trzeba w tym drobnym wycinku znieść ten absurdalny podatek od spadków i darowizn, ale sama idea podatku od spadków i darowizn jest absurdalna. Jak można w ogóle było wpaść na to, że w momencie, kiedy jakaś osoba wręcza coś drugiej osobie, np. umierająca osoba decyduje się na przekazanie czegoś drugiej osobie, albo nieumierająca, po prostu osoba chce przekazać coś cennego drugiej osobie, to państwo kładzie na to łapę i pobiera haracz? Jak można coś takiego robić? A jak działa to w praktyce? W praktyce działa to tak, że jeżeli dam bliskiej osobie z potrzeby serca coś cennego, to ta osoba za to, że przyjęła tę cenną rzecz, musi zapłacić państwu opłatę za przyjęcie prezentu. Za pół roku, jak ta osoba się odwdzięczy i da mi coś cennego, to ja za to, że przyjmuję ten prezent, muszę zapłacić państwu opłatę za to, że przyjąłem ten prezent.

Najlepiej trzymać swój garnuszek i nikomu nie dawać, bo będzie wam zabrane. Bo będzie wam zabrane. Weźmy wesela, śluby. W Polsce pary ślubne są ścigane przez urzędy skarbowe zupełnie serio.

No bo prawo prawem, prawda? To jest sytuacja istotna ekonomicznie. Ludzie się składają w tej sytuacji istotnej ekonomicznie dla pary, żeby miała dobry start, a później ta para przez następne kilkadziesiąt lat życia chodzi na dziesiątki wesel i tak naprawdę ten kredyt, który dostała w istotnym ekonomicznie momencie, oddaje w prezentach. To, że ludzie sobie wzajemnie pomagają w ramach tradycji, jaką jest dawanie sobie finansowych prezentów na weselach, jest za każdym razem opodatkowywane przez państwo. Pary weselne rzeczywiście są ścigane. Oczywiście trzeba znieść podatek od spadków i darowizn. Oczywiście trzeba go znieść. Również na weselach.

On się nazywa „zeznanie podatkowe” Co oznacza to słowo? Zeznaje w Polsce przestępca albo świadek przestępstwa. Ludzie w Polsce są z góry traktowani jak potencjalni przestępcy, bo coś zarobili albo coś dostali. Tak jesteśmy w Polsce traktowani przez aparat fiskalny. Wynika to moim zdaniem z tego, co powoduje zresztą, że Lewica z PiS-em często w sprawach gospodarczych głosują razem. Powiedział tak: Możemy sobie tak szczerze powiedzieć, że ta myśl, robotnicza myśl socjalistyczna, jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Tak naprawdę fundamentem tego projektu ustawy jest wrażliwość, serce i miłość, ale także cudowne, jakże bogate doświadczenia jego pomysłodawczyni pani poseł Henryki Krzywonos. Cieszę się, że mogłem współpracować przy powstawaniu tego projektu. To dla mnie duży zaszczyt.

Cieszę się, że ten projekt uzyskał aprobatę każdej ze stron. Być może (Dzwonek) będzie to projekt, który otworzy następne furtki i bramy do wspólnych osiągnięć legislacyjnych, które będą nie tylko efektem sukcesu tej sali. Przede wszystkim beneficjentami będą Polacy. W procesie opiniowania tego projektu Związek Powiatów Polskich zadał pytanie, czy wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie mogliby też być beneficjentami tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Odpowiem panu posłowi Dzikowskiemu wtedy, kiedy będę zabierać głos jako osoba reprezentująca wnioskodawców. Dzisiaj mam pytanie do rządu. Pomimo deklaracji całej sali plenarnej, przedstawicieli wszystkich klubów liczyć się będzie państwa stanowisko. Ja nie mówię o Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich - miasta i powiaty, samorządy są beneficjentami tego podatku - tylko o stanowisku państwa. Straciliśmy już trochę czasu w zakresie przedłożenia w 2006 r. i pominięcia tej grupy w ubiegłym roku. Może to było przypadkiem. Ale dzisiaj oczekujemy na pozytywne stanowisko i poprosiłabym, aby to padło w dzisiejszej debacie. Dziękuję. Pani poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam prośbę. Chciałam podziękować moim kolegom i koleżankom za ciepłe słowa, ale mam pytanie: Czy możemy przyspieszyć zakończenie prac nad tą ustawą ze względu na tego pana z Wejherowa, żeby miał jeszcze szansę obdarowania swojego wychowanka, którego od początku jego życia wychowywał, wychowuje do dzisiaj? Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Dlatego uważam, że wychowankowie powinni mieć taką samą możliwość jak dzieci biologiczne lub pasierbowie. Należą się ogromne wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich zastępczych rodzin i to one same powinny decydować o swoim majątku, o tym, komu go przekażą, ale ich dzieci, wychowankowie nie mogą być dyskryminowani i karani podatkiem. Panie Pośle Cymański! Jestem w Sejmie trzecią kadencję i po raz pierwszy zgadzam się z panem posłem. Czekam na wspólne pozytywne głosowanie i bardzo dziękuję za taką pozytywną wypowiedź. Dziękuję również mojej koleżance z ławy sejmowej Henryce Krzywonos za tę ustawę. Bardzo proszę, pan poseł Romuald Ajchler, Lewica. Wysoka Izbo! Zwracam się do autorki, pani Krzywonos. Wielkie dzięki, w imieniu wszystkich dzieci, które tutaj pani zaprezentowała przede wszystkim po to, aby one nie musiały płacić podatków, bo jak wiemy, jest wiele podmiotów zwolnionych od podatku od darowizn. Ale mam propozycję, bowiem ta ustawa. Mam wątpliwości, bo jeśli chodzi o niektóre sprawy, można by było je poprawić. Jest wniosek o przejście do drugiego czytania, ale jeśliby nie dało się, pani marszałek, tego pogodzić, to mam propozycję dla pani. Otóż mogłaby pani wyznaczyć termin złożenia sprawozdania, jeśli takowe byłoby konieczne, aby na bieżącym posiedzeniu tę ustawę uchwalić.

Pan poseł Michał Szczerba. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nieodżałowana prof. Maria Łopatkowa mówiła o pedagogice serca, o tym, że dzieci, młodzież potrzebują miłości, przynależności i bezpieczeństwa. I to, co dzisiaj zaproponowała pani posłanka Henryka Krzywonos wraz z klubem Koalicji Obywatelskiej, jest to właśnie również zaspokojenie tej potrzeby bezpieczeństwa.

Ale również trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest projekt zgłaszany po raz pierwszy.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Ministerstwo Finansów ocenia projekt pozytywnie zarówno ze względu na cel, jak i ze względu na adresatów zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie jednak ze względu na pewne nieścisłości zawarte w projekcie konieczne będzie uściślenie niektórych jego przepisów podczas dalszych prac parlamentarnych, w tym uwzględnienie podniesionych uwag dotyczących dziedziczenia przez rodziców po dzieciach wychowanych w ramach pieczy zastępczej. W temacie przyspieszenia prac prowadzonych tutaj, na forum Sejmu, deklarujemy wsparcie i gotowość do pomocy przy odpowiedniej zmianie przepisów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przedstawiciel wnioskodawców pani poseł Krystyna Skowrońska. W imieniu serca, które było wnioskodawcą tego przedłożenia. Na jej osobistym przykładzie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda to podzielenie, rozwiązanie: rodziny biologiczne - pierwsza grupa podatkowa, dzieci i rodzice z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych. Każde nasze osobiste doświadczenie, które służy dobremu rozwiązaniu w przepisach, jest ze wszech miar słuszne.

Nie będę mówić o szkodzie z ubiegłej kadencji dla rozwiązania tego problemu. Jesteśmy w nowej sytuacji, jest ta deklaracja. Chciałabym opowiedzieć i odpowiedzieć państwu posłom na postawione pytania. Dlaczego w tym projekcie nie znalazły się rozwiązania dotyczące wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych? Tam nie ma rodziców. A zatem jeżeli chcemy nawiązać do tej symetrii pierwszej grupy podatkowej, to tylko proponujemy. Odpowiadając koledze z Lewicy, rozwiązaliśmy to w ten sposób, że ten projekt będzie działał zarówno w stosunku do dzieci, jak i do rodziców. Poprzedni projekt takiego kompleksowego rozwiązania nie miał. Ten miał, ale jeżeli będą jakiekolwiek potrzeby doprecyzowania, jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi.

W sprawie związanej z placówkami czy wychowankami z placówek opiekuńczo-wychowawczych - to jest odpowiedź na pytanie pana posła Waldy Dzikowskiego. Mówiliśmy o terminie - pan poseł Ajchler powiedział o korzyściach płynących z tej ustawy i wyznaczeniu terminu.

W tej sytuacji incydentalnie, jeżelibyśmy się zgodzili i nie byłoby protestów związanych z wejściem w życie, jesteśmy skłonni, aby w przepisach przejściowych uregulować, że działa od 1 stycznia br. Jesteśmy w stanie złożyć poprawkę, która wychodziłaby naprzeciw, w przepisach przejściowych, intertemporalnych. Chcę przypomnieć, że ustawa o podatku od spadków i darowizn pokazała jeden element: udokumentowany sposób przekazania darowizny, udokumentowany sposób przekazania spadku. W tym zakresie, jeżeli nawet obyczaje są różne, to mamy po roku 2001 bardzo rygorystyczną ustawę związaną z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

To jest jedyna rzecz, która nas powstrzymywała.

Jeżeli już mówimy o pewnym rozwiązaniu generalnym, to w tym zakresie zgodziliśmy się, że będą to darowizny przekazywane na rachunek, będzie oświadczenie o przyjęciu, będzie przedstawienie urzędowi skarbowemu, że taką darowiznę się otrzymuje, lub taki spadek, że jesteśmy spadkobiercami, chodzi o sporządzenie określonej umowy. Raz jeszcze chciałabym podziękować za tę debatę. To jest krótka, dobrze opracowana ustawa, do której wracamy po raz kolejny. Jeśli zgodzimy się, jeśli taki termin zostanie wyznaczony, to w tym jednym przypadku, sądzę, nikt nie będzie protestował przeciwko temu tempu, do którego przyzwyczailiśmy się w parlamencie. Ta ustawa ze wszech miar zasługuje, żeby nadać jej dobre tempo i czekać na dobre rozwiązanie, a taka była deklaracja pana ministra. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o wyznaczenie przez Sejm terminu przedłożenia sprawozdania. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 32) Proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie uzasadnienia projektu. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

115 tys. osób złożyło ten projekt w 2016 r. Niestety przez opieszałość Sejmu ubiegłej kadencji, przez zamrożenie tego projektu obywatelskiego, nie mogło być dokończone procedowanie nad nim. Te 115 tys. osób, i wiele więcej, które popierają projekt stażowych emerytur, nie doczekało się spełnienia przez Sejm obietnicy poważnego traktowania projektów obywatelskich.

Teraz będziemy dyskutować o emeryturach stażowych. Ten projekt oczywiście, już nawet z racji daty wejścia w życie, która była proponowana, wymaga zmian. Te 4 lata zostały pod tym względem zmarnowane. Nie został ten projekt odrzucony w pierwszym czytaniu, i bardzo dobrze, ale tylko i wyłącznie przez szacunek, mam nadzieję, wszystkich stron do projektów obywatelskich, nie z innych względów. Niestety ci, którzy mówili o poparciu tego, nie chcieli kontynuować. Mam nadzieję, że to się zmieni w tej kadencji, i będziemy robić wszystko, żeby doprowadzić do wprowadzenia emerytur stażowych. Dlatego w uzupełnieniu tego projektu zgłosiliśmy w porozumieniu z OPZZ-em, z reprezentatywną centralą związkową, która zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, nowszy projekt wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniający zmiany, które nastąpiły przez ostatnie 4 lata, uwzględniający uwagi obywateli, które zebraliśmy w czasie nieprocedowania nad projektem obywatelskim, który był zamrożony w ubiegłej kadencji. Dlatego pozwólcie państwo, że będę przedstawiał filozofię emerytur stażowych i mówił o dwóch, a nawet o trzech projektach, bo trzeci projekt dotyczy emerytur rolniczych. Te dwa ostatnie, dotyczące emerytur stażowych i emerytur rolniczych, zostały złożone jako projekty poselskie przez klub Koalicji Polskiej w tej kadencji. Są swoistym uzupełnieniem i wyeliminowaniem niektórych niedociągnięć lub są to zmiany, które były z uwagi na upływający czas konieczne dla tego projektu obywatelskiego. Czyli projekty poselskie, które mam nadzieję będą przedstawione na najbliższych posiedzeniach Sejmu, są jak gdyby kontynuacją projektu „emerytury stażowe” Dlaczego emerytury stażowe i do kogo one są kierowane? Po pierwsze, do tych, którzy ciężko pracują i zaczynają pracę w młodym wieku, zaczynają pracę, i to pracę legalną. To jest jedna z wielkich wartości emerytury stażowej, że zachęca do odprowadzania składek przez pracownika i stwarzania warunków przez pracodawcę, żeby te składki mogły być odprowadzane. Czyli wyciąga z szarej czy czarnej strefy pracowników, których na umowach śmieciowych w ostatnim roku przybyło, samozatrudnionych, na umowach zlecenia.

Od tego momentu nic w tej kwestii się nie działo. A więc bardzo ważne jest zmniejszenie skali zatrudnienia w szarej strefie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest możliwość wyboru dla ciężko pracujących, którzy zaczynają często pracę fizyczną w młodym wieku, kiedy chcą przejść na emeryturę, ale już z zagwarantowanym wyższym świadczeniem emerytalnym niż tylko świadczenie minimalne, bo te okresy składkowe. W tym projekcie ustawy jest mowa o 40 latach dla kobiet i mężczyzn. W projekcie uzupełniającym, który powinien być moim zdaniem wiodącym, to jest 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn, a wiek minimalny, który powinien być wprowadzony, to 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn. To jest również po uwagach, które zgłaszali konstytucjonaliści, zgłaszały różnego rodzaju organizacje, OPZZ się w to wsłuchał.

Jakie będą kolejne pozytywne skutki? Zwiększenie wpływów do budżetu z tego tytułu, że osoby będą się rejestrować, będzie więcej pracy rejestrowanej, będzie wychodzenie z szarej i czarnej strefy, nie będzie zaniżania wynagrodzeń, nie będzie dochodziło do takich sytuacji, bo to się będzie opłacać. Dzisiaj nie tylko wiek emerytalny, a może bardziej często właśnie staż pracy i odprowadzane składki mają ogromny wpływ na wartość późniejszego świadczenia emerytalnego.

To jest też zaczyn do debaty, która powinna się odbyć w trakcie trwania kampanii prezydenckiej. O emeryturach, o emerytach, ale też o młodych, bo ta ustawa jest dla młodych - i tych pracujących, i tych, którzy pracują, dzisiaj zaczęli pracę - jakie będą za chwilę ich obciążenia wobec rodziców i dziadków i kiedy oni będą mogli skorzystać... w ogóle jakie emerytury w Polsce. My mówimy o emeryturze bez podatku. Słyszę, że pan prezydent Duda też planuje złożyć podobny projekt emerytury stażowej. To dobrze. O przyszłości młodego pokolenia, wysokości emerytury - tej dzisiejszej i tej przyszłej - i o obciążeniach, więc taka debata o przyszłości systemu emerytalnego, bezpieczeństwie emerytalnym Polek i Polaków i bezpieczeństwie finansowym młodego pokolenia powinna się odbyć. Debata prezydencka.

Ja do takiej debaty oczywiście jestem gotowy. Ta ustawa jest dobrym zaczynem i dobrym powodem do odbycia takiej debaty. Kolejne pozytywne skutki. Zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków samorządu terytorialnego przeznaczonych na wszelkiego rodzaju pomoc społeczną, bo będzie inny rodzaj zabezpieczenia społecznego tych osób. Ograniczenie kosztów społecznych związanych z zapobieganiem wzrostowi liczby osób wykluczonych społecznie, czyli też te pozytywne skutki nie tylko dla pojedynczych, poszczególnych osób, dla ubezpieczonych, ale również bardzo pozytywne skutki dla wspólnot. Dla wspólnoty samorządowej, która odpowiada, która jest dzisiaj bardzo mocno finansowo drenowana.

Nigdy w historii tyle nie było dokładane.

To są ekonomiczne, pozytywne skutki dla budżetu państwa, dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli też dla tych wszystkich, którzy będą korzystać z usług zdrowotnych, a to są w dużej części osoby w wieku dostojnym, w wieku dojrzałym. Trzeba poważnej dyskusji o systemie emerytalnym i o daniu możliwości wyboru. Ten staż pracy dzisiaj w niezwykle precyzyjny sposób oddaje nasz wkład w cały system zabezpieczenia społecznego. Bez tego, bez myślenia o tym trudno będzie dzisiaj zaproponować lepsze rozwiązania. I to, co się wydarzy pewnie w najbliższych tygodniach, będzie miało bardzo ważne znaczenie, jak do tego podejdzie większość rządząca. Macie państwo większość w Sejmie. Ja gwarantuję, że w Senacie to przeprowadzimy, jeżeli przegłosujecie to w Sejmie. Proszę być spokojnym, ta ustawa uzyska akceptację Senatu. Dopilnuję tego i będę zabiegał o poparcie wszystkich senatorów. Musicie tylko przegłosować i pochylić się naprawdę. Jeszcze o ustawie dotyczącej rolników, bo ta ustawa obywatelska zawiera odniesienie również do emerytur rolniczych. Te dwie nowe złożone ustawy są podzielone: to jest ustawa dotycząca ubezpieczonych w ZUS-ie i tych, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie. I tu proponujemy nie tylko możliwość przejścia na emeryturę po wprowadzeniu 30 lat składkowych, tak jak jest dzisiaj, tylko wracamy do tego wieku, który był, 55 i 60 lat, do 2018 r., ale usuwamy jedną przesłankę, czego potrzebę zgłaszali ubezpieczeni rolnicy, gospodarze na spotkaniach nie tylko w ostatniej kampanii parlamentarnej. To przesłanka dotycząca przekazania lub pozbycia się gospodarstwa.

A więc trzeba dać im szansę, tak jak przedsiębiorcom, którzy mogą pobierać świadczenie emerytalne i prowadzić dalej działalność gospodarczą. Trzeba dać szansę ubezpieczonym w KRUS-ie na prowadzenie działalności rolniczej i pobieranie emerytury.

Drodzy Państwo! Zachęcam do merytorycznej dyskusji, z szacunkiem dla 115 tys. obywateli, którzy od 4 lat oczekują na realizację tego projektu. Dziękuję tym wszystkim, którzy zbierali podpisy, którzy się podpisali. Będziemy drążyć ten temat, i poprzez kolejne inicjatywy poselskie, a jak trzeba, to już niedługo powtórzymy inicjatywę obywatelską. To jest naszym zdaniem najsilniejsza ustawa, od zawsze zgłaszana w Wysokiej Izbie, bo nie dość że potwierdzona wkładem pracy wielu, którzy zbierają podpisy, potwierdzona bardzo dużym poparciem społecznym, to jeszcze dobrze przepracowana. To jest czas bardzo efektywnie wykorzystany. My to powtórzymy.

To ma głęboki sens. Myślę, że to też jest warte odnotowania, bo ma swoje przełożenie na realną dyskusję nad projektem w tym wypadku emerytury stażowej.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam honor w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 32. Przyznam, że z dość mocno mieszanymi uczuciami dzisiaj zabieram głos w sprawie tej ustawy. Idea kryterium stażowego przy emeryturze jest mi bardzo bliska, podobnie zresztą jak „Solidarności” od wielu lat.

Wówczas Jarosław Kaczyński zapewnił, że będzie uwzględniony ten postulat, ale z uwagi na program wówczas mieliśmy nieco inne, bardziej doniosłe priorytety, przede wszystkim kwestię obniżki wieku emerytalnego.

Natomiast deklaracja ta brzmiała tak, że czasem w miarę realizacji innych postulatów, obniżki wieku, 500+ wrócimy do tego. Pewną wzmiankę zrobił tutaj pan poseł Kosiniak-Kamysz. Rozmowy trwają, zobaczymy, co z tego wyniknie.

Chciałoby się powiedzieć, że z przyjemnością odkrywam w panu ludzkie cechy, żałuję, że tak późno się one objawiają, dopiero jak jest pan w opozycji. A więc, wracając do tej sprawy. Przywoływał pan tu kwestię stu kilkunastu tysięcy osób podpisanych pod tym projektem ustawy.

Nie wiem, czy udana. Niewiele czasu mi zostało. Być może w tych zmianach, poprawkach te sprawy są zmienione, ale kryterium 40 lat stażu wyłącznie składkowego wydaje się wręcz niekonstytucyjne.

Chodzi również o te osoby, które ze względu na proces kształcenia trafiły do systemu ubezpieczeń społecznych później, dopiero po zakończeniu nauki. Kwestia szacunków skutków finansowych. Założenie, że jedynie co czwarty uprawniony, jak jest w tej ustawie, skorzysta z tego uprawnienia, jest zupełnie bezpodstawne. Doświadczenia ZUS-u pokazują, że z reguły ponad 80% uprawnionych korzysta z tego uprawnienia, kiedy nabywają oni prawa emerytalne. Również kwestia nieuwzględnienia w tym szacunku kosztów - wspominał tu pan o art. 1 pkt 6 i 7 - podnoszenia emerytury do wysokości emerytury minimalnej ze środków budżetu państwa w momencie, kiedy nie wynika to z wyliczonej wysokości emerytury, jest też ułomnością i na pewno powoduje niedoszacowanie kosztów tej ustawy.

Pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt w swym założeniu dotyczył wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób, które posiadały co najmniej 40 lat okresu składkowego. Natomiast on dobrze pokazuje stosunek partii rządzącej do obywateli: zakrywamy oczy, zamykamy uszy i udajemy, że głosu tych ponad 100 tys. obywateli nie ma. Ale on jest.

Nie tylko przy okazji kampanii wyborczych, czy to prezydenckich, czy jakichkolwiek innych, nawet z tej mównicy ciągle powtarzane jest: jest kampania, rozmawiajmy. Rozmawiajmy o przyszłości, także mojego pokolenia, które perspektywy na emeryturę ma bardzo niewielkie. Spójrzmy na całość: na system emerytalny, na starzejące się społeczeństwo, na rynek pracy, na aktywność zawodową i na bierność zawodową. Jak sprawić, by osoby, które mają prawa emerytalne, chciały być aktywne zawodowo? Jak sprawić, by emerytury były nie tyle szybkie, ile przede wszystkim godne i by pozwalały żyć? Jak sprawić, żeby przyszłość emerytów za kilkanaście, kilkadziesiąt lat była rzeczywiście dobra, a nie tylko symboliczna? I to jest problem. Jak sprawić, by osoby z doświadczeniem, ale osiągające wiek emerytalny, chciały zostać na rynku pracy? To pytanie państwu stawiam, ponieważ doświadczenia pokazują, że gdy obniżamy wiek emerytalny albo gdy jest możliwość przejścia na emeryturę, ludzie na emeryturę po prostu przechodzą. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. W ciągu dekady liczba osób w wieku 50+ wzrosła dwukrotnie. Dziura w systemie emerytalnym jest ogromna, brakuje systemu, który zachęcałby do aktywności zawodowej i do pozostania na rynku pracy. Już teraz emeryci w Polsce mają miliardy złotych długów. Główny powód? Leki, rehabilitacja, prywatne leczenie. Prawie jedenastokrotnie zwiększyła się liczba osób, które pobierają nowosystemową emeryturę, w ciągu ostatnich lat, od 2011 r. do 2019 r. Na koniec grudnia 2019 r. 260 tys. osób pobierało emeryturę nowosystemową, która jest niższa niż najniższa emerytura w Polsce. Już teraz tylko ok. 56% osób jest aktywnych zawodowo. W przypadku kobiet jest to nieco ponad 48%. Stopa zastąpienia kształtuje się na poziomie ok. 50%, za lat 20 będzie wynosić zaledwie 30%. A więc pojawia się dramatyczny problem: z czego emeryci będą żyli? W perspektywie kilkunastu lat te niskie wskaźniki aktywności zawodowej oznaczają mniej pieniędzy dla systemu emerytalnego, mniej pieniędzy do budżetu, więcej pieniędzy wydawanych z systemu świadczeń społecznych, w dłuższej perspektywie kryzys systemu emerytalnego i budżetowego. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w ZUS: teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji, w 2045 r. to będzie 32%, w 2060 r. - 24,9%. Badania jasno pokazują, że kobiety w Polsce chcą pracować, ale są często nieaktywne zawodowo, ponieważ brakuje instytucjonalnej opieki nad dziećmi, ponieważ nie opłaca się podejmować pracy, jeśli wiąże się to z utratą różnego rodzaju benefitów i zasiłków. Te kobiety pobierają emeryturę średnio o 30% niższą niż pozostałe.

Właściwie nazwę to wprost: to jest kradzież, kradzież pieniędzy Polaków z ubezpieczeń emerytalnych. Tak Polaków nie można okradać. Dlatego Polacy nie wierzą w system emerytalny w Polsce i nie ufają państwu. Państwo nic nie robicie, żeby to naprawić. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Kotula, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność prezentować dzisiaj stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy wobec obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającego kryterium 40-letniego stażu pracy umożliwiającego przejście na emeryturę bez osiągnięcia wymaganego wieku. Dodatkowo Konfederacja Lewiatan zgadza się, że potrzebna jest debata o emeryturach stażowych. Należy mieć jednak na uwadze, że głównym ryzykiem związanym z wprowadzeniem obecnego projektu jest obniżenie wysokości emerytur osób przechodzących na emeryturę na podstawie kryterium stażowego w porównaniu z wysokością ich emerytur, gdyby przeszły na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie zmienia to oczywiście faktu, że emerytury stażowe są potrzebne i powinny być obecne jako jedna z możliwych opcji w polskim systemie emerytalnym. Jest to szansa dla osób, które weszły na rynek pracy stosunkowo wcześnie, tj. w wieku kilkunastu lat, po skończonej szkole zawodowej. W przeważającej mierze dotyczy to przecież pracowników fizycznych. W przeciwieństwie do osób mających ukończone studia i pracujących umysłowo jest to też grupa, która jest często mocno wypracowana, a także grupa, która według statystyk żyje krócej. Jest to niestety równoznaczne z tym, że emerytury te będą po prostu bardzo niskie. Wydaje się, że doprecyzowania i dopracowania w ramach debaty o systemie emerytalnym w Polsce, która jest bardzo potrzebna, wymagają pytania o to, co miałoby się wliczać do stażu pracy w przypadku emerytur stażowych. Czy będziemy brać pod uwagę tylko okresy składkowe, czy także te nieskładkowe, bo według proponowanego dziś projektu są to tylko okresy składkowe. Dodatkowo składki te muszą być odprowadzane od minimum najniższego wynagrodzenia. I myślę, że warto przytoczyć tu przykład z Niemiec. Emerytury stażowe zostały tam wprowadzone w roku 2012. Ta opcja przysługuje po osiągnięciu 45 lat pracy i ukończeniu odpowiedniego wieku emerytalnego. Ale do stażu pracy zalicza się zarówno okresy obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia, czas kształcenia się w szkole średniej lub wyższej oraz czas, co bardzo ważne, opieki nad dzieckiem. Prawo do emerytury stażowej jest w Niemczech masowo wykorzystywane przez ubezpieczonych, a ubieganie się o emeryturę stażową nie ma charakteru wyjątkowego, lecz powszechny. Przykładowo w 2018 r. liczba nowo przyznanych emerytur regularnych z tytułu osiągnięcia wieku wynosiła 340 tys., podczas gdy emerytur wcześniejszych, stażowych przyznano aż 240 tys. Być może należałoby rozważyć część tych rozwiązań w polskim systemie, szczególnie wliczenie do stażu pracy opieki nad dzieckiem, co pozwoli polepszyć nam sytuację kobiet. W kolejce do procedowania czeka projekt poselski PSL-u. Czekamy też na projekt prezydenta Dudy, którego założeń co prawda jeszcze nie znamy, ale można z całą pewnością stwierdzić, że proponowane w nim rozwiązania będą przecież podobne. Lewica też przedstawi swój program emerytur stażowych, z tą różnicą, że Lewica nie będzie czarowała rzeczywistości, udając, że rozwiązania w takiej formie są wystarczające. Emerytury stażowe bez gwarantowanej emerytury minimalnej na poziomie minimum 1600 zł netto to właściwie gwarancja emerytur głodowych, szczególnie w przypadku kobiet. Sytuacja polskich emerytów jest zła, sytuacja kobiet na emeryturze jest często dramatyczna. Wielu polskich emerytów nie stać na zakup pełnowartościowej żywności, opłacenie rachunku za prąd, wykupienie leków czy odłożenie na prywatną wizytę u lekarza, bo termin proponowany przez publiczną ochronę zdrowia w obecnym kształcie jest tak odległy, że obawiają się często, że po prostu nie dożyją. Nie można dłużej łatać polskiego systemu emerytalnego, który jest dziurawy jak sitko, jakimiś rozwiązaniami ad hoc.

W Polsce w tej chwili mamy różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn w granicach 20%. Pamiętajmy, że od poborów wynagrodzeń są odprowadzane składki, więc różnica 20% w wynagrodzeniach to różnica 20% w składkach. Kobiety korzystają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Oczywiście od kilku lat są to urlopy płatne składkowo i państwo pokrywa za kobiety składki podczas urlopu. Pamiętajmy jednak, że kiedy mężczyzna zarabia w tym samym czasie normalną pensję i odprowadza składki, składki kobiet odprowadzane od zasiłku macierzyńskiego to nie jest 100-procentowa pensja. W Polsce to kobiety najczęściej opiekują się dziećmi, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami podczas choroby, ale nie tylko. Te okresy często są przecież okresami nieskładkowymi. Przypomnę, że w 2019 r. ponad 250 tys. osób pobierało świadczenie poniżej 1100 zł brutto, tj. ok. 800 zł na rękę. Proszę sobie wyobrazić, jak za to przeżyć. Ubóstwo polskich emerytów rośnie, a nie maleje. 85% najuboższych emerytów to kobiety. Nie możemy proponować rozwiązań, które tylko pogłębią te różnice. Musimy szukać rozwiązań, które pozwolą nie tylko zakopać te rowy nierówności, ale przede wszystkim nie wpędzą polskich seniorów i polskich seniorek w jeszcze większą biedę i jeszcze niższe emerytury, szczególnie jeśli chodzi o kobiety. My jako Lewica poszukujemy rozwiązań, które umożliwią.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Każdy by chciał, żeby tak było.

Boicie się zrobić coś dobrego? Sam pan mówił, że go popieracie.

To rozwiązanie nie burzy systemu.

To nie jest obligo.

To będzie niższe świadczenie, wiec będzie to mniejsze obciążenie dla systemu ubezpieczeń społecznych. Musimy mieć tę świadomość. Takich rozwiązań należy szukać. Ono dzisiaj wychodzi naprzeciw temu.

Ci, którzy doczekają - pewnie niektórzy nie doczekają. To jest sprytny sposób. Kadencja, ten sam projekt. Nie będziemy powtarzać tego samego, bo nawet niektórzy posłowie doszli już do wniosku, że pewne elementy się zdezaktualizowały.

Więc to jest ten dramat, o którym mówimy.

Chwała za to, wprowadziliście to bardzo dobre rozwiązanie.

Też trzeba się nad tym zastanowić, też złożymy taką propozycję.

To nie jest pomysł ani mój, ani prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, tylko to ludzie zgłaszają. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jeżeli nie, zamykam listę.

Wysoka Izbo! Podstawowym zadaniem systemu emerytalnego w Polsce jest zapewnienie obywatelom świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepracowanych lat pracy dopuszczonych ustawą, a także świadczeń ubezpieczeniowych dla osób, które nie mogą świadczyć pracy ze względu na stan zdrowia. Obecna ustawa nie spełnia, szanowni państwo, oczekiwań społecznych, stąd projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 100 tys. osób. Obywatele chcą, aby mogli decydować, czy po przepracowaniu 40 lat pracy chcą zostać na rynku pracy, czy chcą przejść na emeryturę. Obywatele chcą decydować o tym, jaka jest wielkość odprowadzanych składek, ile zgromadzili kapitału początkowego i jak jest on waloryzowany. Należy jednak zadać pytanie, szanowni państwo, jaka będzie ta emerytura, bo jeśli ma być to niska, głodowa emerytura, to nie ma na to zgody. Po 40 latach pracy każdy obywatel powinien mieć godną emeryturę, bo na to zasłużył. Pan poseł Bogusław Sonik, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówimy o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczywiście jest godne zastanowienia, dlaczego dopiero teraz przy robieniu tych remanentów wracamy do tego. Od początku VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej było 20 aktów prawnych zmieniających tę ustawę o emeryturach i rentach. Największe zmiany dotyczyły obniżenia wieku emerytalnego, trzynastej emerytury czy planowanego przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Może warto byłoby teraz rozważyć rzeczywiście rezygnację z opodatkowania emerytur. Te środki przecież były już i tak objęte podatkiem dochodowym.

Nie ma pani poseł? Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak, to dobre rozwiązanie. Ale emerytury stażowe bez emerytury minimalnej? Już nie tak dobre. Przede wszystkim dotyczy to kobiet. Nie chcemy emerytur głodowych, nie chcemy dramatycznych historii o tym, że osoby starsze muszą wybierać między lekami a ogrzewaniem czy wykupieniem jedzenia. W przypadku tej dyskusji, dyskusji o emeryturach, dyskusji o emeryturach stażowych, musimy też zacząć rozmawiać o jednym aspekcie: o pracy kobiet, pracy opiekuńczej, opiece nad dziećmi, oczywiście, ale także opiece nad osobami starszymi, osobami zależnymi, rodzicami, dziadkami. To bardzo często kobiety muszą rezygnować z pracy zawodowej, bo system opieki nad osobami starszymi jest niewydolny. Wtedy to kobiety biorą na siebie ten ciężar.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Temat emerytur jest dość obszerny. Za kilkanaście lat, za 25 lat to będzie 20% ostatniego uposażenia.

Musi być nasz wspólny pomysł, jak rozwiązać te problemy. Czy pracujecie nad jakimś systemem?

To już widać w dniu (Dzwonek) dzisiejszym - malejąca siła nabywcza tych świadczeń itd. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szkoda tych 4 lat, które ten projekt obywatelski przeleżał, bo przez te 4 lata mogliśmy wspólnie, ponad podziałami w istotny sposób poprawić byt polskich emerytów, zbudować racjonalny system, a tak ten czas minął, panie ministrze. W tym czasie serwowaliście państwo różne pomysły i poza takim doraźnym rozwiązaniem jak trzynasta emerytura niewiele tego było.

Pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ubóstwo emerytek i emerytów jest hańbą dla polskiego państwa. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wnosi rozwiązania bez określenia wymaganego wieku.

Pytam o to z troski, by kolejne osoby nie popadły w ubóstwo, będąc w okresie jesieni życia. Dlatego też zachęcam do dyskusji nad tym projektem, również w kontekście zadanych przeze mnie pytań. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Romuald Ajchler, Lewica. Wysoka Izbo!

Zwracam się do pana ministra Szweda. Zresztą to jest stara sprawa. To jakimś sposobem nie wyszło, ale co niektórzy myślą, że warto by było wrócić do tej sprawy, bowiem tragedia emerytów zaczyna się wówczas, kiedy jeden z emerytów - czy rencistów - odchodzi, pozostawiając drugą osobę z wielkimi sprawami dotyczącymi wydatków, a przecież wydatki, np. na utrzymanie (Dzwonek) mieszkania, dwóch czy trzech mieszkań, są te same. Na pewno będzie to kolejna inicjatywa obywatelska, jeśli tego nie zrobicie. Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica. Wysoka Izbo! Przedłożony obywatelski projekt ustawy proponuje potrzebne rozwiązanie, ale obarczony jest ryzykiem zmniejszenia wysokości świadczeń emerytalnych i pogłębiania się nierówności w wysokości świadczeń dla mężczyzn i kobiet. Pokazuje to po raz kolejny, jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie emerytury minimalnej, równej dla kobiet i mężczyzn.

Jak bardzo pogłębią się nierówności między świadczeniami dla kobiet i mężczyzn? Na koniec: Czy wiadomo, czy zbadano, jak dużą liczbę osób obejmie ta emerytura i w konsekwencji ile osób odejdzie z rynku pracy? Ile z tych osób to będą kobiety? Jak to wpłynie na rynek pracy? Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To ważny projekt obywatelski, poruszający kwestię, o której rozmawiamy w tej Izbie od wielu lat. Chciałem przypomnieć, że w 2012 r. w tej Izbie był rozpatrywany projekt obywatelski: 35 lat, 40 lat, emerytury stażowe, wniesiony przez OPZZ, przez Jana Guza.

Wówczas odrzucono te wszystkie projekty.

Wysoka Izbo! Mógłbym przy okazji tego projektu powiedzieć, że tak naprawdę temat mnie nie dotyczy, bo już dawno straciłem nadzieję, że z ZUS-u jakakolwiek złotówka wpłynie na moje konto, kiedy osiągnę wiek emerytalny. Problem jest w tym, że cały czas udajemy, że ZUS jest wydolny, że on będzie jeszcze działał. Możemy w niego pompować krew, możemy w niego pompować tlen, możemy nad nim się modlić, ale on nie wstanie. Trzeba po prostu zreformować system emerytalny.

Otrzymaliście ogromny mandat zaufania od Polaków - macie samodzielną większość, macie 4 lata, żeby zreformować system emerytalny. Może na początek zacznijmy od tego projektu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Dyduch, Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Kiedyś, pamiętam, był taki system emerytalny, że alternatywnie można było pracować: 65 lat - mężczyzna, 60 lat - kobieta, albo 40 lat stażu pracy lub 35 lat stażu pracy. Wtedy było wiadomo, że jak pracuje się systematycznie 40 lat, to cały czas do systemu idzie składka. A dzisiaj mamy taką sytuację, że młodym nie opłaca się pracować, pracują po trzydziestce. Pracują 30 lat, dwadzieścia parę i czekają na wiek emerytalny. Czy te 40 lat pracy i płacenia składki, czy niechęć do pracy i później te dwadzieścia parę lat?

Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. W takim razie bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda.

Wysoka Izbo!

On faktycznie jest już z poprzedniej kadencji, ale problem jest nam doskonale znany, bo przecież o tych sprawach emerytalnych mówimy od lat. Ja bym powiedział, panie pośle, że szkoda tych 8 lat w koalicji z Platformą Obywatelską, gdzie jedynym waszym rozwiązaniem, które zaproponowaliście, było podniesienie wieku emerytalnego. Druga kwestia jest taka, panie przewodniczący, że będzie pan miał problem z ustaleniem w klubie PSL-Kukiz jednolitego stanowiska, bo jeżeli pana kolega mówi, że ZUS jest trupem i do niczego się nie nadaje, to absolutnie z taką tezą nie można się zgodzić, bo ZUS jest dzisiaj jedynym możliwym, że tak powiem, ośrodkiem, gdzie są wypłacane emerytury, i ma się dobrze. I nie ma tutaj dzisiaj żadnego zagrożenia co do wypłat emerytur. Przypomnę, że w tym roku FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego są wypłacane emerytury, to jest 262 mld zł. W ostatnim okresie ponad 60 mld zł przybyło do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z racji dobrej sytuacji gospodarczej, niskiego bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń. Takie wypowiedzi tylko szkodzą tej debacie, bo one powodują, że ktoś, kto przysłuchuje się naszej debacie, będzie myślał, że jest jakieś zagrożenie. Nie ma żadnego zagrożenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma się dobrze, a gwarantem tak jak w innych państwach jest budżet państwa, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Ale co do zasady jesteśmy oczywiście tutaj otwarci na dyskusję, na debatę, bo tak myślę, i pan przewodniczący też o tym mówił, że sam projekt w tej postaci jest nie do zaakceptowania z prostej przyczyny - on powstawał w zupełnie innej sytuacji. Po podniesieniu wieku emerytalnego państwo próbowaliście znaleźć jakieś rozwiązanie dotyczące właśnie wprowadzenia emerytur stażowych.

Tak że ta wersja projektu jest dzisiaj już nie do zaakceptowania z racji upływu czasu i zmian, które wprowadziliśmy, czyli chodzi o przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet - 60 lat i mężczyzn - 65 lat.

Ponad 50 tys. osób z tego skorzystało. Osób, które w ogóle nie miały wypracowanego stażu, jest trochę mniej niż połowa, a w przypadku reszty jest dopłata do minimalnego świadczenia.

Pan przewodniczący Janusz Śniadek doskonale pamięta również decyzje komisji krajowej „Solidarność” dotyczące stażu. Dzisiaj w debacie, powiedziałbym, kandydatów na prezydenta też ten temat jest aktualny, ale nam potrzeba całościowej debaty nad systemem ubezpieczeń, w którym też mieści się kwestia związana z elementem stażowym i na to jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Rozmawiamy o projekcie obywatelskim. To też z tej okazji skorzystam, żeby powiedzieć o innej akcji obywatelskiej, z uwagi na to, że bohaterowie tej akcji są dzisiaj na galerii w Sejmie. Kilka tygodni temu OSP w Porębie Spytkowskiej - to jest miejscowość w gminie Brzesko, w Małopolsce - ochotnicza straż pożarna zaproponowała zbiórkę na rzecz płonącej Australii, tych dramatów, które się tam dzieją, tej krzywdy, która niestety wyrządzona na przyrodzie na wiele, wiele lat pozostanie. I młodzi ludzie z OSP razem z prezesem Krzysztofem Rachwałem, z komendantem i prezesem, z Adrianem Zaleśnym, z Moniką Adamczyk, którzy są na sali, to są młodzi ludzie z OSP. dzisiaj wspólnie z Wojciechem Podlesiem, pułkownikiem Państwowej Straży Pożarnej, i burmistrzem miasta i gminy Brzesko Tomaszem Latochą przekazali 422 tys. na rzecz ratowania przyrody w Australii, na Park Narodowy im. Kościuszki. Więc dla nas to jest naprawdę bardzo symboliczne - na fundację parków narodowych i dzikiej przyrody. To jest przykład skuteczności obywatelskiej. Dziękujemy za to, co robicie. To jest przykład pięknej akcji obywatelskiej. A teraz wróćmy do tematu, o którym rozmawialiśmy. Dziękuję wszystkim za głosy. Myślałem, że unikniemy tych uszczypliwości historycznych, ale skoro nie uniknęliśmy. A to teraz, panie pośle, z wielkim szacunkiem i sympatią do pana, powiem szczerze, do pana posła Śniadka, za jego historię, za pana historię.

Byli jej posłami, byli wojewodami, byli ministrami? No byli. PiS jest spadkobiercą AWS-u. PiS jest spadkobiercą AWS-u i też wtedy rządziliście. Kto wtedy sprywatyzował cukrownie? Kto doprowadził do prywatyzacji banków i PZU? Kto wprowadził patologiczny system OFE, który zjadał 10% prowizji na starcie. Zbudowaliście giganty międzynarodowej finansjery, ale nie polskiego emeryta. To było za waszych rządów. Chcecie takiej debaty? Proszę bardzo, każdą decyzję rządu AWS-u, każdą decyzję rządu. No nie wiem, czy z nich jesteście dumni, bo to były rządy z Romanem Giertychem i z Samoobroną. Pamiętacie, że byliście z Romanem Giertychem w koalicji? Tak jest po drugiej stronie. A wie pani, ja lubię wszystkich, bo pani poseł mówi, że ja kogoś nie lubię. Ja lubię ludzi, tym się może też różnimy. Ja lubię, panią też lubię. Nie ma naprawdę. Chcecie takich debat? Chcecie mówienia, ile z OFE wytransferowano pieniędzy do międzynarodowych korporacji? Kto to wprowadzał? Kto wprowadzał chaos w służbie zdrowia? Kto sprywatyzował górnictwo? Naprawdę, dramaty na Śląsku. Bezrobocie strukturalne. Czemu w 2004 r. tyle osób wyjechało za granicę po wejściu do Unii Europejskiej? Bo rządy AWS-u to było gigantyczne bezrobocie strukturalne, które spowodowaliście. Ja się swojej przeszłości. Nie, to jest przykład, który pan, panie pośle, wywołał. Ja mogę wchodzić, bo ja nie ukrywam swoich działań. Nie wszystko się udało. Ja potrafię powiedzieć: małe niedociągnięcie. Ale dużo się udało, bo np. po waszych rządach ile wynosił urlop macierzyński? 18 tygodni. A po naszych 52. Chodźmy do przodu, bo ta ustawa jest do przodu, nie o polityce historycznej. Ona jest o przyszłości, o tym, co przed nami. Wszyscy poparliście, zgoda. Trzeba pracować nad tym projektem razem z tymi innymi, które są. Połączmy je - i to jest prośba do was. Też do pana ministra, żeby na to wpłynął.

Popracujmy nad tymi projektami. Wiele było pytań, jak to wpłynie na wysokość emerytury. No właśnie wkład, zaangażowanie w staż, odprowadzanie składek to jest dzisiaj zaangażowanie i ma największy wpływ na wartość przyszłej emerytury. Emerytura minimalna jest dzisiaj w Polsce. Jest emerytura minimalna i ona jest równa dla kobiet i mężczyzn, ona nie jest uzależniona od płci w żaden sposób. O matkach 4+ - my poparliśmy ten projekt, bo on był potrzebny. To prawda, bardzo dobrze. Ale on też wprowadził pewną niesprawiedliwość. Przychodzi mama, która mówi: Urodziłam piątkę dzieci i poszłam do pracy. Pracowałam przez 25 lat i odprowadzałam składki.

Dobrze, że jest zabezpieczenie dla matek 4+, dla tych, które nie pracowały, które nie wypracowały emerytury, bo nie mogły, bo nie były w stanie pogodzić życia zawodowego z życiem rodzinnym. To wszystko jest więc do zrobienia, tylko trzeba dobrej woli i poważnej debaty o przyszłości. Nie będziemy mieli problemu z uzgodnieniem stanowiska. Wielkim entuzjastą podniesienia wieku emerytalnego był - chyba pewnie jest dalej - pan premier Jarosław Gowin. Macie też różnice w tej sprawie w Zjednoczonej Prawicy. Martwcie się o siebie, my się będziemy martwić o siebie. Damy sobie radę, wy pewnie też będziecie jakoś się starali. Jest wiele do zrobienia w tej kwestii. Dzięki, że nikt nie zgłosił wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Ale jak ten projekt przeleży kolejne 4 lata i będzie czytany po raz kolejny w kolejnym Sejmie, to za 8 lat w tym projekcie nie będzie już nic aktualnego. Wiele osób po prostu czeka na te emerytury stażowe. Zróbmy jedną wspólną podkomisję. O to wnoszę w imieniu 115 tys. obywateli, bo dzisiaj występuję w roli przede wszystkim przedstawiciela inicjatywy obywatelskiej, podjętej w celu wprowadzenia emerytur stażowych, inicjatywy, która już 4 lata czeka na wdrożenie. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 32, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 35) Proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Tomasza Dybka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Jeżeli jest już pan gotowy, to bardzo proszę.

Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! W 2017 r. zebraliśmy ćwierć miliona podpisów pod projektem obywatelskim ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Usiedliśmy przy jednym stole: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności, elektroradiolodzy, psycholodzy. Porozumieliśmy się. Najważniejszą rzeczą po tylu latach jest to, że wszyscy przy jednym stole doszliśmy do wspólnego konsensusu. 19 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie. Ale oczywiście strona rządowa przekazała: Czego wy chcecie, jak my już mamy swoją ustawę? Mamy ustawę, która została napisana i przeprocedowana w 36 godzin, 7, 8 czerwca 2017 r. 19 lipca 2017 r. z tego miejsca zapowiedziałem protest głodowy w imieniu rezydentów i Porozumienia Zawodów Medycznych. Stało się.

Skończyło się, jak się skończyło. Został zmieniony minister.

Podczas protestu głodowego zebraliśmy 150 tys. podpisów pod kolejnym projektem obywatelskim dotyczącym wzrostu nakładów na ochronę zdrowa. Dzień po procedowaniu, czyli po pierwszym czytaniu w Sejmie, pan minister podpisał z Porozumieniem Rezydentów porozumienie w sprawie wzrostu nakładów, a więc bardzo szybko zostało przykryte to, co było zrobione przez obywateli, czyli to, że zebraliśmy 150 tys. kolejnych podpisów w ciągu 2 tygodni. W 2018 r. zaczęła obowiązywać sławetna ustawa rządowa po raz pierwszy, historyczna chwila.

Są wymyślone wskaźniki, jest średnia odnoszona do 3900 zł brutto.

To nie była podwyżka, to była typowa regulacja, która potęguje biedę.

Wiadomo, pielęgniarki mają swoją regulację prawną, lekarze mają swoją regulację prawną, ale, jak państwo chyba dobrze wiecie, bo każdy korzystał z państwowej służby zdrowia, w placówkach medycznych nie tylko jest lekarz i pielęgniarka, jest fizjoterapeuta, drugi zawód - 65 tys. osób jest uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - diagnosta. Bez dobrej diagnostyki co państwo zrobicie?

Oczywiście każdy obywatel posłucha, bo przychodzi minister i to mówi.

Nie dostali żadnej podwyżki. Ludzie są przemęczeni, ludzie pracują na dwóch, trzech etatach po to, żeby normalnie funkcjonować.

To jest 2300 zł, 2400 zł, 2500 zł brutto.

Tak to dzisiaj wygląda. Idziemy dalej.

A ludzie są odsyłani z kwitkiem, nie ma dostępu do fizjoterapeutów, do diagnostyki. Dwudziestego pierwszego mamy protest głodowy. Oczywiście bardzo szybko ministerstwo przyjeżdża na głodówkę, nie można głodować: ale wiecie, będziemy, jest ustawa, będzie procedowane, przestańcie, usiądźmy do rozmów. Siadamy do rozmów. To 680 mln będzie, ale pan minister mówi: Wiecie, co wam powiem? Mówiąc językiem kolokwialnym, dostaniecie lepsze pieniądze. W 2019 r. zostaje odmrożona kwota i naprawdę przekaz informacji z ministerstwa czy ze strony rządzącej jest bulwersujący dla zwykłego obywatela, bo mówią, że 4200 zł, że została zwiększona kwota bazowa.

To nie jest kwota, którą zarabia fizjoterapeuta, to nie jest kwota, którą zarabia diagnosta.

2847 zł minus minimalna pensja, która była w 2019 r., daje nam 597 zł.

Rodzi się pytanie, po co się kształci w Polsce tych ludzi. Po to, żeby wyjeżdżali na Zachód? Po to, żeby pracowali w dyskontach? jest brutalna prawda. Pracujcie państwo 14 godzin dziennie. Jakie się popełnia potem błędy? Kto wie. Ale to była propaganda sukcesu: tak, zwiększyliśmy kwotę bazową do 4200 zł. Oni jeszcze protestują? Kolejne spotkania z panem ministrem, 4 mld zł zostało przekazane po raz pierwszy, historyczna chwila.

Mówimy o fizjoterapeutach, diagnostach, psychologach, elektroradiologach. Czy dana placówka przekazała grupie zawodowej dane pieniądze? Proszę państwa, poświęciłem 2 miesiące na to, żeby pojeździć sobie prywatnie i posłuchać tego.

Tyle zarabiają. I taki dyrektor mówi: nie, nie mam pieniędzy, nie ma rozporządzenia, to, co powiedział minister, nie do końca jest prawdą, mamy zadłużenie szpitali, mamy zadłużenie.

Niektórym rzeczywiście udało się uzyskać kwotę, ale dam przykład Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”

Kursy są dzisiaj bardzo kosztowne.

Oni muszą. Już nie będę pokazywał niektórym posłankom i posłom, którzy są dyrektorami w placówkach, jak oni z nami rozmawiają, bo to nie jest godne człowieka. To nie jest godne człowieka, jak oni z ludźmi rozmawiają, ze swoimi podwładnymi. Szanowni Państwo!

Dopóki nie zabraknie.

Ja rozumiem. Nie może być dysproporcji, proszę pani.

Pracują przy tym samym pacjencie. Nie może tak być. Nie można dzielić.

Sprawa jest bardzo prosta. Nie ma rozwiązań systemowych, jest potęgowana bieda.

Po co zwiększać wskaźniki? Macie ustawę.

Szanowni Państwo!

Nie zapomnijcie o nas, a my damy w pewnym sensie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Pani Minister! Wysoka Izbo! Przedmiotem obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, druk nr 35, jest określenie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz trybu przyznawania wynagrodzenia. Już na wstępie należy zauważyć, że tytuł projektu ustawy nie oddaje jej faktycznego zakresu, błędnie sugerując, że ustawa reguluje kwestie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, podczas gdy wprowadza ona przepisy ustanawiające najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wątpliwości konstytucyjne budzi określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Wprowadzenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyższego od powszechnej płacy minimalnej dla grupy osób wyodrębnionej jedynie ze względu na miejsce zatrudnienia wydaje się nieuzasadnione i może być uznane za sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2005 r. - sygnatura akt K 31/03 - różnicowanie sytuacji podmiotów podobnych jest dopuszczalne, jeżeli zostały dochowane trzy wymogi: po pierwsze, wprowadzone przez ustawodawcę kryteria różnicowania muszą być racjonalnie uzasadnione i muszą mieć związek z celem i treścią przepisów, w których zawarta jest dana norma, po drugie, waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie podmiotów podobnych, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów podobnych, i po trzecie, różnicowanie podmiotów podobnych musi znajdować podstawę w wartościach, zasadach lub normach konstytucyjnych. W naszej ocenie powyższe wymogi nie zostaną spełnione w przypadku wyodrębnienia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych w stosunku do zatrudnionych w innych podmiotach. Charakter pracy osób, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych i są zatrudnione w podmiotach leczniczych wyłącznie w ramach ich obsługi, jak np. kadra administracyjna czy pracownicy gospodarczy, nie różni się w żaden istotny sposób od charakteru pracy osób wykonujących analogiczne funkcje w innych podmiotach. W projekcie pojawiają się niestety - nie będę tutaj ich wytykać, ale niestety jest ich dosyć dużo - błędy legislacyjne.

Należy zauważyć, że projekt reguluje analogiczne kwestie, co ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r. i była już dwukrotnie nowelizowana w ramach realizowania postulatów zgłoszonych przez związek zawodowy reprezentujący pracowników ochrony zdrowia.

Jednym z efektów podjętych w 2018 r. rozmów była nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. dotycząca sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która podniosła kwotę bazową z 3900 zł do 4200 zł. Przyspieszyło to tempo podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników ochrony zdrowia.

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Rajmund Miller, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej wobec obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, druk nr 35. Proszę państwa, 250 tys. podpisów pod tym projektem. To świadczy o tym, że sprawa jest bardzo poważna. Słyszymy z ust rządzących, że trwają rozmowy. Proszę państwa, 5 lat już trwają te rozmowy, a ludzie mają głodowe pensje, tak jak mówił przedstawiciel pracowników sektora medycznego. Ciągle słyszymy o tym, że rozmawia się osobno z pielęgniarkami, osobno z rezydentami, osobno z innymi grupami. Natomiast ten projekt w sposób bardzo logiczny przedstawia nam sposób ustawiania wynagrodzeń w sektorze medycznym. Fatalna reforma szpitali i sieci szpitali - która doprowadziła do tego, że naprawdę nie są pokrywane realne koszty procedur medycznych, tylko wynagrodzenia są ryczałtowe - spowodowała, że najłatwiejszym elementem, na którym dyrektor może zaoszczędzić, są zarobki pracowników. Więc z czego dyrektorzy zabierają? Zabierają z wynagrodzenia pracowników, bo nie ma stałej zasady wynagradzania. I ta ustawa proponuje nam minimalną kwotę wynagrodzenia i bardzo logiczne przeliczniki, czyli ta minimalna kwota wynagrodzenia będzie przeliczana zgodnie z wykształceniem, z miejscem zatrudnienia wszystkich pracowników w resorcie służby zdrowia, począwszy od pracowników technicznych, przez analityków, fizjoterapeutów, a skończywszy na lekarzach. To jest projekt ustawy, który wreszcie spowoduje, że minister nie będzie jedną decyzją po to, żeby załagodzić konflikty, dzisiaj obiecywał rezydentom, jutro pielęgniarkom, pojutrze komuś innemu. Dlatego jako klub Koalicji Obywatelskiej będziemy popierali tę ustawę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Zdzisław Wolski, klub Lewica.

Ten projekt ustawy, ustawy obywatelskiej, to krzyk rozpaczy. Wielki krzyk rozpaczy pracowników podmiotów leczniczych, którzy to przez rząd byli i są traktowani po macoszemu. Wymagania wzrastają, płace iluzorycznie. To ćwierć miliona podpisów pracowników.

To są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych, farmaceuci, ratownicy medyczni, technicy medyczni, elektroradiolodzy, psychologowie, dietetycy, logopedzi. Ta kolejność nie jest moja, tylko tak jest w projekcie ustawy, tak że ja tu nie chciałbym absolutnie różnicować. Rząd w poprzedniej kadencji, a również i w tej ograniczał się do polityki gaszenia pożarów, bo co chwilę te pożary wybuchały. Pamiętamy wszyscy: a to pielęgniarki, a to fizjoterapeuci, a to ratownicy medyczni.

Czyli były proponowane i były przyjmowane różne ustawy, czasami rozporządzenia, w sposób bardzo nieuczciwy, bo pielęgniarki zaczęły nieco więcej zarabiać.

Czyli głęboko niedofinansowane szpitale, przychodnie - w zasadzie każda placówka, każdy podmiot leczniczy finansowany przez fundusz zdrowia - coraz bardziej się dusiły. Te 14 mld, którymi - mam wrażenie - rząd się w ogóle nie przejmuje. To zadłużenie będzie wzrastało. Rząd lekceważył służbę zdrowia, lekceważył pracowników. Pracownicy słyszeli, że przecież gospodarka kwitnie, mamy deszcz pieniędzy, wszystko idzie w dobrą stronę, tylko jakoś nie w służbie zdrowia. Ja tylko tak informacyjnie. Owszem, były przyjmowane ustawy, były nowelizowane. Kwota bazowa z czerwca 2017 r. to było 3200.

Potem są mnożniki, to jest procedura dochodzenia do zakładanych pensji, proponowana w ustawach, która zwiększa to o 20%, nie mniej niż 20% rocznie. Docelowo pod koniec roku przyszłego ma zarabiać aż 3345 zł. Ratownik medyczny - również. Pracownik działalności podstawowej - też ma swoją ważną rolę - aktualnie zarabia 2436 zł, czyli poniżej minimalnej płacy obowiązującej w gospodarce.

Jak my ich zachęcamy?

Ale jak oni mogą być zadowoleni? Owszem, ale dotyczy to wąziutkiej grupy tych, którzy mają powyżej 40 lat, mają specjalizację i tyrają - sylwestry, Wigilia. Biorą mnóstwo dyżurów, bo nawet jakby ich nie chcieli brać, to są sytuacje szantażu emocjonalnego, bo kolega, ordynator, dyrektor prosi: Weź chociaż ze trzy dyżury, bo inaczej będę musiał oddział zamknąć. Taki jest real. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Wysoka Izbo!

Służba zdrowia potrzebuje naszej pomocy. Pomocy, którą cechować będzie zgoda ponadpartyjna: od prawa do lewa polskiej sceny politycznej. Sprawy zdrowia Polek i Polaków powinny być dla nas absolutnym priorytetem, ponieważ życie ludzkie nie ma ceny i nie można go przedkładać ponad żadną inną rzecz - materialną czy niematerialną. Szkoda, że w Polsce tak mało rozmawiamy o potrzebach pracowników ochrony zdrowia. On ma na celu przede wszystkim chęć poprawy sytuacji w polskiej służbie zdrowia, służbie, która wymaga dofinansowania, doinwestowania, wyższych pensji dla jej pracowników, nowego sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób. Jednak dobrze, że ten temat w ogóle został podniesiony, ponieważ to właśnie od nas zależy kierunek, w którym pójdzie rozwój naszej ochrony zdrowia. Jako klub uważamy projekt obywatelski za potrzebny i słuszny. Ustawa określa sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznawania wynagrodzenia w sposób, który uznajemy za godny. Wyrażamy szacunek do wykonywanego zawodu. Dzięki temu projektowi ustawy mamy szansę zatrzymać wciąż postępującą emigrację pracowników ochrony zdrowia w poszukiwaniu lepszych warunków pracy. Rośnie płaca minimalna, ale wraz z nią w zastraszającym tempie rośnie również inflacja. Za chwilę może się okazać, że propozycje najniższych podwyżek, które przedstawi minister zdrowia, nie przystają do bieżącej rzeczywistości i nie są żadnym sensownym rozwiązaniem. Wynagrodzenia w polskiej służbie zdrowia powinny być wysokie, bo Polki i Polacy zasługują na dobrą opiekę medyczną, zasługują na to, by ludzie, którzy się nimi opiekują, nie musieli się martwić, czy wystarczy im od pierwszego do pierwszego. Poczucie stabilności i bezpieczeństwa związane z lepszym wynagrodzeniem przełoży się na lepszy standard pracy, a właśnie do tego powinniśmy dążyć. Osiągnąć to możemy tylko poprzez ponadpartyjne porozumienie.

To jest bardzo dobry projekt. Rzeczywiście siedliście i ustaliliście, jak to powinno wyglądać. Pani Minister!

Oni powiedzieli jasno, że wiedza lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, wszystkich związanych z ochroną zdrowia jest na poziomie europejskim, a nawet, powiedziałbym, światowym, ale leczenie odbywa się na poziomie powiatowym. Tak usłyszałem od młodych ludzi, którzy chcą się kształcić, którzy chcą zdobywać wiedzę. Jak oni za swoje małe pensje mogą odbywać te szkolenia, kiedy pracodawca nie chce dokładać jeszcze do tych szkoleń? Jest deklaracja, że to zostanie skierowane do dalszych prac w komisjach. Bardzo się cieszę, że ta deklaracja padła, ale chciałbym też, żeby za tą deklaracją poszło procedowanie tej ustawy.

Jeśli te płace będą na tym poziomie, na jakim są dzisiaj, to rzeczywiści ci młodzi ludzie wyjadą za granicę i będzie coraz gorzej z naszą ochroną zdrowia. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Tuduj, klub Konfederacja, koło, tylko koło. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia zawiera propozycje zmian w kwestii finansowania pracowników wykonujących zawody medyczne. Projekt ten jest wyrazem stanu świadomości i postulatów szeroko rozumianego środowiska medycznego, ale niestety przeleżał w Sejmowej zamrażarce ponad 2 lata, jak słyszymy. Bez wątpienia obecnie obowiązujące współczynniki pracy zarówno w kwestii ilości pracowników zawodów medycznych, jak i w kwestii ich wynagradzania nie są adekwatne do odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Jako uwagę natury ogólnej należy odnotować, że w krajach Zachodu zasadnicza pensja medyka zaczyna się w okolicy 1,5 średniej krajowej. W Polsce natomiast według aktualnego prawa jest to ok. 0,64 średniej krajowej, a więc niewiele ponad płacę minimalną. W konsekwencji żenująco niski poziom wynagrodzeń w tym sektorze jest zasadniczą przyczyną odpływu naszych kadr medycznych za granicę. Rząd po raz kolejny próbuje wybrnąć z trudnej sytuacji półśrodkami. Na bieżącym posiedzeniu miało się odbyć głosowanie nad nowelizacją o zawodzie lekarza i lekarza dentysty otwierającą jeszcze szerzej polski rynek pracy na imigrację, m.in. z Dalekiego Wschodu i Afryki. Miała ona wprowadzić ekspresową procedurę nostryfikacji zagranicznych dyplomów wyrobionych poza Unią Europejską. Proces taki skutkowałby obniżeniem jakości leczenia i tym samym mógł narazić na szwank życie i zdrowie polskich pacjentów. Warto przypomnieć, że od lat kształcimy w Polsce bardzo wielu obcokrajowców i oni i tak po ukończeniu studiów w większości wybierają wyjazd za granicę, tak samo byłoby po nostryfikacji dyplomów medycznych imigrantów z Azji i Afryki. Alarmujemy, że już za 5 lat blisko połowa z 200 tys. polskich pielęgniarek przekroczy granicę wieku emerytalnego. A nawet dziś w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców mamy zaledwie 5 pielęgniarek. Średnio w Unii Europejskiej jest ich 8, przy czym w Szwecji, Niemczech średnio po 10, a kraje takie jak Szwajcaria, Dania i Norwegia mają aż 15 pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców. W przeddzień wielkiego kryzysu w zawodach medycznych musimy powiedzieć Polakom prawdę: w Polsce postępuje zapaść kadrowa, a w perspektywie dekady nawet 1/3 szpitali może zostać zamknięta właśnie z powodu braku kadr medycznych. Wobec tak dramatycznej sytuacji zdiagnozujmy, że to sam system opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje uzdrowienia. Trzeba upowszechnić zawody personelu pomocniczego, opiekunów medycznych i asystentów. Należy obudować zawód lekarza personelem, który odciąży go od biurokracji, i tę biurokrację maksymalnie ograniczyć. Należy też urealnić koszty procedur medycznych, zreformować system rozliczania świadczeń przez NFZ i doprowadzić w ten sposób do maksymalnego wykorzystania drogiego sprzętu diagnostycznego i leczniczego znajdującego się w szpitalach. Należy wreszcie, o czym dzisiaj mowa, zmienić tabelkę płac i współczynniki pracy na bardziej przejrzyste, sprawiedliwe i dostosowane do aktualnych warunków ekonomicznych. Mamy nadzieję, że ustalenie satysfakcjonującej siatki płac dla wszystkich zawodów medycznych wyhamuje exodus polskich specjalistów kształconych w Polsce, exodus, wyjazdy za granicę. Koło Poselskie Konfederacja będzie głosowało za skierowaniem projektu obywatelskiego do dalszych prac. Przedstawimy równocześnie własne poprawki opracowane przez zaplecze społeczne Konfederacji zatrudnione w zawodach medycznych. Dziękuję. Do pytań zgłosiło się 15 pań i panów posłów. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Dobrze. Musimy zdążyć przed głosowaniami. Będę przestrzegać dyscypliny czasu, jak zawsze. Nie ma pani poseł.

Wysoka Izbo! Jestem posłem z Podkarpacia, gdzie zapaść służby zdrowia widoczna jest na każdym kroku, jak w soczewce wszystkie problemy służby zdrowia skupiają się właśnie na Podkarpaciu. A służba zdrowia bez ludzi, bez personelu medycznego to tylko mury i nieużyteczne maszyny. Aby tego personelu nie zabrakło, by nie wyemigrował za lepszym życiem, konieczne jest uporządkowanie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w ochronie zdrowia. Dlatego wzywam do poparcia tego projektu społecznego i jednocześnie zwracam się z pytaniem do pana premiera i do każdego z posłów PiS-u: Czy zagłosujecie za bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków, czy też ponownie stwierdzicie, że nie ma na to środków, a jednocześnie za chwilę na tej sali lekką ręką będziecie próbowali przeznaczyć 2 mld zł, które wyciągnęliście z kieszeni Polaków, na przemysł propagandy, uosabiany dzisiaj przez jednego z waszych polityków, który kieruje telewizją zwaną rządową? Innych określeń ze względu na szacunek dla tej Izby nie będę przytaczał. Pan poseł Waldy Dzikowski, również klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy, w którym proponuje się zmianę wynagrodzeń w zawodach medycznych, wymaga dalszego procedowania nie tylko ze względu na to, że jest projektem obywatelskim. Ma ciekawe, innowacyjne rozwiązania, które są realne do wdrożenia w życie w obecnym czasie.

Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, również klub Lewicy. Również nie ma. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy pochodzi od środowisk wykonujących zawody medyczne. Mamy katastrofalną sytuację demograficzną w tej grupie. Przeciętny wiek pielęgniarki czy pielęgniarza wynosi 50 lat i nieubłagalnie zbliża się do wieku emerytalnego. Pensja lekarza stażysty po ukończeniu ciężkich, wymagających nakładów i wyrzeczeń studiów medycznych jest dziś na granicy poziomu płacy minimalnej. Pensja wielu fizjoterapeutów czy pielęgniarek oscyluje wokół płacy minimalnej. To powoduje odpływ młodych pracowników opieki zdrowotnej do sektora prywatnego i ich emigrację. To powoduje zamykanie oddziałów szpitalnych i całych szpitali. Projekt ustawy, który wymaga dostosowania do aktualnego systemu prawnego, słusznie postuluje, aby w tych jakże odpowiedzialnych i społecznie istotnych zawodach medycznych punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia było przeciętne, a nie minimalne wynagrodzenie. To warunek konieczny, aby w Polsce były osoby gotowe świadczyć opiekę zdrowotną w ramach publicznego (Dzwonek) systemu. Moje pytanie: W jakiej perspektywie czasu możemy spodziewać się podniesienia. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Aleksander Miszalski, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! W sumie podpisało ją 230 tys. osób. Od tego czasu minęły już 33 miesiące, a zgodnie z art. 13 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej mają państwo 3 miesiące na procedowanie nad tą ustawą. Oczywiście co do zasady ustawę popieram, natomiast mam dwa pytania, które zadała nam Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mianowicie: Dlaczego dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją proponowany współczynnik pracy ma wynosić 1,75, podczas gdy dla specjalisty fizjoterapii i diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją - 2,0?

Pan poseł Bogusław Sonik, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Szlachetne zdrowie, Fragment fraszki Jana Kochanowskiego ilustruje nam, jakim problemem jest choroba. Dlatego pracownicy zatrudnieni w ochronie zdrowia powinni być odpowiednio wynagradzani. Po pierwsze, lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia podczas pracy powinni być skupieni tylko na niesieniu pomocy chorym, nie powinni zaprzątać sobie głowy koniecznością szukania dodatkowych źródeł utrzymania. Po drugie, nie możemy sobie pozwolić, by nasi specjaliści, którzy zostali wykształceni w Polsce, których koszty edukacji ponieśliśmy, emigrowali. Dlaczego dopiero w dniu dzisiejszym Wysoka Izba zajmuje się obywatelskim projektem ustawy, który wpłynął do Sejmu w 2017 r.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Romuald Ajchler, klub Lewicy.

Za to państwu bardzo serdecznie dziękuję, a te życzenia kieruję do pani Barbary Mazany i dr. Listopadzkiego ze Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy. Nie tylko dlatego, że tutaj jestem, zabieram głos. Wiem, że resort zdrowia ma problem ze środkami finansowymi. Przekażcie to ministrowi zdrowia.

Zapłaćcie tym ludziom. Dziękuję.

Panie Marszałku! Pani Minister!

Tak jest praktycznie w każdym szpitalu. Mamy ogromne braki kadrowe. Trzeba powiedzieć, że resort robi bardzo niewiele, aby ta sytuacja się zmieniła. W zamian za to nie mogą oczekiwać żadnej gratyfikacji finansowej. Utrzymaliście kontrakty na tym samym poziomie, który był w roku 2019. Nawet złotówki więcej nie dołożyliście. Żeby spłacić te koszty specjalizacji, bo nie refundujecie tego, a izby również tego nie refundują - tak, tak, proszę sobie sprawdzić, jaki odsetek refundujecie - muszą pracować kolejne 13 lat. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W tym projekcie obywatelskim ukazuje się cała bardzo trudna sytuacja w służbie zdrowia, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenie kadry pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych. W lipcu 2018 r. zostało zawarte porozumienie między pielęgniarkami, ministrem zdrowia, pracodawcami i Narodowym Funduszem Zdrowia. Chciałbym zapytać, w jaki sposób jest realizowane to porozumienie.

W bardzo wielu szpitalach, w tym w szpitalach powiatowych, często poszczególne oddziały są. Ten brak kadry medycznej wynika z samego faktu niewystarczającej ilości kadry medycznej, ale z także bardzo niskich płac. Dziękuję. Pan poseł Michał Szczerba, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Pamiętamy, co mówił premier Morawiecki wtedy, kiedy protestowali nauczyciele. Mówił, że nauczyciele pracują mniej niż reszta Polaków, a zarabiać chcą więcej. Teraz dowiedzieliśmy się, Wysoka Izbo, co rząd, co premier w szczególności myśli o zarobkach polskich pielęgniarek. 12 lutego podczas rozmowy transmitowanej na Facebooku został on zapytany, czy przekonałby własną córkę do pozostania w Polsce, gdyby ta zdecydowała się zostać pielęgniarką. Premier odpowiedział: Koszty życia w Polsce w porównaniu do Norwegii czy Londynu są dużo niższe, w związku z tym wynagrodzenia, które są niższe, niestety cały czas niższe, istotnie niższe, one są kompensowane poprzez to, że koszty życia są niższe. To jest wkład pana premiera w wyjaśnienie skandalicznych zarobków medyków, w tym także polskich pielęgniarek. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, szanowni państwo, że w tym roku z zawodu może odejść nawet 60 tys. pielęgniarek. Trzeba bić, szanowni państwo, na alarm.

Wysoka Izbo! Pod względem liczby lekarzy na 1 tys. mieszkańców Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. W 2016 r. Porozumienie Zawodów Medycznych, które było pierwszą tak szeroką inicjatywą przedstawicieli różnych środowisk medycznych, przygotowało dwa projekty ustaw i zebrało pod każdym ponad 100 tys. podpisów. Projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia leży w Sejmie od stycznia 2017 r. Możemy więc zauważyć, jak rząd interesuje się Polakami i ich zdrowiem. Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Wzrost nakładów na zdrowie w rządowej wersji jest niższy i wolniejszy, a widełki płac dużo mniej korzystne. Dlaczego rząd oszczędza (Dzwonek) na zdrowiu Polaków i bagatelizuje problem braków kadrowych? Zagapiłem się, nie zdążyłem przerwać. Pan poseł Radosław Lubczyk, klub PSL. Wysoka Izbo!

Dzisiaj wiemy, że nie zatrzymamy polskich medyków, pracowników ochrony zdrowia w kraju z tak niskimi pensjami.

Czy rzeczywiście deklarujecie, mam nadzieję, że rząd, czy Prawo i Sprawiedliwość, przychyli się do procedowania, że całą grupą przyjdziecie na posiedzenie komisji i będziemy próbowali wypracować jakieś porozumienie, żeby rzeczywiście (Dzwonek) w ochronie zdrowia działo się dużo lepiej?

Panie Marszałku! Dzisiejszy projekt ustawy jest przykładem tego, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje Polaków. Jak traktuje projekty obywatelskie, które trafiają do Sejmu. 200 tys. podpisów złożonych pod projektem ustawy zostało zamrożonych na kilka lat jeszcze w ubiegłej kadencji. Drugi przykład to projekt dotyczący emerytur strażaków - też został zamrożony na kilka lat. Projekt o deputacie węglowym to też kolejnych kilka lat. Dzisiaj mamy do czynienia z projektem, który ma, można powiedzieć, ratować nasze zdrowie i życie, ludzkie życie, bo przecież te pielęgniarki na co dzień stoją przy chorych, sprawują opiekę nad tymi osobami. Ile z tego powodu zamknięto oddziałów w szpitalach?

Wysoka Izbo! Jestem posłem z Lubelszczyzny.

Szanowni Państwo! Jeśli nie dołoży się pieniędzy do służby zdrowia na szpitale, na oddłużenie, na zniesienie limitów, które nie pokrywają faktycznych kosztów, w tym kosztów płac, jeśli nie zadbamy o to, aby godziwie zarabiali lekarze i pielęgniarki, to lekarze, którzy są kształceni w naszym kraju, pielęgniarki również, odpłyną nam za granicę. Co jest ważniejsze od zdrowia i życia obywateli? Czy telewizja publiczna, czy zdrowie? Apeluję do rządu, aby przyjął ustawę i aby dołożył pieniędzy na ustawę, bo nie wystarczy uchwalić ustawy. Ważne jest to, aby znalazły się pieniądze na realizację ustawy (Dzwonek) Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę, pani minister. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie państwu dziękuję za tę troskę o pracowników ochrony zdrowia. Rzeczywiście pracownicy są największym kapitałem. Prawdą jest, że maszyny ani budynki nie stanowią o jakości udzielanych świadczeń, tylko wyłącznie pracownicy, którzy zatrudniani są w podmiotach leczniczych i od których wymagamy wysokich kompetencji. Cieszę się, że wszyscy wspólnie tę dbałość wyrażamy. Chcę zapewnić, że rząd od 2015 r. dostrzega ten problem, który państwo wielokrotnie definiujecie, brak kadr, starzejąca się kadra medyczna. Chcę przypomnieć, że średnia wieku, którą w tej chwili osiągają pielęgniarki czy lekarze, nie nastała z dnia na dzień. Wiedzieliśmy 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu, że następuje katastrofa demograficzna, i dopiero od 2015 r. zaczęliśmy podejmować konkretne działania, aby poprawić sytuację kadrową w Polsce.

Mieliśmy 74 szkoły, w tej chwili mamy 106 szkół. Od 2015 r. zwiększyliśmy o 6 liczbę uczelni, na których kształceni są lekarze. Niestety proces kształcenia tych profesjonalistów trwa długo i te osoby do systemu trafią za kilka bądź kilkanaście lat. Szkoda, że te działania nie były podejmowane odpowiednio wcześnie. Wszyscy państwo wskazujecie na nierówne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, a przede wszystkim na bardzo niskie wynagrodzenia w ochronie zdrowia, więc żebyśmy wiedzieli wszyscy, o czym mówimy, chcę przypomnieć jedno, że my po raz pierwszy w 2017 r. przygotowaliśmy projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To była pierwsza taka regulacja, która wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, w zależności od wykształcenia, od specjalizacji, jakie posiadają, od stanowiska, na którym pracują, gwarantowała minimalne wynagrodzenie. Nie można było zatrudnić pracownika poniżej, co bardzo często się zdarzało wcześniej. Zagwarantowaliśmy minimalne wynagrodzenie uzależnione właśnie od tych wskaźników, o których państwo dzisiaj mówicie.

I te środki do systemu trafiły i trafiają. Ta ustawa ewoluowała. Kolejna zmiana była w 2018 r., kiedy rozszerzyliśmy zakres jej działania, włączyliśmy pracowników, którzy biorą udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, którzy nie byli objęci tą regulacją. A w ubiegłym roku podwyższyliśmy kwotę bazową, czyli to jest gwarancja, że z roku na rok pracownicy ochrony zdrowia mają zagwarantowany przyrost wynagrodzenia. Efekty są różne w różnych grupach zawodowych: w jednych grupach zawodowych ten wzrost był szybszy, w innych wolniejszy.

Systematycznie pracujemy nad tym, żeby zadbać o wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

To my przygotowaliśmy projekt, który pozwala nam teraz realizować wiele zobowiązań m.in. wobec pracowników. Dzięki niemu mamy coraz więcej środków w systemie i możemy finansować te wynagrodzenia.

Widać wyraźnie wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Odnosząc się teraz do projektu obywatelskiego, szanowni państwo, chcę tylko poinformować, że kwestia wynagradzania pracowników ochrony zdrowia jest szeroko dyskutowana - o czym przedstawiciel wnioskodawcy wspomniał - w Radzie Dialogu Społecznego w formule trójstronnej z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, pracodawców i strony rządowej. My rozmawiamy - minister zdrowia spotyka się z poszczególnymi grupami zawodowymi na spotkaniach bilateralnych, jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o dialog społeczny. My nie boimy się tematów, nie boimy się wyzwań. Rozmawiamy i dzięki temu powstają nowe projekty. Szanowni państwo, chcę poinformować, że już jesteśmy na etapie rozmów z Radą Dialogu Społecznego.

Podejmujemy kolejne działania i nadal będziemy poprawiać warunki wynagradzania.

Tak też się stało, w wielu podmiotach leczniczych wprowadzono podwyżki dla fizjoterapeutów, diagnostów, farmaceutów, techników - dla tych pracowników, którzy także są bardzo ważni, jeśli chodzi o udzielanie świadczeń. Niestety część z tych pracodawców do tej pory nie zrealizowała tego przyrzeczenia. Dlatego wspólnie, nawet z panem, który reprezentuje wnioskodawców, na co dzień się spotykamy i rozmawiamy na ten temat, aby wspierać tych pracowników, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem od pracodawcy tychże wynagrodzeń. Tak że mam nadzieję, że te działania, które podejmujemy, będą kontynuowane, że spowodują, że kadry medyczne, które w Polsce są warunkiem dobrego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, będą zatrzymane. Przy okazji chciałabym państwu przekazać informacje, ponieważ w wielu pytaniach się to przejawiało. Kwestia kształcenia podyplomowego, lekarzy, pielęgniarek czy w przypadku innych zawodów medycznych. Oczywiście koszty kształcenia są bardzo wysokie, ale chcę przypomnieć, że to rząd finansuje koszty rezydentur, czyli specjalizowania się lekarzy. Z roku na rok zwiększamy środki na rezydentury. To jest koszt budżetu państwa. Również zwiększamy nakłady na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek. W ubiegłym roku wydaliśmy 8 mln, a w tym roku wydajemy 9 mln na kształcenie podyplomowe. Z roku na rok to wzrasta, aby rzeczywiście przedstawiciele tych zawodów nie musieli z własnych środków finansować szkolenia podyplomowego.

Kolejne grupy zawodowe, bo już kolejne projekty są przygotowane, będą miały taką możliwość, aby wykorzystać płatny urlop szkoleniowy w wysokości 6 dni, żeby mogli spokojnie realizować doskonalenie zawodowe. Myślę, że te działania, o których mówimy, o których powiedziałam, świadczą o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o kadry, ma na celu poprawę ich sytuacji. Z roku na rok podejmujemy działania, żeby coraz więcej środków na finansowanie świadczeń było zabezpieczonych w budżecie państwa. Głos zabierze przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pan Tomasz Dybek. Bardzo proszę.

Państwo Ministrowie! Szanowni Państwo! Odpowiem pani minister w bardzo prosty sposób: bajka, bajka, bajka, propaganda i tylko tyle. To nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Odniosę się do pytań, za które serdecznie dziękuję. Pierwsze z pytań było odnośnie do trybu legislacyjnego, że daty się nie zmieniają.

Szanowni Państwo!

W procesie pisania tego projektu uczestniczyło całe środowisko: pielęgniarki, fizjoterapeuci i lekarze.

Nieładnie, panie pośle. Odsyłam pana, żeby pan przeczytał tę ustawę. Jedną tabelkę wystarczy przeczytać ze zrozumieniem.

Pan chyba reprezentuje swoją grupę.

Panie pielęgniarki uczestniczyły w procesie tworzenia. Mam nadzieję, że pan poseł zrobił to nieświadomie.

Dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, zawarty w druku nr 35, do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 37) Proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Tomasza Dybka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Zebraliśmy 150 tys. podpisów w 2 tygodnie.

Są spekulacje. Czy państwo słyszycie ze strony rządzącej: pacjent, szybki dostęp, opieka nad pacjentem? Oni nie dbają o pacjenta, oni dbają o to, jaka ma być metodologia przeliczania i jaki ma być wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Muszę państwu powiedzieć w bardzo prosty sposób: 6,8% to jest minimum, które musi dane państwo mieć, żeby normalnie funkcjonować. Średnia w Unii Europejskiej jest powyżej 10% produktu krajowego brutto. Już nie wspomnę o takich państwach jak np. Niemcy - 11%, Szwecja.

Bo muszą być odpowiednie środki, odpowiedni nakład, żeby normalnie funkcjonować. Diagnostyka. Oprę się na raporcie takiej instytucji, która się nazywa Najwyższa Izba Kontroli. Nakłady ponoszone na badania laboratoryjne w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. W Polsce diagnostyka laboratoryjna jest niedoceniana, a nakłady w zakresie dostaw wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej na tle krajów Unii Europejskiej są niewielkie i wynoszą: 8,5 euro w Polsce na osobę, natomiast w Słowenii - 23 euro, w Niemczech - 27 euro, w Belgii - 33 euro.

Tak to dziś funkcjonuje, niestety. To jest brutalna rzeczywistość.

Czas oczekiwania - 6, 7 miesięcy. Po udarze to fizjoterapeuta z pacjentem pracuje, logopeda i psycholog. Nie wspomnę o rehabilitacji. Co to jest za rehabilitacja po urazie, jeżeli jest prowadzona za 2 miesiące, 3 miesiące, 5 miesięcy? A przecież konstytucja gwarantuje nam wszystkim dostęp równy do ochrony zdrowia. Szanowni Państwo! Pani minister powiedziała o kształceniu. Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni.

Nie mają urlopu, o którym pani minister mówiła. Ani jednego dnia nie mają urlopu. Trudno tu mówić o frustracji środowiska. My się spotykamy, z tego nic nie wynika, dlatego mamy dość tych bajek.

Ale w pewnym momencie trzeba było sobie powiedzieć: stop, stop, bo my już rządzimy.

To są tylko bajeczki.

Propaganda sukcesu. Mają na umowach po 2100 zł, 2200 zł, 2300 zł. Od tej kwoty liczona jest wysługa lat.

Nie wiem, kto z tego będzie tak szybko korzystał, bo ktoś potrzebuje szybkiej pomocy.

Tam wszystkie środowiska się podpisały. Te środowiska również uczestniczyły w Radzie Dialogu Społecznego i w zespole trójstronnym. Tu i teraz to państwo macie. Podsumowując tę propagandę sukcesu, zacytuję jednego europarlamentarzystę. Jak się okazuje, ten europarlamentarzysta parę dni temu na Twitterze - oczywiście jest ze strony obozu rządzącego - podsumował to w bardzo prosty sposób: W żadnym innym zakresie Polska nie pozostała tak bardzo obrzydliwym państwem i społeczeństwem postkomunistycznym jak w dziedzinie służby zdrowia. Nie mówię tu o wyjątkach, o poszczególnych lekarzach i pielęgniarkach, lecz o całym systemie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwsza w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Violetta Porowska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Deklarowanym celem projektu ustawy jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia poprzez zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2020 nie może być niższa niż 5,2% PKB z roku poprzedniego w 2018 r., do 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r., czyli w obecnym roku. Już tylko te przytoczone założenia pokazują, że projektowana ustawa w szerokim zakresie odnosi się do przeszłości. Co więcej, 1 stycznia 2018 r. weszła w życie - z późniejszymi zmianami - rządowa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która swoim zakresem reguluje m.in. kwestie zawarte w omawianym projekcie obywatelskim ustawy. Warto w tym momencie podkreślić, że rządowe rozwiązania to niespotykany w przeszłości wzrost nakładów na ochronę zdrowia i nie jest to żadna propaganda, tylko fakty. Otóż żaden wcześniejszy rząd, żadna partia wcześniej - poza chlubnym wyjątkiem projektu autorstwa prof. Religi, którego to projektu ani Platforma Obywatelska, ani PSL nie chciały kontynuować - powtórzę raz jeszcze: żaden wcześniejszy rząd nie wziął na siebie odpowiedzialności za regularne, stałe, progresywne, bez względu na koniunkturę gospodarczą coroczne podnoszenie wydatków na ochronę zdrowia. Inni tylko mówili - często nieprawdę - ale to rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie i odpowiedzialnie powoduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia. A teraz fakty. Między rokiem 2015 a 2019 nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 25 mld zł, a tylko na ten rok przewiduje się kolejny znaczący wzrost finansowania ochrony zdrowia, bo aż o 8,5 mld zł.

Mówiąc krótko, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje swoje deklaracje i plany szybciej, niż obiecał. Czy to oznacza, że zadowala nas obecny stan rzeczy w służbie zdrowia? Oczywiście, że nie. Ale trzeba mieć wielce złą wolę, by nie zauważyć tych historycznie wielkich nakładów. Powtórzę jeszcze raz: historycznie wielkich nakładów po raz pierwszy. Dziś możemy obiektywnie stwierdzić, że naprawa polskiego systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia już się odbywa. Chciałoby się powiedzieć - wreszcie. Ale odbudowa polskiej służby zdrowia powinna się odbywać także poprzez wprowadzanie mechanizmów zwiększających efektywność wydatkowania, racjonalizację procesów systemowych. Nad tym powinny dziś toczyć się odpowiedzialne, dalekowzroczne dyskusje. Bezprecedensowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia właśnie się odbywa. Ten kierunek będziemy kontynuować. Dlatego, mimo że obywatelski projekt omawianej ustawy został w większej części wyczerpany, skonsumowany przez rządową ustawę z 2017 r., klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje przekazać projekt do dalszego procedowania w Komisji Zdrowia. Teraz głos zabierze pan poseł Marek Hok, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego w ogóle mówimy o tych kłopotach?

Oczywiście odbyło się pierwsze czytanie.

A doskonale wiemy, że sytuacja, wbrew temu, co mówi pani poseł, pogarszała się praktycznie z miesiąca na miesiąc albo z roku na rok.

Jesteśmy też na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, w Europie. W Austrii jest ponad 5,2, a średnia europejska to jest 3,7 lekarza na 1 tys. mieszkańców.

Gdyby oni jednego dnia złożyli wypowiedzenie, a już byli blisko w związku z receptą elektroniczną, panie ministrze, to system ochrony zdrowia, można powiedzieć, by padł.

I rzeczywiście przychody w związku wprowadzeniem sieci szpitali, dla naszych szpitali, które są w sieci, wzrosły z roku 2017 na 2018 o 13%, ale koszty wzrosły o 17%.

Zadłużenie polskich szpitali w ciągu ostatnich tylko 4 lat powiększyło się o 3 mld. Pani poseł, nie tylko pani poseł mówiła o wielkich nakładach na ochronę zdrowia, o wzroście historycznym. To są pieniądze ze składek, które wynikają z wynagrodzeń, i te środki wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale każda propozycja wzrostu finansowania ochrony zdrowia, w tym przypadku projektu obywatelskiego 6,8, oczywiście będzie popierana przez nasz klub i będziemy za dalszym procedowaniem nad tym projektem. I o to też będę prosił Wysoki Sejm. Pani poseł Marcelina Zawisza, klub Lewicy. Szanowni Państwo! W trakcie kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość obiecywało zmiany w ochronie zdrowia, ponadpartyjny pakt, piątkę Kaczyńskiego. Tej piątki w waszej propozycji budżetu nie widać. Mówiliście też inne rzeczy, że sytuacja w ochronie zdrowia to skutek wieloletnich zaniedbań. Ale co zrobiliście przez ostatnie 5 lat? Prawie nic. Teraz macie drugą kadencję i gdzie jest ten przełom? Od przedstawienia planów Ministerstwa Zdrowia na posiedzeniu komisji odnoszę wrażenie, że ta kadencja też będzie wypełniona pustosłowiem, bo cel Prawa i Sprawiedliwości de facto pozostał taki sam: utrzymać realne nakłady na ochronę zdrowia na tym samym poziomie względem PKB. Średnia w krajach OECD to 6,7% PKB. Więcej, postanowiliście kłamać w tej sprawie, przyjmując kreatywny sposób obliczania nakładów na zdrowie. Niewidziane w świecie. Nakłady liczycie w stosunku do PKB sprzed 2 lat. Jakoś wydatki na wojsko potraficie liczyć do roku bieżącego. O wojsko się troszczycie, a o ludzi już nie. Ale wy nie okłamujecie mnie, Lewicy, nie okłamujecie opozycji. W żywe oczy okłamujecie pacjentki i pacjentów, personel ochrony zdrowia, chorych i umierających. Nie będę mówić, ile czasu ludzie czekają w kolejce, bo my wiemy, ile czekamy w kolejkach. Jak się martwimy o to, czy zdążymy przed pogorszeniem czy śmiercią. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile musimy czekać do lekarza specjalisty czy po prostu na zwykłą wizytę. Diagności, rehabilitantki, pielęgniarki zarabiają grosze, a każdy z tych zawodów musi się na bieżąco szkolić, oczywiście za swoje. Rozmawiałam z fizjoterapeutami, 2 tys. na rękę, koszt szkolenia 20 tys., oczywiście za swoje. A premier? Premier uważa, że skoro w Polsce koszty życia są niskie, to niskie pensje nie są największym problemem świata. Mówi to człowiek, który zarabiał dziesiątki tysięcy miesięcznie. Zamiast pracy w systemie ochrony zdrowia wymagacie wciąż i wciąż heroicznych czynów w imię misji. Personel ma takie hasło, bardzo trafne: powołaniem się nie najem, głosuje nogami i wyjeżdża. Kiedy to w końcu do was dotrze, że ludzie nie będą pracować za grosze? W trakcie kampanii 2015 r. dużo mówiliście o godności pracy. Ludzie, którzy ratują życie naszych dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pracują za głodowe pensje. A podwyżki? Podwyżki widzą wtedy, kiedy podwyższana jest płaca minimalna. Oddziały położnicze w mniejszych miejscowościach są zamykane. Poza dużymi miastami zwija się nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Wydłuża się czas oczekiwania na karetkę. Szpitale mają problemy z organizacją pracy SOR-ów, brakuje kadry, a ludzie umierają w oczekiwaniu na dobrą ochronę zdrowia. To wszystko skutek tego, że nie potraficie kolegom z finansjery powiedzieć: nie, za te pieniądze się nie da. I w efekcie system reformuje się sam, przez rozkład. Nie macie odwagi przyjąć podatku cyfrowego, opodatkować korporacji międzynarodowych i przeznaczyć tych pieniędzy na ochronę zdrowia, bo się ich boicie. Dlatego apelujemy do was: podnieście realnie nakłady na ochronę zdrowia. Te pieniądze pójdą na wynagrodzenia personelu, żeby Polska w końcu przestała eksportować pracowników i pracownice do Niemiec, Holandii czy Czech. Pani poseł mówiła tutaj, że nie ma problemu z wyjeżdżaniem.

Pójdą też na zniesienie limitów przy udzielaniu świadczeń, tak żeby w końcu realnie zacząć likwidować kolejki do specjalistów, i na leki, żeby już żaden rodzic nie musiał błagać o pieniądze na leczenie swojego dziecka w Internecie, na Facebooku, błagać o to, żeby ludzie dorzucili się na operację, na kosztowne terapie. Całym sercem popieramy projekt Porozumienia Zawodów Medycznych dotyczący podniesienia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB, bo wiemy, że bez tego nie naprawimy systemu ochrony zdrowia. Na początku roku klub Lewicy złożył swój własny projekt, stopniowo podnoszący nakłady do 7,2% PKB i zmieniający ten haniebny sposób liczenia nakładów na ochronę zdrowia. Jeżeli naprawdę zależy wam na tym, żeby Polki i Polacy mieli dobrą ochronę zdrowia, przestańcie ich okłamywać, przyjmijcie projekt strony społecznej, przyjmijcie projekt Lewicy, podnieście nakłady na ochronę zdrowia, dofinansujcie ochronę zdrowia, tak jak robią to inne kraje Europy. Nie możemy być ciągle w ogonie. Musicie coś zrobić.

Wysoka Izbo! Opieka zdrowotna w Polsce choruje na brak pieniędzy. To pierwsza i najważniejsza przyczyna kolejnych dolegliwości systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Polska jest na szarym końcu pod względem wydatków na służbę zdrowia. Mówią o tym wyraźnie kolejne raporty Komisji Europejskiej i OECD. Eksperci mówią jasno: bez zwiększenia wydatków na system ochrony zdrowia nie zrobimy ani jednego kroku naprzód. Jak bardzo tych pieniędzy brakuje, widać choćby po wynikach finansowych szpitali za rok 2018. Strata netto w szpitalach marszałkowskich chociażby w województwie łódzkim to 71 mln zł. Ale to są szpitale, które mają relatywnie bogatego właściciela, który zapewnia wsparcie inwestycyjne, a tym samym amortyzację, która ratuje wyniki poszczególnych placówek. Niestety dużo gorzej jest w szpitalach powiatowych, które dzieli wręcz przepaść od placówek samorządu województwa. Problem, który musi zostać wreszcie zauważony, to pogłębiające się zadłużenie dużej części podmiotów leczniczych. W tym przypadku hasło dotyczące zrównoważonego budżetu państwa odbierane jest w wielu miejscach w Polsce jako ponury żart albo wręcz kpina z uczciwych ludzi. Nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że pacjenci muszą czekać na pewne świadczenie medyczne, zabiegi, a nawet porady lekarskie, ponieważ NFZ nie ma możliwości finansowania tych świadczeń na bieżąco. Kolejnym bardzo ważnym argumentem na to, że pieniędzy w systemie musi być więcej, jest fakt, że z roku na rok zwiększa się przepaść między wiedzą medyczną a tym, co państwo może zaoferować pacjentowi w ramach ubezpieczenia powszechnego. Tworzy się swego rodzaju opieka zdrowotna dwóch prędkości: dla tych, którzy mają pieniądze, i dla tych, którzy korzystają z ubezpieczenia powszechnego i leczenia w NFZ. Finanse realnie ograniczają dostęp pacjentów do nowoczesnych metod leczenia. W wielu przypadkach nasi lekarze mają wiedzę światową, a leczenie mogą zaoferować powiatowe. Sam doświadczyłem sytuacji, w której młody, zdolny chirurg odchodzi ze szpitala, ponieważ dyrekcji ani właściciela tego szpitala nie stać na zakup sprzętu i dostosowanie infrastruktury do możliwości, którymi dysponują wspomniany lekarz i jego zespół. Przykładem jest chociażby medycyna nuklearna, dostęp do badań PET-owskich i ograniczenia w stosowaniu nowych radiofarmaceutyków. To są jedynie zmiany prawne, których nikt w Polsce nie wprowadza, nie dokłada też pieniędzy. Kolejnym problemem jest zbyt mała liczba personelu medycznego w zakresie świadczeń publicznych, zwłaszcza lekarzy i pielęgniarek.

NIK, Najwyższa Izba Kontroli, co roku upomina się o większe nakłady na służbę zdrowia. Niedofinansowany system ochrony zdrowia jest barierą nie tylko dla pacjenta, ale również dla personelu, osób zarządzających placówką oraz właściciela tego podmiotu. Wielu ekspertów apeluje nie tylko o zwiększenie nakładów na zdrowie w Polsce, ale wręcz o skokowy wzrost środków przeznaczanych z budżetu państwa. Ceny idą w górę, a szpitale z tymi finansami żyją w permanentnym systemie pogotowia strajkowego. Czy będzie likwidowany, czy nie będzie? Po wyborach nie słyszałem dyskusji na ten temat. Niestety samorządy nie mają wpływu na wysokość finansowania. Nasuwa się pytanie, czy nie warto zastanowić się nad usamorządowieniem systemu opieki zdrowotnej, łącznie z finansami NFZ.

Głos zabierze teraz pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszystkie partie poza Konfederacją mają dokładnie to samo podejście do ochrony zdrowia: dosypać więcej pieniędzy. Jest to filozofia, która opiera się na założeniu, że jeśli dodamy więcej pieniędzy do systemu, to ten system zacznie lepiej działać. My jedyni uważamy, że to nie jest możliwe. Ten system jest od samego początku źle skonstruowany. Musimy pamiętać, że jest on dziedzictwem rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli na pewno nie może dobrze działać.

Musimy doprowadzić do gruntownej reformy systemowej. Inspiracji powinniśmy szukać chociażby w Czechach, gdzie umożliwiono pacjentom podwyższenie standardów zdrowotnych dzięki współpłaceniu. Inspiracji możemy szukać w Singapurze, gdzie pozwala się ludziom zarządzać własnymi składkami zdrowotnymi. Trzeba podkreślić, że wszystkie inne kluby opozycyjne mają podobne pomysły. Licytują się, kto da więcej. Jednocześnie partie te nie wskazały w sposób odpowiedzialny źródeł finansowania, którymi chciałyby pokryć rosnące wydatki w systemie ochrony zdrowia. Nie chcemy się licytować z innymi partiami, lecz chcemy wskazać, gdzie należy szukać pieniędzy na podwyższenie poziomu finansowania opieki zdrowotnej.

W tym kierunku, myślę, powinniśmy zmierzać, aby naprawdę zabezpieczyć nasz system zdrowotny. Mając w perspektywie czekający nas głęboki kryzys z uwagi na braki kadr medycznych, musimy jednak zastanowić się nad wsparciem personelu medycznego przez szerzej niż dotychczas zatrudnionych pracowników personelu pomocniczego, opiekunów medycznych i asystentów medycznych. Wprowadzenie takich elementów w systemie docelowo pozwoli łagodniej przetrwać okres kryzysu kadrowego, który nieubłaganie zbliża się, oraz trochę zracjonalizować poniesione koszty. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Drodzy Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej! Wysoka Izbo!

Wiecznie tylko reformujemy, reformujemy, a jest coraz gorzej. A więc proponowałbym, żebyśmy przestali reformować, posłuchali fachowców, dali środki finansowe i wymagali. Natomiast chciałbym powiedzieć, że dzisiaj cieszę się z tego, że debatujemy nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mimo że ten komitet inicjatywy złożył projekt w tamtej kadencji, w roku 2017. W dalszym ciągu cel, który został określony, jest do osiągnięcia i chciałbym w tej debacie zaapelować, abyśmy naprawdę pochylili się nad tym projektem.

A więc proszę was, siądźmy naprawdę ponadpartyjnie, merytorycznie do tego, aby ten problem rozwiązać. Bo jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Przecież na każdym kroku dyskutujemy o stanie służby zdrowia. Dzisiaj o godz. 9 rano w nowym budynku było posiedzenie zespołu ds. szpitali powiatowych. Szanowni państwo, jeden ze starostów powiedział: My już nie gasimy pożarów, my po prostu przygotowujemy wnioski o zamknięcie działalności, o likwidację. To jest totalne bankructwo. Oczywiście może część szpitali klinicznych, szpitale marszałków są w nieco lepszej kondycji, ale też nie do końca. Od wielu lat jestem przewodniczącym rady społecznej w jednym ze szpitali wojewódzkich i muszę powiedzieć, że mimo że ten szpital zawsze kończy rok z w miarę dobrym wynikiem, to ma niesamowite problemy.

To są wskaźniki, które bardzo wyraźnie mówią o tym, że powinniśmy pochylić się nad tym, aby jednak przyspieszyć nasze działania.

Myślę, że mielibyśmy o wiele lepszą sytuację w szpitalach. Mamy naprawdę wielu fachowców, którzy nam to wyraźnie wskazują.

Wtedy współpracowaliśmy także z organami powiatowymi, czyli ze starostami, którzy prowadzili szpitale powiatowe. Zróbmy w tych placówkach reformę, trochę tych pieniędzy jest.

Dlatego też prosiłbym, abyśmy naprawdę ponadpartyjnie tutaj, w parlamencie, usiedli i ten problem rozwiązali, abyśmy nie musieli omawiać następnych takich projektów. Przy tej okazji miałbym jeszcze jedną prośbę. Raz - wielkość tych środków, ale dwa - sposób podziału na poszczególne oddziały. Jestem z województwa opolskiego. Szkoda, że pani Porowska wyszła, bo ona dokładnie wie, jaka jest sytuacja.

Nie możemy doprosić się kontraktu. Panie Ministrze!

A potrzeby są. Dziękuję. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Jako pierwsza pani poseł Krystyna Skowrońska.

Wysoka Izbo! Polacy nie mogą czekać latami w niekończących się kolejkach na operacje ratujące zdrowie i życie. Dlatego konieczność podniesienia poziomu finansowego chyba nie podlega żadnej dyskusji. Jest na to prosta recepta, wystarczy po prostu nie kraść. Wystarczy nie rozdawać pieniędzy między sobie, swoim i między swoimi. Proszę państwa, trzymam w ręku dramatyczny w treści list kobiet z powiatu ustrzyckiego, którym poprzez likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego zabiera się prawo, równy dostęp do ochrony zdrowia i możliwość bezpiecznego porodu. Przypominam, że takie zasady są obwarowane zapisami w polskiej konstytucji. I, o dziwo, proszę państwa, dzieje się to pod rządami partii, która w niskiej demografii widzi bardzo wielkie zagrożenie, która pochyla się nad każdą poczętą istotą, a jednocześnie likwiduje oddziały położnicze. Dzisiaj nadszedł czas testu i prawdy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zdrowie Polaków to dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla rządu. To wyzwanie, którym rządzący powinni się zająć jak najszybciej. Dodam, iż Koalicja Obywatelska deklarowała skokowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Przedstawiciele rządu wielokrotnie obiecywali wzrost nakładów na ochronę zdrowia i wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów czy pielęgniarek. W związku z tym chciałam zapytać wnioskodawców: Czy rozmawiacie państwo na temat proponowanych przez państwa rozwiązań z przedstawicielami rządu? Jeśli tak, to jak wyglądają te rozmowy? Jakie było i jakie jest stanowisko rządu? Uważam, iż temat ochrony zdrowia powinien być przedmiotem ogólnopolskiej, szerokiej debaty, w tym okrągłego stołu, tak by jak najszybciej zająć się najbardziej palącymi, pilnymi sprawami w systemie ochrony zdrowia. Pani poseł Marta Wcisło, klub Koalicji Obywatelskiej. Pani poseł Magdalena Łośko, również klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Z roku na rok sytuacja publicznej służby zdrowia staje się coraz bardziej dramatyczna. Od kilku lat zadłużenie szpitali rośnie w rekordowym tempie. Sytuacji nie poprawiają braki kadrowe i brak troski rządu o pracowników wykonujących zawody medyczne. Są jednak środki na propagandę, i to wyjątkowo niskich lotów. Z jednej strony prezydent przyznający, że koszty życia rosną, a z drugiej premier mówiący, że brak podwyżek rekompensowany jest niższymi kosztami życia. Szkoda, że to wszystko odbywa się kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego naszych rodaków. Autorzy projektu słusznie zwracają uwagę na fakt, że środki przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych są niewystarczające. Dodatkowym wsparciem na opiekę zdrowotną mogą być przesunięcia środków, które rząd zamierza wydać na telewizję publiczną, kwoty 2 mld zł, i przeznaczenie ich na służbę zdrowia, na walkę z rakiem. Działanie to wesprze postulaty autorów ustawy. Czy zatem rząd podejmie się takiego działania? Środki są, tylko trzeba dokonać przesunięć, a w tym Prawo Sprawiedliwość jest już wprawione. Wysoki Sejmie! Polacy w badaniach opinii publicznej na pierwszym miejscu uważają, że najważniejszą dla nich kwestią jest sprawa naprawy służby zdrowia.

Na pewno jest tak, że jednym z tych elementów jest niewystarczające finansowanie służby zdrowia. Dlatego też ten projekt obywatelski wpisuje się w drogę poszukiwania rozwiązania, czyli pełniejszego finansowania potrzeb służby zdrowia, tak jak projekt Lewicy, o którym mówiła pani poseł Marcelina Zawisza. Skoro jest tak dobrze, jak mówiła pani poseł, to skąd dzisiaj ponad 14 mld zł zadłużenia szpitali powiatowych? Te powiaty, w których zadłużone szpitale funkcjonują, mają ograniczone funkcjonowanie i rozwój. Chciałem zapytać (Dzwonek) rząd, w jaki sposób będzie w tym roku udzielana pomoc tymże szpitalom. Pan poseł Michał Szczerba, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Było takie powiedzenie: rząd się wyżywi.

Mówiąc o poważnych sprawach, każdy przyzwoity Polak i każda przyzwoita Polka musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 2 mld z budżetu państwa zostaną wydane na Narodową Strategię Onkologiczną, na leczenie raka - 30 tys. Polek i Polaków przedwcześnie umiera na choroby nowotworowe - czy te 2 mld zł będą wydane na propagandę TVPiS? Kolejki do lekarzy stają się przeszłością” - pamiętacie państwo ten pasek. I kolejny: „Wynagrodzenia rosną jak na drożdżach” Pan poseł Ryszard Galla, poseł niezależny. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Chciałbym bardzo konkretnie zapytać o to, o czym na końcu powiedziałem, czyli o system kontraktowania usług. Czy państwo przewidujecie może pracę, powrót do bardziej sprawdzonego systemu kasowego? Czy myślicie o tym, aby jednak zmienić ten algorytm podziału środków na poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia? Nie ukrywam, że w przypadku tych mniejszych województw jest to wielce niesprawiedliwe. Podział tych środków powoduje, że bardzo często w jednym regionie można pozwolić sobie na wiele, a w tym regionie, który ma mniej środków, jest o wiele, wiele trudniej. Pan poseł Marek Hok, klub Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Panie ministrze, mówicie państwo o historycznym co roku podwyższaniu nakładów na ochronę zdrowia. To wynika, tak jak powiedziałem, oczywiście z zwiększonej składki, ze zwiększonych wynagrodzeń.

Wysoka Izbo! Mam pytanie dotyczące leczenia za pomocą medycyny nuklearnej, która w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwija i jest niezwykle pomocna pacjentom. Czy Ministerstwo Zdrowia wreszcie zareaguje na płynące wnioski o rozszerzenie listy refundacji badań ze wskazaniami PET? Chodzi przede wszystkim o nowe rodzaje radiofarmaceutyków i liczbę badań, które należałoby zwiększyć o ok. 30%, jak wskazują eksperci z tej dziedziny. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Paszyk, klub Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj chciałbym skorzystać z okazji, którą stwarza ta debata, by zapytać przedstawiciela rządu, kiedy rozpocznie się realizacja zapisów paktu dla zdrowia. Przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz przed wyborami zaproponował pakt obejmujący wzrost nakładów na służbę zdrowia do minimum 6,8% PKB, podniesienie pensji wszystkim pracownikom służby zdrowia o 30% oraz upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki. Wydaje się, że są to niezbędne działania do tego, żeby postawić na nogi służbę zdrowia.

Dziękuję bardzo. Wysoki Sejmie! Marszałek Sejmu zwołała Konwent Seniorów i jestem zmuszony na chwilę przerwać obrady, ale mamy jeszcze parę minut. No to ogłaszam 15-minutową przerwę.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przewodniczący, wnioskodawca mówił o tym, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to wszystko, co się dzieje w służbie zdrowia, to są pewne bajeczki i słychać dyskusję ze strony rządowej o tym, jak liczymy nakłady, a nie o pacjencie, nie o dostępności. Żeby tego nie rozwijać, nie ciągnąć tych faktów jakoś wyjątkowo długo wstecz, to podam krótkie fakty tylko z roku 2020, który dopiero się zaczął. Wiele razy, również na tej sali, mówiliśmy o psychiatrii dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży, o jej niedofinansowaniu, o braku nakładów w tym zakresie.

To nie bajeczki, to fakt. To fakt i te środki, twarde środki, zostaną skierowane do tego bardzo wrażliwego obszaru - psychiatrii dziecięcej. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. To również nie jest kolejna bajeczka, to nie jest mrzonka i pierwszy od wielu lat będziemy podnosić wyceny w AOS: w tym roku o prawie 20%, od 1 stycznia 2021 r. o kolejne 10, a to wiąże się właśnie z bezlimitowością świadczeń i zniesieniem limitów do neurologa, ortopedy, kardiologa, endokrynologa. Na to chcemy przeznaczyć ok. 300 mln zł. To również nie jest bajeczka, to fakt. Dopiero co na początku lutego, 4 lutego, w Światowym Dniu Walki z Rakiem uchwalona została przez Radę Ministrów Narodowa Strategia Onkologiczna.

To długo oczekiwana inwestycja konsolidująca trzy szpitale kliniczne, które funkcjonowały w bardzo trudnych warunkach infrastrukturalnych.

Kolejny fakt. Zwiększenie o ponad 136 mln środków na kształcenie na uczelniach wyższych, zwiększenie limitów na studia. Kolejny fakt. Z tej mównicy wielokrotnie dzisiaj padała kwestia braku kadr. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę.

To nie jest znowu bajeczka, to jest fakt. I ostatni już fakt również wynikający z tej samej ustawy budżetowej.

To nie są bajeczki. To są fakty również spowodowane właśnie tym, co wydarzyło się w roku 2017 i później w roku 2018, czyli właśnie najpierw przygotowaniem przez rząd, a potem uchwaleniem przez Sejm tzw. ustawy 6%, czyli ustawy, która ma przybliżać nas do tego, o czym była mowa na tej sali. Ma nas przybliżać, czyli zwiększać rzeczywiście finansowanie służby zdrowia poprzez ten stabilny - rozłożony wprawdzie na kilka lat - wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Patrzymy na to realnie i zdajemy sobie sprawę, że te wzrosty oczywiście mogły być większe. Ja w szczególności jako przedstawiciel resortu zdrowia pewnie nawet bym bardzo chciał, żeby one były znacznie wyższe. Ale ta dyskusja musi odbywać się też na forum rządu, na forum rozmowy z ministrem finansów, na forum możliwości, które dzisiaj mamy. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Kamińskiemu za wystąpienie, w którym wskazywał na mówienie o czymś, co jest realne, czyli pokazywanie pewnych projektów ustaw. Mówię tu o projekcie obywatelskim, ale myślę, że za chwilę Sejm pochyli się nad projektem bardzo podobnej ustawy Lewicy, podobnej ustawy PSL-u, gdzie rzeczywiście będziemy rozmawiać o zwiększeniu nakładów na zdrowie. Ponawiam więc tak naprawdę pytanie pana posła Kamińskiego. Będę wdzięczny - myślę, że ja, a nawet bardziej minister finansów - jeżeli pokażecie państwo źródło finansowania tych ustaw. Telewizja padała z tej mównicy, więc ja może uzmysłowię panu i Wysokiej Izbie, gdzie są nakłady na telewizję, a gdzie są te, o których mówimy dzisiaj, przy tej ustawie. Jeżeli tę ustawę byśmy przyjęli, Sejm by ją przyjął, to nakłady na ochronę zdrowia trzeba byłoby zwiększyć automatycznie już teraz, już w roku 2020, o prawie 30 mld zł. Jeżeli przyjęlibyśmy ustawę Lewicy, ustawę PSL-u, te wzrosty byłyby jeszcze większe. Nie możemy więc dzisiaj porównywać ustawy, o której rozmawiamy, ustawy, o której pewnie będziemy rozmawiać - chodzi o dojście do kolejnych zwiększonych procentów PKB - z tymi 2 mld, które idą na telewizję. Bo to jest w ogóle dyskusja o całkiem innym poziomie kwot i całkiem innym poziomie zaangażowania budżetu państwa.

To jest fakt, to nie jest coś mitycznego, to nie jest coś, czego nie realizujemy. Co więcej - również z tej mównicy to padało - jest to wynik dobrej koniunktury, jest to wynik tego, że składki rosną i Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje większymi środkami. To jest fakt, ja z tym faktem nie polemizuję. Ale też proszę zwrócić uwagę na to, czego wcześniej nigdy nie było - na rok 2017, na rok 2018, na rok 2019, czyli środki skierowane z budżetu państwa właśnie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczerze mówiąc, słucham czy chociażby ostatnio czytam bardzo ciekawy wywiad z przewodniczącą Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, która mówi: Wreszcie zaczęto nas szanować, wreszcie nie jesteśmy na granicy wynagrodzenia minimalnego, wreszcie ktoś nas dostrzegł i te wynagrodzenia zwiększył. Słucham przedstawicieli okręgowych izb lekarskich, Naczelnej Izby Lekarskiej - mówią jednoznacznie, że już nie chcą i nie postulują zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, że nie taki jest cel ich działań. Ratownicy - kolejna grupa.

Pani poseł Zawisza mówiła również o pewnym strachu przed podniesieniem podatków, a słyszę z drugiej strony coś, co stoi z tym całkiem w sprzeczności.

Poseł Klimczak mówił o tym, że potrzebny jest skokowy wzrost. Właśnie ten skokowy wzrost następuje. Ciężko, wydaje mi się, szanownym państwu z tym dyskutować.

Przyjmiemy jako rząd, przyjmiemy jako Sejm 6,8% PKB, minie pół roku, pojawi się postulat 7,5%. Pewnie jako minister zdrowia bym był do tego chętny.

Poseł Hok pytał o bezlimity, o to, czy świadczenia bezlimitowe w tych czterech dziedzinach zostały zabezpieczone finansowo. Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje środkami na to. Tak jak mówiłem, chcemy przeznaczyć na to ponad 300 mln zł i te środki będą zagwarantowane w planie Narodowego Funduszu Zdrowia. O Telewizji Polskiej już mówiłem i odniesieniu tych 2 mld do tego, jakie są oczekiwania wynikające z tej ustawy. Bardzo ciekawe i szczegółowe pytanie zadał poseł Klimczak dotyczące medycyny nuklearnej.

Jak rozumiem - tak rozumieliśmy zresztą intencje tego paktu - był to pakt, który miał obowiązywać przez następną kadencję. Był to pakt złożony i podpisany przed obecną kadencją Sejmu, więc wydaje mi się, że jeszcze prawie 4 lata przed nami, żeby ten pakt dla zdrowia móc spokojnie realizować. Szanowni Państwo! Rzeczywiście, potrzebny nam jest wzrost nakładów na zdrowie i nie będę z tym polemizował. Absolutnie się z tym zgadzam. Bardzo bym chciał pewnie nawet, żeby ten wzrost był szybszy niż dzisiejszy, zagwarantowany ustawą, 6-procentowy. Ale może zwróćmy uwagę na to, że w kilkudziesięcioletniej już historii Polski po 1989 r. i po kolejnych reformach takiej ustawy nie było, ustawy wiążącej nakłady na ochronę zdrowia z pewnym poziomem rozwoju czy dobrobytu państwa nie było. Ta ustawa funkcjonuje od roku 2017.

Myślę, że owocna będzie ona wtedy, jeśli zastanowimy się wspólnie merytorycznie nad źródłami finansowania tego wzrostu. A szczęśliwie dzisiaj, patrząc na ostatnie 2 lata, tak właśnie jest. Dziękuję. Teraz głos ma przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pan Tomasz Dybek.

Koleżanki i Koledzy!

Panie Ministrze! Faktem jest, że ta ustawa przeleżała 3 lata w Sejmie. Faktem jest, że ustawa poprzednia, pod którą było ćwierć miliona podpisów, przeleżała 3 lata w Sejmie.

Pracują w dwóch, żeby normalnie funkcjonować w Polsce, to jest fakt.

Tak samo poprzednia ustawa.

Jaki jest dostęp do medyków? Trzeba sobie zadać pytanie, po prawej stronie, po lewej: Co trzeba zrobić, żeby to się zmieniło? Mam na koniec taką propozycję. Państwo stalibyście w tych kolejkach i wtedy byście to zrozumieli.

Dziękuję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawarty w druku nr 37, do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jedna z komisji nie dostarczyła jeszcze sprawozdania, dlatego ogłaszam przerwę do głosowań, czyli do godz. 19.30.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekty uchwał: - w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, druk nr 256, - w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci, druk nr 259. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych projektów. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, - o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, - o ochronie roślin przed agrofagami. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 235, 225 i 226. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, - o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, - o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, - o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw, - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 232, 224, 228, 230, 229, 237, 250 i 254. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (druk nr 256) Proszę państwa posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Dokładnie 80 lat temu rozpoczął się dramat mieszkańców wschodnich Kresów Rzeczypospolitej zajętych przez Sowietów na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow. Pierwsze deportacje objęły osadników wojskowych, leśników, kolejarzy oraz urzędników państwowych. Wraz z całymi rodzinami stawali się oni ofiarami zbrodniczego systemu. Bezkresne stepy i tajgi obwodów irkuckiego, omskiego, nowosybirskiego czy archangielskiego miały być ich domem na lata zsyłki. Dla wielu stały się również grobem.

W ich efekcie na zsyłkę trafiło około miliona Polaków, ale również wielu Ukraińców, Białorusinów i Żydów, obywateli Rzeczypospolitej. Życie na zesłaniu straciło prawie 200 tys. spośród nich. Wielu z tych, którzy przeżyli, nie dostało szansy powrotu do Ojczyzny. Ich żywot dokonał się na obczyźnie, a ich potomkowie żyją tam do dziś. Deportacje naszych rodaków na Wschód, w tym na Sybir były niezwykle bolesnym i tragicznym doświadczeniem dla całego Narodu. Komunistyczny reżim zamierzał dokonać eksterminacji elit politycznych, gospodarczych i intelektualnych oraz rozbić strukturę społeczną Polski. Pomimo skali i charakteru podjętych działań nie udało się zniszczyć ducha w naszym Narodzie. Nie ma słów, które by w pełni oddawały dramat naszych rodaków. Żyli i pracowali ze świadomością, że niewielu spośród nich może być dany powrót do domów. Pamięć o zesłaniach niech będzie przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Niech stanowią one dowód tego, do czego zdolny może być człowiek. Mając w pamięci tragiczny los i bohaterską postawę setek tysięcy deportowanych, w 80. rocznicę pierwszych deportacji Polaków na Wschód Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim zesłańcom oraz ich rodzinom” Proszę o przyjęcie uchwały przez aklamację. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci (druk nr 259) Proszę państwa posłów ponownie o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci. W 2020 roku obchodzimy 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego, zmarłego na emigracji, redaktora, wydawcy, krytyka literackiego i dziennikarza. Od 1920 roku Mieczysław Grydzewski wydawał miesięcznik 'Skamander', wokół którego skupiła się grupa młodych poetów, kojarzona do dzisiaj z tytułem tego pisma. W 1924 roku rozpoczął wydawanie 'Wiadomości Literackich' - jednego z najważniejszych czasopism Polski międzywojennej - które przetrwały, w różnych wcieleniach, niemal 60 lat. Ostatni przedwojenny numer 'Wiadomości Literackich' ukazał się z datą 3 września 1939 roku. Mieczysław Grydzewski opuścił Polskę i udał się na emigrację, z której nigdy nie wrócił. Wróciły jednak 'Wiadomości...' pod jego redakcją: najpierw w Paryżu jako 'Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie', a później w Londynie jako 'Wiadomości' Przez kilkadziesiąt lat 'Wiadomości' redagowane na uchodźstwie przez Grydzewskiego, następnie przez Michała Chmielowca i aż do wiosny 1981 roku przez Stefanię Kossowską, były najważniejszym ośrodkiem integrującym polskich emigracyjnych poetów i pisarzy. Mieczysław Grydzewski i skupione wokół niego środowisko 'Wiadomości' pozostaje symbolem nieprzejednanej postawy wobec Rosji Sowieckiej i komunistycznych władz oraz niezłomnego przywiązania do idei niepodległości Polski. Życie i dzieło Mieczysława Grydzewskiego przypominają o tym, o czym wciąż zbyt łatwo zapominamy: że życie twórcze i duchowe społeczeństwa nie opiera się wyłącznie na indywidualnym wysiłku jednostek. Literatura powstaje w procesie pracy zbiorowej: od redaktorki, tłumacza, księgowej po drukarza. Nie ma literatury bez życia literackiego i nie ma kultury bez instytucji kultury, które muszą być dla twórców oparciem. W 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć jego pamięci i dziełu” Bardzo proszę, żebyśmy przyjęli projekt uchwały przez aklamację. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci. Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL-Kukiz15. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, druk nr 234. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o to sprawozdanie. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, druki nr 211 i 234, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 201-A. Proszę pana posła Jarosława Krajewskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu wniosków i poprawek na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. wnoszą o odrzucenie dwóch wniosków w sprawie odrzucenia projektu ustawy w całości oraz wnioskują o przyjęcie ośmiu poprawek oraz odrzucenie dziewięciu poprawek. Dziękuję bardzo. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 201. Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość propozycji komisji. Przepraszam, pani poseł, nie mam zgłoszenia. Przepraszam.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Jeszcze nikt w Polsce nie dopuścił się takiej grabieży środków obywateli.

wy zamierzacie po prostu roztrwonić w 1 rok. Obywatele odkładali to, by dożyć godnej starości. A wy roztrwonicie to w 1 rok. Niech wam to dźwięczy w uszach. Dodatkowo ukrywacie, że ci, którzy zabiorą środki na IKE, po prostu w przyszłości będą mieli niższe emerytury wypłacane z ZUS. Od początku pracy nad tą ustawą proszę rząd, żeby przedstawił raport (Dzwonek) w tej sprawie.

Jest jeszcze czas. Ale zgłosiliśmy poprawki, które robią ją strawniejszą dla ubezpieczonych.

Dlaczego ZUS nie może być pośrednikiem między przekazaniem deklaracji do otwartych funduszy emerytalnych i ułatwić ubezpieczonym tę operację? Dlaczego to jest niemożliwe? Zwykle ludzie i tak wybierają opcję domyślną, czyli tę, którą proponuje państwo, więc nie ma się czego tak bardzo bać.

Pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. Wysoka Izbo! Ten projekt, tak jak mówiła pani posłanka Fedak, jest głęboko szkodliwy. Wprowadzenie OFE wygenerowało 330 mld dodatkowego długu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale przynajmniej te pieniądze nadal były publiczne i były zarządzane tylko przez prywatne instytucje. W tej chwili oddajecie 150 mld pozostałych jeszcze w OFE w zupełnie pełne prywatne zarządzanie instytucji finansowych bez żadnej kontroli. Bez absolutnie żadnej kontroli. Nie mamy żadnej gwarancji, że kiedykolwiek zobaczymy te emerytury z IKE, ponieważ nie zagwarantowaliście państwo w tej ustawie żadnych mechanizmów kontroli nad tym, w co dokładnie będą inwestowane te fundusze. Już teraz mogę państwa zapewnić, że banki i instytucje finansowe nie działają w interesie emerytów, nie działają w interesie stabilności państwa ani systemu emerytalnego. Działają we własnym interesie. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Rozumiem, że są różnice dotyczące tego, gdzie to zostało przelane, czy obligacje zostały umorzone, czy po prostu w formie podatku to zostało zagrabione, ale prawda jest taka, że prywatne konta obywateli zostały uszczuplone, wtedy o 150 mld, teraz o 24 mld. Powinni państwo być z tego dumni. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. W 1. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują ustawie nadać inny tytuł.

Panie Premierze! Panie Pośle! Proszę nie bawić się w rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

To, co miało kiedyś miejsce, było przepisaniem 1 do 1 na subkoncie w ZUS pieniędzy odłożonych przez obywateli. Nie popierałam tego, koledzy i koleżanki z klubu o tym wiedzą, ale różnica jest ogromna, bo nikt wtedy nie zmniejszył oszczędności odłożonych na OFE, przepisując je do ZUS 1 do 1. Co więcej, środki te były dziedziczone. To jest druga podstawowa różnica.

Dziękuję, pani marszałek, za możliwość wypowiedzenia się z mównicy. Zadania pytania, panie pośle. Porównanie Koalicji Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości to nie jest komplement, to jest obelga z moich ust, naprawdę. A co do tej zmiany nazwy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Konsekwencją ich przyjęcia będzie bezprzedmiotowość poprawki 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. W 3. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie art. 59. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją jej przyjęcia będzie bezprzedmiotowość poprawki 4. Proszę.

Bardzo dziękuję.

Ustawa wymusza gromadzenie kapitału na emerytury właśnie w spółkach, nawet w 90%, w tym także w spółkach Skarbu Państwa nieudolnie zarządzanych przez rząd premiera Morawieckiego. Z powodu tego nieudolnego zarządzania Polacy stracą oszczędności na emerytury. Panie premierze Morawiecki, czy zwrócicie Polakom te oszczędności, które stracą w wyniku waszego nieudolnego zarządzania, żeby nie cierpieli głodu, kiedy przejdą na emeryturę? Mówicie, że kochacie polskie rodziny. Panie premierze, dlaczego wydziedziczacie dzieci?

Czy to jest troska o polskie dzieci? Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 4. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę w art. 59 ust. 6 pkt 10. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 4. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 11. poprawce do art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wnioskodawcy proponują nowe brzmienie ust. 5. Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Bardzo proszę.

Proszę o spokój, proszę państwa. Rozumiem, że państwo posłowie PiS-u chcielibyście tej dyskusji uniknąć. Ale sprawa jest tak naprawdę bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy państwo wycofuje się z obietnic emerytalnych i po raz pierwszy państwo prywatyzuje odpowiedzialność za przyszłe emerytury.

Druga sprawa, która jest związana z tą ustawą, to jest tak naprawdę wydziedziczenie Polaków. Jeżeli ktoś wybierze ZUS, to środki, które dotychczas były w OFE, nie będą mogły być dziedziczone. Nie będą mogły być dziedziczone również nowo opłacane składki, bo trafią na konto, a nie trafią gdzie? Na indywidualne subkonto. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Proszę. Panie i Panowie Posłowie! Pewnie na koniec debaty, na koniec głosowania przy tej ustawie wyjdzie minister Buda i powie, że prywatyzujecie środki emerytalne. Ale nie powie, bo ukrywacie to cały czas, że Polacy nie dostaną 100% środków na konto w IKE, tylko dostaną 85%. Czyli jeżeli ktoś ma na koncie w OFE 50 tys. zł, to wy uznajecie, że za przelanie pieniędzy z konta na konto macie prawo pobrać 15%, czyli 7,5 tys. od tych 50 tys. Jeszcze nikt w Polsce nie pobierał takich opłat manipulacyjnych za przelanie środków z konta na konto.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Proszę. Panie Premierze! 15% twardego majątku Polaków, pieniędzy ulokowanych na giełdzie, w akcjach, w obligacjach korporacyjnych i innych papierach skarbowych czy też właśnie bardziej agresywnie inwestowanych, to jeszcze zabieracie tak naprawdę najbezpieczniejszą część portfela OFE i zmuszacie obywateli, którzy zabiorą swoje środki na IKE, do bardziej agresywnej polityki inwestycyjnej. Dzisiaj wymóg jest taki, żeby środki w OFE w siedemdziesięciu paru procentach były inwestowane w akcje, a wy chcecie zmusić Polaków, by w pierwszych latach zaostrzyli tę politykę inwestycyjną i zwiększyli środki inwestowane w akcje na giełdzie do ponad 90%. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość 5. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. W 6. wniosku mniejszości do art. 76 wnioskodawcy proponują inny termin wejścia w życie ustawy. Proszę. Wysoka Izbo! My tu dyskutujemy o szczegółach, robimy poprawki do tego systemu, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten system nie polega na tym, że odkładamy wypracowane pieniądze na emeryturę i później, jak przejdziemy na emeryturę, to z nich korzystamy, tylko polega na tym, że osoby obecnie pracujące opłacają emerytury obecnych emerytów. To oznacza, że ten system może działać tylko wtedy - tylko przy tym założeniu - kiedy rodzi się dokładnie tyle samo dzieci co wcześniej. Ten system ma błąd genetyczny, który prowadzi nas do katastrofy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Przed przystąpieniem do głosowania nad całością projektu ustawy mamy pytania. Proszę. Panie i Panowie Posłowie! Istotnie, polski system emerytalny wymaga zmian, zwłaszcza po jego dewastacji, którą robicie przez ostatnie 4 lata. Dzisiaj stopa zastąpienia, czyli wysokość emerytury dla mojego pokolenia, moich rówieśników, to 20% minimalnego wynagrodzenia, a minimalne wynagrodzenie na koniec życia, bo o tym mówię, jest zazwyczaj niższe niż wynagrodzenie przeciętne. Skazujecie moje pokolenie i moich następców, naszych następców na głodowe emerytury. jeszcze niższe niż te emerytury, które emeryci odbierają dziś. Wy patrzycie na system emerytalny tylko z jednego punktu widzenia - ile z niego dla siebie, na własne obietnice wyborcze i na przejadanie w ministerstwach źle zarządzanych przez waszych ministrów, możecie dziś wydrenować. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Jeden z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości powiedział z dumą: prywatyzujemy ten system. Nie macie z czego być dumni. Prywatyzacja systemu emerytalnego nigdzie na świecie się nie sprawdziła. Szczerze mówiąc, dziwię się, kiedy patrzę na twarze kilku państwowców w ławach Prawa i Sprawiedliwości - patrzę na jedną z nich - że podnoszą rękę za czymś tak szkodliwym.

Dziękuję.

Wysoka Izbo! To, co najbardziej być może szokuje w tych wszystkich pseudoreformach.

Jedyne, co wam pozostało w tej kadencji Sejmu, to robienie jakiejś kosmetyki, żeby to ratować i pudrować roszady kadrowe, które były istotą waszej władzy przez ostatnie 4 lata. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pana Waldemara Budę. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

My dzisiaj tą ustawą przesądzamy, że są to środki prywatne Polaków. Już 27 listopada te środki będą przelane na indywidualne konta Polaków. Co to oznacza?

Jest zapis, art. 50 ust. 1 pkt 2, który mówi o tym, że są to środki prywatne i nie podlegają transferowi do budżetu państwa. Polacy mają możliwość zdecydowania.

Jest różnica?

Dzisiaj mówicie, że bronicie systemu emerytalnego? To nieprawda. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 201, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? To podejdę zaraz osobiście i sprawdzę. Działa?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 169-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury w dniu dzisiejszym rozpatrzyła poprawki złożone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie

Dotyczy to klauzulowania materiałów, które geodeta w wyniku wykonanej pracy przekazuje zleceniodawcy. Ta procedura nie jest nowością, funkcjonowała od lat.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 169. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Nie mam zgłoszenia, panie pośle. Zgłosił się pan? Ale, panie pośle, na przyszłość proszę zapisać się wcześniej, bo ja nie mam zgłoszenia, że pan się zgłasza do pytania. Proszę bardzo. Państwo z PiS-u obiecali deregulację, zlikwidowanie weryfikacji, ale znowu okazuje się, że to jest zamiana siekierki na kijek, a raczej kijka na siekierkę, ponieważ to klauzulowanie, które się tutaj wprowadza, jest w rzeczywistości bardziej dotkliwe dla przedsiębiorców niż dotychczasowa weryfikacja. Dolegliwość polega przede wszystkim na tym, że w zakład rozliczeń między geodetą a urzędem bierzemy teraz inwestora, który nie będzie mógł rozpocząć pracy bez czerwonej pieczątki z urzędu, więc tym samym główna patologia, jaka toczy polską geodezję, czyli to, że urzędnicy w sposób nieuczciwy konkurują z przedsiębiorcami, stanie się jeszcze głębsza.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Z poprawką tą łączy się poprawka 20. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czy liberalizacja przypisów powinna oznaczać wprowadzenie nowych procedur i nowych obowiązków dla przedsiębiorców i inwestorów? Czy państwo powinno nakładać na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie świadczeń różnego rodzaju usług, czy też powinno to komunikować i finansować z podatków? Czy ustawa powinna wprowadzać drakońskie podwyżki, czy też regulować to w taki sposób, żeby one odpowiadały kosztom?

Trzeba zachować proporcje. Składamy poprawki, które mają za zadanie wprowadzenie takich proporcji i upłynnienie procesu inwestycji. Myślę, że każdy, komu zależy na tym, żeby biznes działał, gospodarka funkcjonowała, a z drugiej strony odpowiednie rejestry miały odpowiedni poziom (Dzwonek), zagłosuje za tymi poprawkami. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2. i 20., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 3. i 4., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 8. Proszę. W tym punkcie prosimy o zniesienie absurdalnego ograniczenia przy zgłaszaniu pracy na tylko rok do przodu.

Wszystko to po to, żeby dostosować prawo do programu komputerowego, który wyprodukowała firma, której współwłaścicielem był główny geodeta kraju. Po prostu przycinamy rękę pod zegarek w ten sposób.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 11. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Proszę. W tym punkcie znowu szczycimy się zniesieniem licencji, a de facto wprowadzamy taką quasi-licencję, która spowoduje, w największym uproszczeniu, że w pewnych sytuacjach geodeta będzie musiał płacić urzędowi za swoje własne dane, żeby je z powrotem wykorzystać. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 12. i 25., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 15. Proszę. Ta poprawka znosi kolejną niedogodność, jaką jest sprawdzenie dodatkowych kryteriów w postaci spójności danych z dotychczasowymi danymi w systemie. Nie określono w żaden sposób kryteriów tej spójności, co spowoduje prawdopodobnie liczne nieporozumienia, kontrowersje, spory sądowe i znowu opóźni procesy inwestycyjne. Zachodzi po raz kolejny podejrzenie, że chodzi o spójność danych z programem komputerowym ePODGiK, który ma problemy z przyjmowaniem danych w najbardziej powszechnym formacie. W związku z tym prawdopodobnie geodeci będą musieli zakupić program byłej firmy pana głównego geodety. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 17. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. W tej poprawce proponujemy wprowadzenie zasady milczącej zgody w sytuacji, kiedy organ nie wyrobi się w terminie z weryfikacją. Wiem, że tę poprawkę w głębi serca popiera pani sprawozdawca Anna Paluch, tylko pan główny geodeta nie pozwolił jej na sali zagłosować za tą poprawką, ale dzisiaj go chyba nie ma. Proszę. Proszę państwa, jeżeli rzeczywiście wprowadziłoby się zasadę milczącej zgody, tzn. zobowiązanie dla organu, żeby przyjął wadliwy materiał, będzie to rzutowało na jakość mapy i stracą na tym wszyscy: inwestorzy, wykonawcy, ten, który zrobił złą robotę, i wszyscy inni. W ostatecznym rozrachunku doprowadziłoby to do pogorszenia jakości zasobów, a pomimo że kilka lat temu wydano bardzo pokaźne pieniądze na informatyzację zasobu geodezyjnego, to treść tego zasobu nadal pozostawia wiele do życzenia.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Pan poseł Dobromir Sośnierz. Proszę bardzo. Ta poprawka wprowadza instytucję uzgodnienia terminów, w sytuacji kiedy geodeta sam przyznaje, że popełnił błąd i musi coś poprawić, żeby mógł uzgodnić z organem termin wprowadzenia tej poprawki. Takie przyjazne państwo po prostu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił.

Pan poseł Mirosław Suchoń.

Dziękuję bardzo. Panie Premierze! Wysoka Izbo!

To oznacza drakońskie podwyżki. Pytanie do rządu. Czy to jest sposób sprawowania władzy, że każdą opłatę, każdy podatek, który istnieje, podwyższacie, a jeżeli brakuje wam tych podatków i opłat do podwyższenia, to wprowadzacie nowe?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 27. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują inne brzmienie ust. 4. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Proszę. To jest podobna poprawka.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 28. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują nie wprowadzać zmian w tabeli nr 6. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 29. Proszę.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 28. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 29. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują nie wprowadzać zmiany w kolumnie trzeciej tabeli nr 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 29. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Proszę. W tym miejscu podnosimy znowu współczynniki, w niektórych przypadkach nawet kilkunastokrotnie, bo współczynnik, który wynosił do tej pory 0,02, będzie wynosił 0,3, a więc to jest kilkunastokrotna podwyżka. Miejmy litość dla naszych geodetów, przedsiębiorców. Proszę o poparcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 30. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 33. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Proszę. To już po raz ostatni. Wprowadzamy tutaj zryczałtowaną opłatę.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 35. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 36. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Pan poseł Zbigniew Girzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Wzruszony troską pana posła Sośniarza. Przepraszam bardzo pana posła. o to, aby deregulować tak bardzo usługi geodezyjne, a jednocześnie znając doskonale troskę pani poseł Anny Paluch, która z wykształcenia i kiedyś z zawodu jest wytrawnym geodetą, chciałbym zadać pytanie pani poseł sprawozdawcy, powołując się na pewien przykład historii, choć nieco związany bardziej z fikcją, ale pokazującą pewną rzeczywistość. Otóż przed wojną także funkcjonowało prawo geodezyjne. Ono nie było tak bardzo doregulowane jak obecnie i w odległej miejscowości na Kresach, Krużewnikach, był konflikt, który państwo znacie doskonale z filmu, o miedzę, który Kargul z Pawlakiem zaledwie o dwa palce tej miedzy musieli rozstrzygać w sposób powszechnie wiadomy. co skończyło się emigracją jednego z nich. Pani poseł, pytanie. Dziękuję, panie pośle. Pytanie zada pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Wysoka Izbo! Geodeta musi być jednocześnie dobrym prawnikiem, musi być specjalistą od lokalnego urzędu ze znajomościami, z niesamowitą umiejętnością lawirowania w absurdach tej biurokracji, absurdalnych decyzjach urzędników i przez to trwoni on co najmniej połowę swojego czasu, który mógłby przeznaczyć na zlecenia, właśnie na tę biurokrację. Już nie mówię o tych absurdalnych opłatach za każdym razem, np. opłacie za uzyskanie z urzędu informacji, które musi uzyskać, które sam do tego urzędu wstawił. My głosowaliśmy za państwa poprawkami, które były dobre. Wy zagłosowaliście przeciwko wszystkim naszym poprawkom. I wy mówicie, że ktoś tu jest totalną opozycją? Dziękuję, panie pośle.

Wysoka Izbo! Wczoraj pytałem z tej mównicy, czy faktycznie ta zmiana ustawy ma służyć społeczeństwu, ma przyspieszyć, ułatwić procedowanie. Nie dowiedziałem się.